są obarczone znacznie większym ryzykiem.

Dyskusja na posiedzeniu komisji finansów koncentrowała się właściwie wokół kilku spraw. Myślę, że najistotniejszą było zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i wyznaczenie górnych limitów wydatków ze strony Skarbu Państwa.

W ustawie wprowadzono również szereg poprawek legislacyjnych i redakcyjnych, m.in. z pierwotnego projektu skreślono wyraz „dla”, czyli zostało: o wsparciu rynku ubezpieczeń społecznych.

Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy przedstawionego w sprawozdaniu z przyjętymi poprawkami. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Jarosław Krajewski w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, druki nr 431 i 482. Na początku zacząłbym od tego, że przed chwilą minęło 110 dni od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. W trakcie tych 110 dni mieliśmy bardzo wymierną pomoc dla polskich przedsiębiorców i dla polskich pracowników - w wysokości ponad 115 mld zł. Mówimy o bezprecedensowym wsparciu ze strony rządu w czasach kryzysu światowego wywołanego przez koronawirusa. Mówimy w tym przypadku o skutecznych działaniach, które mają na celu ochronę ponad 5 mln miejsc pracy w naszym kraju. Projekt ustawy, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest dodatkowym elementem wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Z uwagi na sytuację związaną z wpływem COVID-19 na gospodarkę zakłady ubezpieczeń mogą znacznie obniżyć limity lub zlikwidować w ogóle ekspozycję na ryzyko w odniesieniu do wybranych branż, kontrahentów lub rynków. Taki scenariusz byłby zdecydowanie negatywny z punktu widzenia polskiej gospodarki, ponieważ polscy przedsiębiorcy mieliby ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, w wyniku czego obniżeniu uległyby obroty handlowe oraz potrzebna byłaby dodatkowa płynność w sytuacji ograniczenia możliwości sprzedaży w kredycie kupieckim. Projekt ustawy ma na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W tym celu rząd proponuje umożliwienie zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reasekurowanie części ryzyka przez Skarb Państwa. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Zgodnie z ustawą reasekuracja będzie realizowana w ramach programu pomocowego, który będzie mogła przyjąć Rada Ministrów. Program będzie wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej z uwagi na przewidywaną w nim pomoc publiczną. Pomoc zakładom ubezpieczeń realizowana będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a danym zakładem ubezpieczeń. To projektowane rozwiązanie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która umożliwia pełnienie przez Skarb Państwa roli reasekuratora tzw. ostatniej szansy w przypadku ubezpieczeń należności handlowych. Należy dodać, że w chwili obecnej w co najmniej kilku państwach Unii Europejskiej trwają intensywne prace nad podobnymi rozwiązaniami. Warto przypomnieć, że do tej pory Komisja Europejska zaakceptowała podobne programy pomocowe m.in. w Niemczech i we Francji. Ten projekt ustawy przewiduje rozwiązania zbliżone do tych, które zostały już przyjęte i zaakceptowane przez Komisję Europejską w Niemczech. Chodzi o program wsparcia bazujący na reasekuracji i gwarantowaniu ryzyk zakładom ubezpieczeń. Ta ustawa powinna przynieść pozytywne efekty w postaci ograniczenia ryzyka spadku transakcji handlowych realizowanych przez polskich przedsiębiorców, tym samym zmniejszenia ryzyka istotnego pogorszenia płynności finansowej i ryzyka niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. W konsekwencji, jeśli chodzi o Skarb Państwa, może się to przełożyć na zmniejszenie ryzyka istotnego pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszenia wpływów podatkowych w porównaniu do sytuacji, gdyby takich rozwiązań nie wprowadzono. Intencje wynikające z projektowanej ustawy w naszej ocenie są słuszne i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku. Ta ustawa ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców oraz zapewnić zachowanie przez nich płynności finansowej. Projekt ustawy implementuje rozwiązania zbliżone do wdrażanych już rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej w odpowiedzi na światowy kryzys związany z COVID-19. Panie Marszałku!

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze przedstawiony rządowy projekt ustawy w tej sprawie. Dziękuję bardzo. A, przepraszam, pani poseł, jeszcze moment, bo o głos poprosiła pani minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pani Olga Semeniuk. Ale to może państwo pozwolą mi się teraz wypowiedzieć. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Z uwagi na COVID-19 i jego istotny wpływ na gospodarkę zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności handlowych dokonują przeglądu swoich portfeli.

Dlatego potrzebna jest systemowa odpowiedź, jaką proponujemy w niniejszej ustawie. Przyznane limity ubezpieczeniowe umożliwiły polskim przedsiębiorcom zrealizowanie i zabezpieczenie ponad 533 mld obrotów handlowych, w tym 118 mld zł dotyczyło transakcji zagranicznych, co stanowiło ogółem ok. 12% eksportu Polski. W zależności od rozwoju sytuacji istnieje zagrożenie, że ekspozycja ta może zostać zredukowana o 20% do 50% w porównaniu ze stanem sprzed pojawienia się pandemii COVID-19, a to może oznaczać redukcję limitów ubezpieczonych należności o 80 mld zł. Znaczne ograniczenie ubezpieczeń dla polskich przedsiębiorców oznaczać będzie tak znaczne podniesienie ryzyka transakcji, że tym samym doprowadzi do spowolnienia wymiany handlowej i całej gospodarki. Natychmiastowym skutkiem będzie istotne pogorszenie płynności finansowej, w tym znaczny wzrost ryzyka niewypłacalności. Dla Skarbu Państwa spadek transakcji handlowych będzie oznaczał pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszenie wpływów zarówno z tytułu podatków CIT, jak i VAT. Projektowane rozwiązanie ma na celu zniwelowanie tych wszystkich zagrożeń. Proponowany w przedłożonym Wysokiej Izbie projekcie ustawy mechanizm będzie polegał na zawarciu przez ministra rozwoju odpowiednio wystandaryzowanych umów reasekuracji z zakładami ubezpieczeń, które wyrażą chęć przystąpienia do programu rządowego. Tego typu reasekuracja zakłada, że Skarb Państwa w zamian za stały udział z składce ubezpieczeniowej przejmuje część ryzyka ubezpieczeniowego możliwych odszkodowań. Te poziomy składek będą ewoluować: 80%, potem 100% - po przekroczeniu pewnych kwot wypłaconych odszkodowań. Staramy się tym samym chronić przychody i płynność finansową zakładów ubezpieczeń, sprawiając jednocześnie, że po przekroczeniu określonej kwoty odszkodowań udział Skarbu Państwa w ryzyku ustaje. Wyznaczamy bezpieczną granicę zaangażowania państwa. Przeniesienie ryzyka dotyczy całych portfeli ubezpieczeniowych. Zakłady ubezpieczeń nie wybierają, co chcą nam przekazać, a czego nie. Nie ma zatem możliwości dokonywania przez ubezpieczycieli negatywnej selekcji ryzyka. Tym samym działamy systemowo, ale i zabezpieczamy interesy Skarbu Państwa przed szczególnie ryzykownymi zobowiązaniami. To rozwiązanie jest wzorowane ma mechanizmie niemieckim, które tam uruchomione na znacznie większą skalę już z powodzeniem jest wdrażane. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie projektu w kształcie zreferowanym przez komisję sejmową. Dodatkowo chciałam dodać informację związaną z wczorajszym posiedzeniem Komisji Finansów Publicznych, na którym w ciągu 2 godzin padło wiele pytań, na które starałam się razem z dyrekcją Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju odpowiadać.

Pani Wiceprzewodnicząca!

Chciałabym jeszcze tylko dodać, że wczoraj pojawiały się pytania dotyczące konstytucji, praworządności w związku z tym projektem, dlatego chętnie ustosunkujemy się drogą pisemną. Panie Marszałku! Pani Minister!

W tej ustawie wprowadzacie kontrolę incydentalną, ale ona jest niewystarczająca, bo ten rynek jest bardzo często przedmiotem fraudów, nieprawidłowości i wyłudzeń. Państwo nie może nad tym rynkiem przejmować odpowiedzialności, nie mając wpływu na poziom ryzyka. Dlatego nasz klub, klub Koalicji Obywatelskiej, złoży poprawkę, która rozszerza nadzór KNF-u właśnie nad tą częścią rynku finansowego w Polsce. Od przyjęcia tej poprawki uzależniamy tak naprawdę poparcie dla całej ustawy. Tak, dzisiaj jest tak, że firmy ubezpieczeniowe zawęziły gardło ubezpieczeń w obrocie wierzytelnościami. Prawdą jest, że nie chcą ubezpieczać. Ale dlaczego nie chcą? Bo zdają sobie z tego sprawę, że dzisiaj ryzyko wywracania się transakcji, niepłacenia należności przez kontrahentów jest bardzo wysokie, a ratingi poszczególnych kontrahentów mogą się zmieniać z dnia na dzień w zależności od sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach. I wy chcecie wejść w to miejsce i gwarantować, nie mając, tak jak powiedziałam, systemowego nadzoru. Podam pani minister przykład z ostatniego miesiąca.

Napisałam do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą, żeby skontrolowali tę transakcję, czy firma faktoringowa i ubezpieczyciel wywiązali się z umowy, czy faktycznie mieli podstawy do tego, żeby przerzucić całą odpowiedzialność na dostawcę, na kontrahenta. Mówili: my nie mamy nadzoru nad tą częścią rynku finansowego. I wy za tę część rynku finansowego, za wolny rynek i jego decyzje chcecie przejmować odpowiedzialność. To jest prosta droga do tego, co już w tym kraju przeżywaliśmy. SKOK-i zostały objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale nie zostały objęte nadzorem KNF-u, co spowodowało straty w postaci 5 mld zł.

Chcecie ratować system ubezpieczeń? Zróbcie to, jak należy. Bo ja nie mam pewności, że dzisiaj nie zaczniecie skupować wierzytelności od kolegów, polityków, ministrów, w przypadku których transakcje już się wywróciły, bo ustawa będzie sięgać wstecz, od kwietnia do końca tego roku. Jaką ja mam pewność, że ryzyko będzie odpowiednio ważone, że firmy ubezpieczeniowe będą ubezpieczać zdrowe należności i takie zdrowe należności będziecie przejmować, że w tych grubych, tłustych portfelach ubezpieczeń, które ostatecznie przejmie Skarb Państwa, nie będzie kolejnych pięciu czy dziesięciu dużych transakcji przyjaciół królika, w przypadku których się te transakcje wywróciły, ale w ten sposób odzyskają swoje należności? Nie, tak się nie robi, tak się nie zabezpieczy interesu Skarbu Państwa, a co za tym idzie - podatnika. To są pieniądze innych podatników.

Rynek wierzytelności handlowych i ubezpieczania tych wierzytelności handlowych jest jednym z tych rynków, które częściej padają ofiarą wyłudzeń, nadużyć i fraudów. I są firmy, które potrafią mieć 6% nieściągalnych należności, 6-procentowy poziom ryzyka, a są firmy, które potrafią mieć 50-procentowy. Tak jak powiedziałam, ona jest racjonalna, ona jest w obronie interesu państwa polskiego i polskich podatników.

Wysoka Izbo! Wszystko ma sprawiać wrażenie profesjonalizmu i troski o polskiego przedsiębiorcę, który stanął w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19, tyle że to tylko przykrywka. Tak, ryzyko nieściągalności należności wzrasta i wpływy maleją. Jest zrozumiałe, że w tej sytuacji powinniśmy znaleźć rozwiązania, które są adekwatne do danej sytuacji. Wszyscy przechodzimy kryzys, polscy przedsiębiorcy to wiedzą i starają się znaleźć rozwiązania, aby utrzymać biznes w tych trudnych warunkach. A co robią firmy ubezpieczeniowe? Czy negocjują umowy z klientami? Czy przyglądają się ryzyku? A może nie wypłacają sobie premii? Nie, nie, nie, nic z tych rzeczy.

Przygotowuje na kolanie ustawę, spieszy się, robi to bardzo szybko, aby zdążyć przed wakacjami. Nawet nie kryje się z tym, że celem ustawy jest, i tutaj zacytuję, utrzymanie dochodów ubezpieczycieli na tym samym poziomie co przed pandemią. Czyli troską rządu jest utrzymanie dochodów finansistów, żeby czasem nic nie stracili. To jest jasno napisane w uzasadnieniu. I nie myślcie, że w ten sam sposób rząd zatroszczy się o małych przedsiębiorców. O nie, nie, nie. Oni dostaną jednorazową zapomogę na przetrwanie, podobnie zresztą jak emeryci trzynastą emeryturę, a potem niech sobie radzą sami. Wszędzie na świecie od lat 60. dzieje się tak, że rządy wykorzystują wojny i katastrofy naturalne do bogacenia się bogatych. Świetnie opisała to Naomi Klein w swojej książce „Doktryna szoku”

Czy naprawdę chcemy mieć taki system agresywnego kapitalizmu jak w USA, ze słabą ochroną zdrowia, gdzie człowiek, gdy zachoruje, jest bankrutem, w kraju, w którym, żeby wyedukować dziecko, trzeba wziąć kredyt na dom? Rządzenie krajem to kwestia wyboru, jak podzielić ograniczone środki finansowe: czy przeznaczyć je na pensje dla nauczycieli, czy przeznaczyć je na pensje dla finansistów, czy zadbać o to, żeby każdy miał prawo do wizyty u lekarza specjalisty, czy też dać trzynastą emeryturę i powiedzieć: radź sobie sam, zapłać za kardiologa, za okulistę, za drogie leki, a jak sobie nie poradzisz, to trudno, to twoja sprawa. To politycy dokonują za nas tych wyborów. A dodam jeszcze, że te pieniądze pochodzą z podatków, czyli ciężko zarobionych naszych pieniędzy. Cała ta otoczka ministrów, krawatów ma sprawiać wrażenie, że projekt jest przygotowany profesjonalnie. Przyjrzyjmy się temu profesjonalizmowi. Po pierwsze, konsultacje. To jest projekt rządowy, zatem z mocy prawa powinien podlegać zaopiniowaniu, m.in. przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Biegłych Rewidentów, Radę Dialogu Społecznego i inne. Tych opinii nie ma. Pytam, dlaczego. Dlaczego ten projekt nie został skonsultowany i jest przepychany kolanem tuż przed wakacjami? Po drugie, konstytucja. Proszę państwa, ten projekt to jest gniot. Art. 3 ust. 1 ustawy mówi o tym, że Rada Ministrów może przygotować program wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych. Ten program ma określić: diagnozę sytuacji gospodarczej, oczekiwane efekty, cele programu, szczegółowe warunki realizacji, sposób raportowania, ocenę efektów i kwotę środków przeznaczonych na finansowanie programu. Pięknie, czyli ten artykuł, art. 3, mówi nam o tym, że głosujemy za ustawą, o której nic nie wiemy. Nie znamy diagnozy sytuacji gospodarczej, nie wiemy, jakie będą efekty gospodarcze, ekonomiczne i finansowe, nie wiemy, jakie są cele programu, nie wiemy, jak będzie wykonana ustawa, czyli w jaki sposób państwo będzie podpisywać umowy i jakie zawrze klauzule w tej umowie, nie wiemy, jak to będzie raportowane, i nie wiemy, ile to będzie kosztowało.

Przypominam rządowi, że. w Polsce źródłem prawa są: konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe i rozporządzenia. Nie ma w tym wykazie uchwał czy programów. Na Węgrzech.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska nasze stanowisko w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Można by powiedzieć w skrócie: taka kolejna odsłona kolejnej tarczy antykryzysowej, niestety po raz kolejny równie dziurawa jak te poprzednie, na potwierdzenie czego wiele argumentów wybrzmiało już z ust przedmówców. Omawiany projekt zakłada umożliwienie zakładom ubezpieczeń scedowania czy tzw. reasekurowania części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. Na tym ogólnym czy generalnym etapie chciałoby się powiedzieć: idea bardzo szczytna, ale przejdźmy do szczegółów. Rozwiązania zawarte w projekcie są reakcją na sytuację polskiego rynku ubezpieczeń - twierdzicie państwo jako projektodawcy. W otoczeniu, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa zakłady ubezpieczeń dokonują przeglądu swoich ofert, czego efektem może być znaczne obniżenie limitów albo likwidacja propozycji ubezpieczeń dla kontrahentów czy też niektórych branż i rynków. Skutkiem takich decyzji może być ograniczony dostęp przedsiębiorców do zabezpieczenia swoich transakcji. Znacznemu obniżeniu mogłyby również ulec ich obroty handlowe. Twierdzicie państwo, że według projektu Skarb Państwa pokryje 80% kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń, dotyczących ww. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r. W teorii wszystko się zgadza.

To jest dosyć zdumiewające, i to nie tylko w kontekście minionej kampanii prezydenckiej, gdzie ten przymiotnik „niemieckie”, „niemieckich” był, i to niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, odmieniany. Otóż kiedy Koalicja Polska przy pracach nad wszystkimi czterema tarczami antykryzysowymi powoływała się na przykłady rozwiązań właśnie wprowadzanych w Niemczech, wówczas państwo nie byliście zainteresowani, a takim kluczowym przykładem był fundusz płynnościowy właśnie przez Niemcy wprowadzony, dzisiaj pozytywnie, z powodzeniem oddziałujący na niemiecką gospodarkę.

Myślę, że ze strony Koalicji Polskiej jest taka rada dla projektodawców: zważcie państwo na te dziury i niedoskonałości tego projektu.

My musimy tworzyć rozwiązania, które będą sprzyjały wszystkim, i nasze poparcie dla tego projektu ustawy będzie właśnie uzależnione od tego, w jaki sposób ten projekt zostanie przez pomysłodawców uszczelniony i przygotowany, tak aby mógł służyć jak najszerszej grupie osób, którym rozwiązanie w nim zawarte ma być dedykowane.

Panie Marszałku! Po raz kolejny ze zdumieniem słyszę o stratach spowodowanych przez COVID. Nawet śmiertelność jest mniejsza, ponieważ rząd w tej sprawie nic nie zrobił.

Panie Marszałku! Wysoka Pustawa Izbo! O, Większości Parlamentarna! Wołacz - czasem zaniedbywana forma. O, Większości Parlamentarna! Przestańcie wreszcie szkodzić, to nie będziecie musieli rozwiązywać problemów, które sami wywołujecie. Polecam lekturę pożyteczną, świeżą: „Fałszywa pandemia” Fałszywa pandemia” - zbiór tekstów krytycznych naukowców i lekarzy. Uwaga. Szanowni Państwo! Socjalizm to jest ustrój, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów i wyprowadzaniem z kłopotów, które się samemu wygenerowało. I teraz ta socjalistyczna zasada w socjalistycznym - cóż, że eurosodosocjalistycznym - państwie, na którego czele państwo teraz stoicie, została podniesiona do potęgi przez walkę z mniemaną pandemią. Podnieśliście do rangi głównej zasady ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej nadużycie uprawnień. Stworzyliście mgławicę bezprawia, dopuszczając do tego, żeby życie Polaków, w tym także polskich przedsiębiorców, handlowców, także ubezpieczycieli, zostało podporządkowane działaniu nie prawa, poważnego prawa, aktów wyższej i najwyższej rangi, ustawowych, konstytucyjnych. Dopuściliście do tego, żeby nasze życie, ze szczególnym uwzględnieniem życia gospodarczego, było zdane na łaskę i niełaskę władzy, która poprzez rozporządzenia ministerialne i następnie zmieniające się w czasie w tempie kalejdoskopowym wytyczne do tych rozporządzeń. No i teraz przychodzicie po raz kolejny do Wysokiej Izby z rozwiązaniami rzekomo pomocowymi. Jeszcze raz powtórzę: nie szkodźcie. Przestańcie podtrzymywać pandemiopsychozę, przestańcie podniecać koronapanikę w Rzeczypospolitej Polskiej. Skierujcie służby i administrację - po, rzecz jasna, jej należytym odchudzeniu - do ich właściwych zadań. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić, kiedy przyjdzie czas rozważać wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych, koordynatora Kamińskiego. Będziemy mówić o hańbieniu munduru polskiego policjanta przez kierowanie funkcjonariuszy do zadań, które hańbią i ośmieszają polską Policję. Wycofajcie się z tego obłędu. Nie budujcie polityki państwa na podstawie dezinformacji, która w zagranicznej telewizji jedzie na pasku. Nie podporządkowujcie się, nie działajcie, jakbyście byli na pasku zagranicznej telewizji, ale prowadźcie suwerenną politykę. Otwórzcie gospodarkę. Przestańcie terroryzować klientów i handlowców tymi właśnie rozporządzeniami i wytycznymi. Przestańcie inicjować łapanki na normalnych ludzi. Przestańcie generować w narodzie gestapowskie, enkawudowskie donosicielstwo, które już przeszło do historii, boście to rozbuchali.

Jeszcze raz polecam panu marszałkowi i panu posłowi sprawozdawcy - za chwilę wręczę egzemplarz - książkę „Fałszywa pandemia”, która dzięki Fundacji Osuchowa jest już dostępna. Do pytań zgłosili się państwo posłowie. Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Pierwsza pani poseł Hanna Gill-Piątek, Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Pośle! Wysoka Izbo!

Dotyczy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która miała zastąpić wydziały handlowe ambasad. Niestety zamiast promować polską gospodarkę za granicą, agencja nie umie się sama zorganizować. Według doniesień „Pulsu Biznesu” otwierane z pompą biura na całym świecie w wielu miejscach okazały się zupełnie niewydolną, jednoosobową działalnością mającą kłopot z legalizacją działań czy ubezpieczeniem pracowników. Za to poziom zatrudnienia na stanowiskach dyrektorskich w centrali wzrósł w 2019 r. z 10 do 40, czyli o 400%. Art. 8 to wrzutka dolewająca do PAIH kolejną kasę, tym razem z funduszy COVID-owych.

Wysoka Izbo! Wsparcie dla przedsiębiorców, tworzenie nowych miejsc pracy, a także utrzymanie istniejących miejsc pracy powinno być zadaniem i priorytetem rządu nie tylko wtedy, kiedy jest COVID, ale generalnie każdego miesiąca i każdego dnia. Na to, czy ludzie w Polsce będą prowadzić działalność gospodarczą, czy będzie się rozwijała przedsiębiorczość, ma wpływ bardzo wiele elementów.

Jeśli nie będzie dobrej atmosfery, jakakolwiek jednorazowa pomoc z okazji COVID-u czy innej okazji nigdy nie będzie wystarczająca. Weźcie państwo pod uwagę te propozycje, które padają ze strony opozycji.

Panie Marszałku! Pytanie zasadnicze: Kogo tak naprawdę chcecie wspierać? Czy instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe tym razem? Niedawno takie wsparcie przygotowaliście dla instytucji bankowych. To im tak naprawdę gwarantujecie ograniczenie ryzyka do minimum, gwarantujecie rentowność, wpychając, nawiasem mówiąc, kasę do instytucji prywatnych bez żadnej kontroli i bez żadnego nadzoru, o czym już mówiła koleżanka. Mamy świadomość, że ubezpieczenie transakcji ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu także przedsiębiorców. Jest instytucja, którą państwo ma pod pełną kontrolą, którą wystarczyłoby dokapitalizować, mówię tu o KUKE, żeby sytuację, jeśli chodzi o eksporterów w tych trudnych czasach wyraźnie poprawić. Pan poseł Michał Szczerba. Nie ma pana posła. Pan poseł Paweł Krutul, klub Lewicy.

Daleko, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przedstawiona przez rząd ustawa pokazuje, że cała polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości jest de facto życzeniowa i nie działa. Przecież przeprowadziliście państwo repolonizację, macie swoich ludzi w bankach, w zakładach ubezpieczeń. Teraz pani minister przychodzi i mówi, że ci ludzie będą zwijać działalność ubezpieczeniową. Po co była ta cała repolonizacja, skoro jest tak, jak było? Posadziliście tam swoich i to po prostu nie działa. Oczywiście przedsiębiorców trzeba wspierać, ale to, co rząd proponuje, to jest de facto zwolnienie z odpowiedzialności korporacji.

W jaki sposób rząd zamierza zabezpieczyć prawidłowe szacowanie ryzyka, bo na ten temat w ustawie nic nie ma (Dzwonek), a zakłady ubezpieczeń będą miały gwarantowane zyski? W związku z tym jak zabezpieczycie prawidłowe szacowanie ryzyka? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jakie mamy gwarancje zachowania transparentności oraz uczciwości przy sprawowaniu kontroli przez KNF nad sposobem realizacji umów i wniosków związanych z projektem ustawy? Jak sami państwo przyznają w uzasadnieniu, kluczowe jest uzyskanie oceny Komisji Europejskiej. Kto będzie odpowiadał za czas rozmów oraz ich przebieg i ewentualne skutki? Rząd weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnej porażki rozmów z Komisją Europejską. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pewnie projekt ustawy i te założenia idą w dobra stronę, bo nie ma wątpliwości, że przedsiębiorcom w Polsce trzeba pomagać, natomiast jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Moje pytanie jest następujące. Po pierwsze: Czy polski rząd ma ocenę sytuacji, jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe?

Czy ta informacja była przedstawiana przez polski rząd? Proszę się nie dziwić, że opozycja ma duże obawy, że rząd może wprowadzić program, minister może refinansować.

Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym powiedzieć o dwóch mankamentach tego projektu. Po pierwsze, powołujecie się państwo, przedstawiając projekt, na rządowy program wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych, a tego programu nie przedstawiono.

Jak możemy zważyć ryzyko, jeżeli państwo zapisali fakultatywność zwrócenia się do Komisji Nadzoru Finansowego o opinię w zakresie realizacji ustawy i umów o przejęciu gwarancji za 80% rynku ubezpieczeń, portfela ubezpieczeń, należności handlowych? To są dwa główne mankamenty, które, jeśli nie zostaną wyeliminowane, będą stanowiły mocne zagrożenie dla rzetelności przeprowadzenia takiego zabezpieczenia dla kontrahentów.

Pani czas się skończył. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Mam pytanie do pana posła sprawozdawcy. Panie pośle przewodniczący, mówił pan w sprawozdaniu, że w czasie prac przyjęto rozwiązania ograniczające górną granicę ryzyka ubezpieczonego ponoszonego przez Skarb Państwa. Chciałem wobec powyższego zapytać: Czy rozwiązania przyjęte przez komisję w trakcie prac w drugim czytaniu ograniczą udział Skarbu Państwa planowany pierwotnie na kwotę 2,7 mld zł na najbliższe 4 lata, czy jednak to tylko i wyłącznie uszczelnia tę ustawę, a poziom zaangażowania Skarbu Państwa pozostaje na zakładanym poziomie? Dziękuję. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, Lewica. Wysoka Izbo! W przedłożeniu proponuje się, żeby należności, o których w nim mowa, dotyczyły umów z kontrahentami mającymi siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w krajach wymienionych w załączniku i są to enumeratywnie, konkretnie określone kraje. Są to kraje Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Stany Zjednoczone Ameryki.

Dlaczego po raz kolejny zapominamy o naszych sąsiadach na wschodzie, mam na myśli konkretnie Ukrainę.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Jakub Kulesza, koło Konfederacji. Wysoka Izbo! Fryderyk Bastiat powiedział, że dobrego ekonomistę od złego odróżnia to, że dobry ekonomista jest w stanie zauważyć te niewidoczne, dalekosiężne skutki pewnych działań politycznych i ekonomicznych. Mam wrażenie, że za sytuację, którą mamy w Polsce, nie odpowiadają dobrzy ekonomiści z rządu. Mam wrażenie, że nawet źli ekonomiści nie odpowiadają, tylko epidemiolodzy, którzy, nie patrząc na skutki ekonomiczne dla kraju, stwierdzili, że jedynym celem rządu jest walka z tą a nie inną chorobą. Jaki mieliśmy tego efekt? Szybko po zamknięciu kraju okazało się, że cała gospodarka stanęła. Ta gospodarka została odmrożona, uwaga, w sytuacji, w której wszystkie wskaźniki epidemiologiczne były gorsze niż przy zamykaniu, co pokazuje, że to była zła decyzja.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam dwa, może trzy pytania.

I ostatnie pytanie: Czy nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym będzie rozszerzony w ramach funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego?

Pani Minister!

Tam jest mowa o zniesieniu odpowiedzialności polityków PiS za przekroczenie uprawnień, za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Pani minister, kto jest autorem tego przepisu?

Czy chodzi o to, żeby w kręgu ministra zdrowia nadal pojawiały się podmioty, kolejni instruktorzy narciarstwa, kolejni handlarze bronią, którzy potraktowali pandemię jako żyłę złota? I jak zabezpieczyć, pani minister, Skarb Państwa przed nieuczciwymi kontrahentami? Teraz głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Henryk Kowalczyk. Panie Marszałku! Do sprawozdawcy komisji padło jedno pytanie o górny limit wydatków Skarbu Państwa. A więc odsyłam oczywiście do art. 4 tej ustawy, ust. 3 określa, że zobowiązanie Skarbu Państwa nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w roku 2019. Chodzi o 375% przypisanej składki brutto.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 455 i 480) Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! Wczoraj, 14 lipca, odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poświęcone pierwszemu czytaniu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, druk sejmowy nr 455.

Wprowadza ona definicję drewna energetycznego umożliwiającą wykorzystanie niszczejących obecnie w lasach nadwyżek drewna, wynikających z epidemii koronawirusa, do celów energetycznych. W trakcie procedowania nad ustawą został zgłoszony wniosek o jej odrzucenie w pierwszym czytaniu. Komisja w głosowaniu nie poparła tego wniosku. Posłowie zgodzili się na poprawki legislacyjne, a także został zmieniony termin jej wejścia w życie z dnia 1 lipca na dzień 1 października 2020 r. Niniejsza ustawa została notyfikowana przez Komisję Europejską w dniu 4 czerwca 2020 r.

Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedłożyć nasze stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, druk nr 455. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa i po wielu godzinach dyskusji komisja poparła ten projekt.

Dlatego projekt przewiduje czasową zmianę definicji drewna energetycznego zawartej w ustawie o OZE. Klub Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt ustawy. Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nie palcie naszych lasów. Polska stoi przed szansą uzyskania dodatkowych 8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, natomiast wypłata tych środków, zgodnie z zapowiedziami, może zostać uzależniona od deklaracji osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do roku 2050 na poziomie krajowym. W skrócie: Europa każe nam odchodzić od węgla i przejść na energię odnawialną. Co robi polski rząd? Co robi Ministerstwo Środowiska? Jako jedyne w Europie nie popiera wyzwania dotyczącego przejścia na neutralność klimatyczną do roku 2050 i składa projekt ustawy, który de facto pozwala na palenie w polskich elektrowniach polskim lasem, który nazywacie państwo biomasą. To jest okradanie Polaków z zasobów naturalnych, z bioróżnorodności, z polskich drzew.

Przedstawiciele ministerstwa uspokajają nas i uspokajali nas wczoraj, że nowelizacja nie doprowadzi do niekontrolowanych wycinek i wywózek martwego drewna. Ale, proszę państwa, historia brutalnej wycinki Puszczy Białowieskiej, ekstensywnych wycinek, które dzieją się dzisiaj choćby w Puszczy Karpackiej, na terenie całej Polski, pogłębia nasz brak zaufania do państwa, kiedy próbujecie nas uspokajać.

Tymczasem Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego mówi nam, że trudności w zbyciu drewna przez Lasy Państwowe narastają już od lat i nie wynikają z epidemii, ale ze zbyt wysokich cen, w jakich drewno jest oferowane. Ministerstwo skarży się na problemy z płynnością finansową Lasów Państwowych. To też nas martwi. Natomiast pytam: Co zrobiliście państwo od roku 2015, od czasu ogłoszenia raportu NIK, który jasno wykazał, iż problemy finansowe Lasów Państwowych mają źródło w wysokich kosztach administracyjnych, w wysokich kosztach stałych, natomiast Lasy Państwowe zbyt mało inwestują w ochronę polskich lasów? Podsumowując, ta zmiana, którą państwo nazywacie remedium na poprawę finansów Lasów Państwowych i krokiem w kierunku rozwoju energii odnawialnej, zasługuje na miano ustawy dewastującej polską przyrodę, bioróżnorodność, a w efekcie - nasz klimat i nas samych. My na to nie pozwolimy. Chcemy dalszych prac i porządnych konsultacji społecznych, które się nie odbyły. Dlatego składam poprawkę na ręce pani marszałek.

Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Ja też powtórzę to samo: nie palcie naszych lasów.

Od tego czasu są stale przymiarki do zamiany Lasów Państwowych nie tylko w plantację desek, ale także plantację opału. Tym opałem chcecie palić w elektrowniach, chcecie spalić polskie lasy, tak jakby to była wasza własność. To jest dobro narodowe, dorobek całej Polski, wszystkich Polek i Polaków. Dysponuje się nim bez konsultacji społecznych, bez rozmów z kimkolwiek, z ekspertami. Niszczy się bioróżnorodność na taką skalę, która zagraża wyginięciem gatunków. Jedynym kryterium jest kryterium czysto merkantylne: uprawa lasów, czyli plantacja dla pieniędzy, dla destrukcji. Las jest dla Polaków czymś więcej niż taką plantacją, las jest naszym największym bogactwem, tak samo jak nasze parki narodowe i puszcze. Nie palcie tego największego bogactwa, które mamy, bo przyrody nam nikt nie zwróci. Tej przyrody nie zawdzięczamy sobie ani żadnym kolejnym władzom i kolejnym ministerstwom. Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, klub Lewicy. Szanowna Izbo! Panie Ministrze! Lasy są niezbędne dla zachowania bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu, a także regulowania zasobów wody. Kryzys klimatyczny i środowiskowy będzie tym silniej nas dotykał, im gorzej będziemy chronić bioróżnorodność, różnorodność biologiczną. Im bardziej będziemy wycinać, ingerować, tym mniej będziemy przygotowani na kryzys klimatyczny, na katastrofę klimatyczną. To jest konsensus naukowy, to są fakty. Wiem, że w uszach części leśników zabrzmi to jak bluźnierstwo, ale przypomnę: lasy to nie plantacje, to nie farmy. Bilans ich funkcjonowania to nie są cyferki w dokumentach księgowych Lasów Państwowych. Lasy są dobrem wspólnym, dobrem wszystkich obywateli i będą kluczowe dla zapewnienia nam wszystkim bezpiecznej przyszłości. Co tymczasem przygotował dla polskich lasów minister Woś pod dyktando Lasów Państwowych? Projekt nowelizacji, który możemy podsumować jednym absurdalnym zdaniem: A teraz, żeby obniżyć emisję dwutlenku węgla, będziemy ścinać jeszcze więcej drzew w lasach, będziemy palić nimi w elektrowniach i udawać będziemy, że tak nam każe Unia Europejska. No nie, nieprawda. Absurdalna w tym przypadku jest ta propozycja rozszerzenia pojęcia drewna energetycznego, tak by mogło być traktowane jako biomasa. Biomasa jest wprawdzie dopuszczalna jako OZE w bilansie energetycznym, ale tylko jako źródło dodatkowe. Plus, co jest bardzo ważne, w dobie katastrofy klimatycznej eksperci jasno mówią, jasno pokazują, że od tej biomasy, od drewna energetycznego powinniśmy odchodzić. To nie jest rozwiązanie. A to, co proponuje nam minister Woś, to umożliwienie spalania w charakterze biomasy pełnowartościowego drewna pochodzącego z polskich lasów. Wbrew temu, co mówi ministerstwo, ta zmiana niewątpliwie doprowadzi do dewastacji polskich lasów. Mówicie: Nie zwiększymy wycinek, bo są plany urządzania lasów. Jak możemy w to wierzyć, skoro te pule są aneksowane i wycinki się zwiększają z roku na rok? Minister Woś tłumaczy, że wycinki drzew są konieczne ze względów sanitarnych, ze względu na walkę ze szkodnikami. Tak, to jest pretekst. Oczywiście każdy pretekst jest dobry, żeby zwiększyć wycinkę, tylko podkreślmy: właściwe zarządzanie lasami nie może prowadzić i nie prowadzi do tak drastycznych wycinek. Minister Woś chce wycinać martwe, zamierające drzewa. Dlaczego? Dlatego że one nie przyniosą pieniędzy Lasom Państwowym. I to nie pierwszy raz, kiedy przyszłość, kiedy ważne rozwiązania są odrzucane dlatego, że liczy się jedynie zysk kilku osób, które teraz zajmą dobre miejsca w Lasach Państwowych i będą mogły uprawiać politykę. Nawet jeśli chodzi o stronę kosztową, to zaledwie 13% jest przeznaczone na cel podstawowy, jakim jest uprawa lasów i zwiększanie ich powierzchni. Okresowy spadek przychodów ze sprzedaży drewna nie zachwieje podstawami finansowymi tego przedsiębiorstwa. Może zachwiać pensjami dyrektorów, polityków, których państwo zatrudniają na stanowiskach regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych. Ja wiem, że ten antyobywatelski rząd nie interesuje się dialogiem z organizacjami pozarządowymi. Widzieliśmy to wczoraj i widzimy to na co dzień. Wiemy, że ten antynaukowy rząd nie interesuje się także dialogiem z ekspertami. To widzimy w codziennych pracach Ministerstwa Środowiska. To może chociaż, jak już tak machacie tymi chorągiewkami pt. „przedsiębiorcy”, posłuchajcie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego mówią, że ta ustawa to katastrofa, to marnotrawstwo, że to zalegające podobno drewno, którego nikt nie chce kupić, oni chcą kupić. Nie mogą tego zrobić. Dlaczego? Ponieważ ustanowiliście państwo tak wysokie ceny, że ich po prostu na to nie stać. Pisali do Ministerstwa Klimatu, zwracali się do Ministerstwa Środowiska, napisali do Ministerstwa Rozwoju. Zobaczyli tę wyciągniętą rękę? Jeżeli już jesteśmy przy Ministerstwie Rozwoju - nawet to ministerstwo w opinii do tej ustawy pisze o jej negatywnym wpływie na sektor polskiej gospodarki, na ten sektor, który zatrudnia 350 tys. pracowników i generuje 2,5% PKB. Więc może odnieście się państwo - i tu zwracamy się do Ministerstwa Rozwoju - do tego, co ta ustawa zrobi polskim przedsiębiorcom. My wnosimy nasze poprawki, ale także chcemy, aby ta ustawa była dyskutowana w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jako komisji odpowiedniej do dyskusji o lasach. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.

To nie jest żadna ustawa o OZE. To jest ustawa o wycince lasów, o niszczeniu polskich lasów.

Po prostu uwalniamy CO2 do atmosfery, spalając. I stąd, panie pośle, te wszystkie zakłócenia w klimacie są. I bardzo dobrze - niech się ludzie topią, niech giną.

Ale wracając do ustawy: spalanie drewna w piecach, w elektrowniach jest bardzo złym rozwiązaniem - i od tego trzeba zacząć - bo ono niczym nie różni się od spalania węgla. My krytykujemy spalanie węgla, nieodchodzenie od czarnej energii, natomiast spalamy drewno.

Ja sobie przypominam czasy, kiedy PiS walczył z prywatyzacją lasów.

Zabierał głos, mówiąc: nie dopuścimy do prywatyzacji lasów.

To jest nieuczciwe. Wykorzystujecie sytuację związaną z COVID-em. Trudna sytuacja itd., COVID jest wszystkiemu winien, więc idźmy do lasu, tnijmy lasy, niszczmy lasy. Dzisiaj, kiedy zaczynają się kłopoty - racjonalne rozliczenie zacznie się już z końcem roku, czy mamy 15%, czy nie mamy - kiedy przyjdzie nam kupić prawdopodobnie energię odnawialną albo zapłacić karę, trzeba szukać innych rozwiązań, które pozornie stworzą - zgodnie z prawem oczywiście - ale to prawo źle funkcjonuje. Bioróżnorodność, to jest bardzo ważne i bardzo istotne, bo dzisiaj, gdy mówimy o ochronie lasów, to znaczy, że chcemy zachować lasy w naturalnej ich formie, a nie mechanicznie robić czystkę i co się da, to dawać do pieców. Jeżelibyśmy popatrzyli z kolei na inwestycje w energetykę, to popełniamy ogromny błąd, dlatego że inwestujemy w te urządzenia, które są przy bardzo starych już blokach energetycznych, które za kilka czy kilkanaście lat, za kilka lat przestaną funkcjonować, a my inwestujemy we współspalanie. I pytanie, co dalej, kiedy te bloki energetyczne nam się skończą. Z czego będziemy się rozliczać w energii odnawialnej? Dzisiaj mamy możliwości pozyskania energii odnawialnej ze słońca, z wiatru, z biogazu, z czystych źródeł - to są czyste źródła, naturalne źródła, niewyczerpywalne źródła.

Przypominamy sobie dyskusje tutaj, kiedy mówiono, że już mamy nadmiar energii odnawialnej, że już nie potrzeba nam więcej, że zapłaciliśmy ogromną cenę. Dzisiaj okazuje się, że energia odnawialna jest znacznie tańsza.

Wysoka Izbo! Patrzymy na projekt ustawy i widzimy ograniczoną w czasie regulację wprowadzającą definicję drewna energetycznego, i widzimy to jako rozwiązanie problemu, który pojawił się w związku z epidemią. Problemu, który de facto, i to jest raczej problem, powiedziałbym, ustrojowy, nie powinien być rozwiązywany przez kolejną ustawę, tylko powinien być rozwiązywany - i taka powinna być konstrukcja naszego państwa i naszego prawa - żeby tego typu problemy, że drewno zalega, to drewno gorszej jakości, chrust, igliwie, drewno małowymiarowe, liście, kora, korzenie i karpy, drewno pełnowymiarowe gorszej jakości.

Natomiast, szanowni państwo, to jest racjonalne. I oczywiście Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną. Tak, prowadzą gospodarkę leśną. Mówienie o lasach naturalnych jest jakąś aberracją, nieporozumieniem. To, czy ta polityka zasadzeń była właściwa przez dekady, a mamy problem z monokulturą i inne tego typu rzeczy, to jest zupełnie inna dyskusja.

Proszę państwa, to, co dzisiaj pada tutaj z tej mównicy, jest bardzo groźne, dlatego że my - i w ogóle powinniśmy na ten temat przeprowadzić fundamentalną debatę - stoimy wobec zagrożenia, jakim jest Europejski Zielony Ład.

Teraz mamy, to jest informacja z wczoraj, najwyższe ceny, jeśli chodzi o handel emisjami. Gwałtownie wzrasta to, co musimy płacić ze względu na ideologiczną, błędną politykę Unii Europejskiej. Dzisiaj polską racją stanu jest odrzucenie tych regulacji. Zwracam państwa uwagę, że czeski senat już przetarł nam szlak, naprawdę. Są odważni w naszej części Europy. Proszę państwa, rozprawmy się też z mitem, że gwałtowna likwidacja polskiej energetyki opartej na węglu cokolwiek zmieni w sprawie klimatu w skali ogólnoświatowej.

Tam będą wzrosty.

Chodzi o powszechne wprowadzenie energii jądrowej, również w Polsce. I wszystkie ekipy są za to odpowiedzialne, że ta energetyka jądrowa leży i kwiczy. I PiS też od 5 lat zapowiada, pan prezydent Duda w kampanii wybrał się do Stanów Zjednoczonych, coś tam mieli niby obiecywać, gadać. Chcecie czystej energii? To jest prawda.

Jako pierwszy pan poseł Andrzej Szewiński, klub Koalicji Obywatelskiej.

Wysoka Izbo! Nie palcie polskich lasów. Wszyscy mamy w pamięci wprowadzone niedawno prawo, którego efektem była dewastacja polskiego drzewostanu. Mówię tu o lex Szyszko. Obecnie pochylamy się nad kolejnym bublem, który umożliwi wycinanie i spalanie w charakterze biomasy drzew pochodzących z polskich lasów. Spalane będą drzewa martwe i zamierające, czyli takie, które nie są wartościowe z punktu widzenia produkcji surowcowej, ale są kluczowe jeśli chodzi o ochronę różnorodności biologicznej ekosystemu leśnego. Mam wrażenie, że projektodawcy nie wzięli pod uwagę, iż wycinka i systemowa likwidacja tzw. drzewostanu martwego zasiedlonego przez gatunki fauny spowoduje, że wiele gatunków zwierząt bezpowrotnie zginie.

Panie Ministrze!

Przypomnę, że 8 lat temu dokładnie to miało miejsce i trzeba było wprowadzać zmiany w przepisach, żeby ograniczyć właśnie spalanie drewna w elektrowniach.

To jest bardzo istotne z punktu widzenia przyjmowanej ustawy.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak łatwo zmienić definicję. Może lepiej od razu wpisać, że węgiel też jest energią odnawialną, mielibyśmy 100% wykorzystania energii OZE w Polsce.

No, Ostrołęka czeka cały czas na wsad, to może to drewno będzie zbawieniem dla elektrowni w Ostrołęce. Pani poseł Mirosława Nykiel, klub Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Nie palcie polskich lasów. Rząd, zmieniając definicję drewna energetycznego w tej ustawie, chce spalać drewno w elektrowniach. Jakby ktoś zapytał: O co tu chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie słuchacie opinii posłów opozycji, do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Nie słuchacie opinii ekspertów, nie słuchacie organizacji przyrodniczych i ekologicznych. Wszyscy - tutaj już było to mówione - wiemy, że to nie jest towar, który przynosi zysk. I moje pytanie do przedstawicieli rządu jest następujące: Czy macie świadomość, że wprowadzając te przepisy pod dyktando Lasów Państwowych będziecie odpowiedzialni za skalę wycinek i dewastację najcenniejszych przyrodniczych obszarów, lasów [[Dzwonek]] w Polsce?

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze!

To jest 285 mln zł. Pan minister Kowalczyk takie zarządzenie wydał. Powstaje pytanie: Czy polscy przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani tym drewnem, dzisiaj nie mogą go nabyć ze względu na wysoką cenę?

Pan poseł Andrzej Grzyb, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wykorzystanie drewna powinno być zgodne z zasadami piramidy wykorzystania biomasy.

Wydaje mi się, że to byłby doskonały moment, żeby w ramach pomocy COVID-owej również to stymulować (Dzwonek) i zgromadzić pewnego rodzaju zasoby.

Wysoka Izbo! PiS zawsze musi mieć wroga, nawet w naturze: kiedyś kornik, dzisiaj owady. Tak wygląda polityka partii rządzącej, ekologiczna polityka. Muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo nie wiedziałam, że odnawialne źródła energii oznaczają wycinkę, sprzedaż i spalanie drzewa z lasów państwowych. To jest oszukiwanie społeczeństwa. To nie jest ratowanie środowiska, tylko ratowanie katastrofalnej sytuacji przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, o czym pisze w raporcie NIK wasz kolega, Banaś. Jeśli chcecie coś ratować, to zacznijcie od zdrowia i życia ludzi i stwórzcie przepisy, na które czekamy, o które proszę, po to aby powstał lek na COVID-19 z osocza ozdrowieńców. Tym powinniście się zająć, tym właśnie, a nie ratowaniem lasów państwowych przed owadami.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedłożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii to kolejny akt prawny, który został przygotowany w pośpiechu, wbrew zasadom prawidłowej legislacji i dobremu obyczajowi parlamentarnemu. Projektu nie przekazano do konsultacji organizacjom ekologicznym, nie dostały go także samorządy. Konsultacje obejmowały jedynie organizacje związane z Lasami Państwowymi i branżą energetyczną. Najbardziej bulwersująca jest zmiana dotycząca definicji surowca drzewnego, który mógł być wykorzystywany energetycznie. Jeśli ustawa zostanie przegłosowana w obecnej formie, to sektor energetyczny praktycznie bez ograniczeń będzie mógł spalać surowiec wykorzystywany obecnie przez przemysł drzewny, co pogłębi kryzys w branży spowodowany pandemią COVID-19 i doprowadzi do wzrostu cen, a także ograniczy konkurencyjność polskiego przemysłu meblarskiego na rynkach zagranicznych, a trzeba pamiętać, że jesteśmy szóstym na świecie producentem mebli.

Szeregowy Pośle Kaczyński! Wysoka Izbo! Po pierwsze, jednym z najważniejszych założeń demokracji jest tworzenie prawa oparte na dialogu pomiędzy społeczeństwem a jego przedstawicielami. W takim razie dlaczego zaniechali państwo konsultacji społecznych dotyczących tego projektu? Proszę o wyjaśnienia. Po drugie, kilka lat temu zadałam pytanie w Internecie: Po co komu drzewa? Przecież zabierają miejsca parkingowe, brudzą i zasłaniają widok na Polskę wstającą z kolan. Była to smutna satyra na masowe wycinanie drzew i lasów rozpoczęte za rządów PiS-u. Niestety w kraju, gdzie rządzący nie potrafią zrozumieć ironii, potraktowali tę moją wypowiedź poważnie. Dzisiaj znaleźli kolejny absurdalny powód, by tym razem palić lasy. Zrobicie wszystko, by postawić na swoim. Tylko pamiętajcie, że w Polsce bez drzew, lasów, wody, zwierząt, zabetonowanej, z najgorszym powietrzem w Europie, czarnej od węgla - na tej pustyni zostaniecie sami, nawet bez ludzi. Bo kto chciałby mieszkać w takim smutnym, szarym od dymu, betonowym świecie? Pomyślcie o tym. Poseł Wanda Nowicka, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Lasy narodowe to nasze dobro narodowe i dlatego chciałabym powtórzyć za obywatelami, którzy wczoraj protestowali przed Sejmem: nie palcie naszych lasów. Ludzie czują, że lasy należą do nas, chcą decydować o lasach, tymczasem wy, traktując lasy jak deski, a teraz - biomasę, nawet nie chcecie z ludźmi na ten temat rozmawiać, nie chcecie wysłuchać ich stanowiska, co oni sądzą o takiej polityce, która lasy traktuje wyłącznie, jak mówię, jak deski, jak coś, co można spalić i nie troszczyć się o nasze dobro i o środowisko naturalne. Nie palcie naszych lasów - tak mówili wczoraj ludzie. Weźcie to wreszcie pod uwagę. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jeżeli nie potraficie tego zrobić, to może my wam podpowiemy. Nasi przedsiębiorcy, którzy przetwarzają drewno, potrzebują tego drewna, ale nie w takich cenach, w jakich dzisiaj im oferujecie. To jest jedna rzecz. Może warto pomyśleć, w jaki sposób ograniczyć dopływ tego taniego drewna z zagranicy. To jest drugi temat, którym można byłoby państwa zainteresować.

Ironizując, można by powiedzieć tak: szanowni państwo, może spalmy lepiej te niewykorzystane karty do głosowania z pierwszej tury. Może to byłoby lepsze. Szanowni państwo, dlaczego chcemy, żeby Polacy dotowali dzisiaj Lasy Państwowe?

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Z całego serca dziękuję wszystkim aktywistom i aktywistkom, którzy protestowali wczoraj w Sejmie przeciwko tej barbarzyńskiej ustawie. Ustawie, która forsowana jest bez prawdziwych konsultacji społecznych, o czym organizacje pozarządowe informowały we wspólnym apelu. Władzy po raz kolejny brakuje odwagi, żeby rozmawiać. Gdy cały świat zastanawia się, co zrobić w obliczu katastrofy klimatycznej, propozycja palenia drzew w elektrowniach jest jakąś kpiną, jest jakimś żartem. W tym czasie pan minister woli rozmawiać przez telefon. Nie będę w takim razie przerywał, powiem do reszty. Z inspiracji rządu drzewa stają się towarem, a leśnicy są biznesmenami, którzy mają wypracowywać zysk. Zwracam się do rządu z prośbą o wycofanie się z tego projektu, a także z pytaniem. Według projektu drewnem energetycznym mają być także drzewa pozyskiwane z wycinki przy drogach publicznych i szlakach kolejowych.

Szanowni Państwo! Rozszerzenie definicji biomasy o najwyższej jakości drewno to biomasakra. Dlaczego nie wykorzystacie okazji, że branża meblarska zanotowała krótkotrwały kryzys wynikający z pandemii, do zmniejszenia limitów pozyskiwania drewna w wieloletnim planie urządzenia lasu? Zmniejszcie podaż, skoro jest mnóstwo drewna posuszowego. Mierzymy się ze skutkami zmian klimatu i wielkiego wymierania gatunków. Teraz fundujecie puszczanie lasów w komin. To nie jest miks energetyczny, to masakra. Ministerstwo twierdzi, że chroni lasy przed zagrożeniem pożarowym. To wytnijcie wszystkie lasy, nie będzie miało się co palić. Według Najwyższej Izby Kontroli tylko 13% wydatków Lasów Państwowych przeznaczanych jest na ochronę i hodowlę lasów. Co się dzieje z resztą pieniędzy?

Wysoka Izbo! Najpierw definicja OZE. Są to takie źródła energii, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawialne. Proszę mi powiedzieć, jaki ekspert dokonał tej interpretacji, że drzewo, które rośnie kilkadziesiąt lat, jest takim samym źródłem energii jak woda, wiatr czy słońce. Chciałbym go szybko poznać, bo wiem, że niebawem da wam taką interpretację węgla, który także będzie spełniał definicję odnawialnego źródła energii. Bądźmy szczerzy, ta nowelizacja jest grubymi nićmi szyta. Chodzi o pieniądze. Dowodem jest fakt, że niedawno zmieniliście matrycę VAT. Na tej transakcji chcecie po prostu więcej zarobić, przy okazji krzywdząc wiele tych osób, które niestety jeszcze do dzisiaj ogrzewają swoje mieszkania drewnem opałowym. Pani poseł Małgorzata Tracz, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu czytamy, że za przyjęciem nowelizacji przemawia rzekomo fakt, że drzewa martwe występujące w lasach na terenie Polski mają miąższość wynoszącą dziesiątki milionów metrów sześciennych. Tymczasem wiadomo, że Polska jest krajem o niskich zasobach martwego drewna na tle lasów w innych państwach Unii Europejskiej. Wiadomo także, że drzewa martwe i zamierające są siedliskami i żerowiskami wielu cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej. Wiemy także, że już obecnie przeciwko Polsce toczy się postępowanie o naruszenie prawa Unii Europejskiej z uwagi na zwolnienie gospodarki leśnej z zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Jak projektodawca zamierza wytłumaczyć się z kolejnej zmiany prawa, która zezwalając na spalanie drzew martwych i zamierających, uderza w ochronę leśnych gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej? Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dlaczego ustawodawca nie przyjmuje do wiadomości opinii niezależnych ekspertów i autorytetów naukowych? Wzrasta populacja kornika. Obniża ona odporność lasów na szkodniki. Nie jest spowodowana zbyt dużą ilością drzew lub gęstością zalesienia Polski. Powodem są zanikające warunki atmosferyczne. Chodzi o zbyt małe opady deszczu. Proponuję, abyście się zajęli podniesieniem stanu wód gruntowych w lasach, co jest główną przyczyną wysychania i obumierania drzewostanu w naszym kraju. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest złe rozwiązanie, dlatego w międzyczasie złożyłem w imieniu klubu Koalicja Polska wniosek o odrzucenie w drugim czytaniu tego projektu.

Czy dzisiaj, przy spadających cenach energii pochodzącej ze słońca, z wiatru, bo jej produkcja już jest bardzo tania, to jest racjonalne rozwiązanie?

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Panie Ministrze! W uzasadnieniu piszecie, jakie to potężne straty poniosą polskie lasy. Dzisiaj zalega prawie 3 mln

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Skąd pomysł, by wycinkę drzew i spalanie drewna określić energią odnawialną? Przecież OZE właśnie miało to środowisko chronić. W uzasadnieniu oszacowano ilości drewna, które zalega. Ale co z wartością tego drewna? W obliczu katastrofy klimatycznej każde drzewo jest bezcenne. Czy mamy gwarancję, że zostanie spalone tylko nagromadzone drewno? Ile środków trzeba będzie przeznaczyć, by to drewno odzyskać, by te drzewa znów urosły? Bo wiemy, jak długo rośnie las, las rośnie 100 lat. Trochę długo jak na odnawialne źródło energii.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pochodzę z Obornik Wielkopolskich, miejscowości położonej na skraju Puszczy Noteckiej. Ilość połaci objętych w ostatnich kilku latach zrębem, muszę powiedzieć, przeraża nie tylko mnie, ale też wszystkich lubiących las, lubiących korzystać z darów przyrody oferowanych przez ten las.

Organizacje śledzące te dane biją na alarm. Tak nie powinno być. Przestrzegamy dzisiaj, byście nie szli tą drogą. Pan poseł Tomasz Nowak, klub Koalicji Obywatelskiej.

Pogubiliście się zupełnie.

Chcecie się ratować, żeby uniknąć kar z Unii Europejskiej, organizując pseudoodnawialne źródła energii w postaci współspalania.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Polska nie ma szczęścia do ministrów środowiska. Mieliśmy lex Szyszko, teraz mamy lex Woś. Przypominam panu, że jest pan ministrem ochrony środowiska, a nie destrukcji środowiska. Przypominam panu również, że lasy są naszą własnością, a nie pana własnością ani własnością Lasów Państwowych. Lesistość w Polsce wynosi tylko 30%. W Unii Europejskiej średnia lesistość to 38%. Jesteśmy na szarym końcu, jesteśmy na 19. miejscu w Unii Europejskiej. Zadaję panu pytanie: Co pan jako minister ochrony środowiska zrobił i zamierza zrobić, aby lesistość w Polsce wyniosła 38%, czyli średnią w Unii Europejskiej?

Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Muszę powiedzieć, że z rządu wychodzą coraz bardziej absurdalne projekty dotyczące Lasów Państwowych. Najpierw przedstawili państwo Komisji Finansów Publicznych projekt przepisów, który zwalniał z całkowitej odpowiedzialności Lasy Państwowe za odzyskiwanie należności w związku z COVID-19. Widać, że to chyba nie zadziałało. Nie zadziałało, tak? Panie ministrze, to też nie zadziała.

Pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panowie Posłowie! Ta ustawa jest bardzo szkodliwa dla polskich lasów, przyrody i klimatu. Jedynym rzeczywistym celem tej ustawy jest jak najszybsze uzyskanie pieniędzy. Ta sytuacja bulwersuje jeszcze bardziej, kiedy czyta się raport Najwyższej Izby Kontroli, który obnaża niegospodarność Lasów Państwowych. Okazuje się, że tylko 13% swoich wydatków Lasy Państwowe przeznaczają na ochronę i hodowlę lasów oraz utrzymanie zasobów i upraw leśnych, czyli podstawowe cele swojego funkcjonowania. Nie możemy pozwolić, żeby tradycja patrzenia wyłącznie na krótkofalowe zyski monetarne pozwoliła na kontynuację szkodliwych praktyk w lasach.

3 lata temu zezwolili państwo na dewastację Puszczy Białowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Odpowiedzią na kryzys klimatyczny i utratę różnorodności biologicznej nie mogą być działania, które ten kryzys jeszcze bardziej pogłębią poprzez spalanie i uwalnianie dwutlenku węgla. Chcecie umożliwić pod pretekstem cięć sanitarnych spalanie w charakterze biomasy drzew pochodzących z polskich lasów, m.in. w elektrowniach. Nie chodzi wam o żadną ochronę przyrody, tylko o czysty zysk. Wprowadziliście w 2016 r. opłatę za sprzedaż drewna i regularnie doicie Lasy Państwowe z pieniędzy. Dlaczego tak ważny projekt nie został poddany rzetelnym konsultacjom społecznym i opinii ekspertów? Nie palcie polskich lasów. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Jana Szopińskiego, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tryb, w jakim rząd próbuje przeforsować tę ustawę, musi budzić wątpliwości. Ustawa nie powinna być przygotowywana na kolanie. Zmiany powinny być konsultowane z organizacjami pozarządowymi, samorządami i przemysłem meblarskim. Chciałbym zapytać pana ministra, czy są w tej sprawie jakieś przepisy europejskie. Jak obecnie w Polsce ustalane są ceny w przypadku przemysłu meblarskiego? Zaprezentowane w ustawie rozwiązania są szkodliwe zarówno dla przyrody, jak i dla przemysłu meblarskiego. Ta ustawa to pomoc dla monopolisty, a nie dla polskich zakładów przemysłu drzewnego. Chciałbym też zapytać, jaki to będzie miało wpływ na cenę energii elektrycznej. Panie Ministrze! Nie palcie polskich lasów, ratujcie polski przemysł meblarski. Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania panią poseł Małgorzatę Chmiel, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska zobowiązała się, że do 2020 r. będzie wytwarzała 15% energii z odnawialnych źródeł. Szanowni państwo, od 4 lat, odkąd zlikwidowaliście, zniszczyliście wytwarzanie energii odnawialnej z elektrowni wiatrowych, mówię o tym, mówię o tym przy każdej okazji. Nic nie zrobiliście przez 6 lat swoich rządów, żeby zwiększyć ilość produkowanej energii odnawialnej.

Bardzo dziękuję.

Wysoka Izbo! Projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii to dramatyczny pomysł, sprzeczny z celami Unii Europejskiej - osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Premier Mateusz Morawiecki musi go pojutrze przyjąć, jeśli nie chce stracić 8 mld euro dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dlatego też pytam i zachęcam: Dlaczego nie odblokujecie budowy farm wiatrowych, przy postępie technologicznym ich produktywności? Wzmocnijcie wsparcie dla przemysłu meblarskiego, pożytecznego również w kontekście pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla. Dlaczego nie tworzycie korzystnych warunków dla inwestycji w biogazownie, a więc w energetykę rozproszoną? Wspierajcie ideę fotowoltaiki w każdym gospodarstwie domowym.

Bardzo dziękuję. Nie widzę na sali pana posła Michała Szczerby. Zatem stwierdzam, że lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę teraz o zabranie głosu pana Michała Wosia w imieniu ministra środowiska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rozpocznę od podziękowań z całego serca wszystkim aktywistom, którzy wczoraj chcieli się zebrać pod Sejmem, którzy znaleźli czas, którzy poświęcają swój czas, swoje serce ochronie przyrody. Rzeczywiście jest to bardzo wartościowe. Niestety skala kłamstw i manipulacji jest tak gigantyczna, że rzeczywiście także tym, którzy mają dobro polskiej przyrody w sercu, te kłamstwa i manipulacje się udzieliły, zresztą podobnie jak, niestety, zdecydowanej większości posłów i posłanek opozycji. Szanowni państwo, nie kłamcie, proszę, nie kłamcie, zachowajcie resztki rzetelności, zachowajcie resztki zdrowego rozsądku. Wielokrotnie tłumaczyliśmy państwu, że ani jedno drzewo z powodu tej ustawy nie będzie wycięte ponad to, co jest zaplanowane. Ani jedno drzewo nie będzie spalone w polskich elektrowniach w związku z jakimikolwiek wycinkami, o których państwo tyle mówią. Państwo kłamiecie, a kłamiąc, manipulujecie społeczeństwem. Akurat o osoczu ozdrowieńców trochę wiem, bo regularnie je oddaję. Drodzy Państwo! Pytaliście państwo o definicję, gdzie są ci eksperci, którzy tak definiują. Otóż te definicje są wprost w dyrektywie Unii Europejskiej. Wprost w dyrektywie są definicje związane z drewnem energetycznym. Szanowni państwo, Lasy Państwowe, nasze wspólne dobro, tu akurat się zgadzamy, dobro całego społeczeństwa, sadzą w Polsce 500 mln drzew rocznie, co minutę 1 tys. drzew. Skala zalesienia Polski z roku na rok rośnie. Jest coraz więcej drzew i dbamy o to, żeby było coraz więcej drzew, żebyśmy mogli cieszyć nasze oko rozwojem polskiej przyrody.

W czyim interesie jest tak gigantyczne zainteresowanie, z tą skalą kłamstwa i manipulacji?

Skąd jest importowane? Z Czech, z Austrii, ze Wschodu. To jest, proszę państwa, odpowiedź, skąd nagle takie wielkie zainteresowanie i taka skala manipulacji. Otóż, drodzy państwo, informuję państwa, że ani jedno drzewo ponad to, co jest w planach urządzania lasu, nie będzie wycięte. Kto podpisał plan urządzania lasu w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Państwo wiedzą, kto podpisał plan urządzania lasu dla Puszczy Noteckiej? Rząd Platformy i PSL, akurat wiceminister z PSL był za to odpowiedzialny, w 2013 r., i jest realizowany plan urządzania lasu. Otóż ustawa o odnawialnych źródłach energii odnosi się do definicji drewna energetycznego.

Tylko z powodu szkodników i tylko z powodu suszy, która tam panuje. Lasy Państwowe podejmują szereg działań, żeby wzmocnić stan lasów, żeby zwiększyć retencję.

W tym kontekście jeszcze raz państwu powiem, w czyim interesie są te wszystkie krzyki, te kłamstwa i te manipulacje, które tutaj były, drodzy państwo. W czyim interesie? 2,5 mln t biomasy polskie elektrownie importują od Niemców, od Austriaków, od Czechów i ze Wschodu. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Rozpoczniemy niezwłocznie, jak pan minister przybędzie.

Mamy informację, że pan minister będzie dosłownie za minutę, 2 minuty.

Jak widać, pan minister dotarł. Może jeszcze pozwolimy, aby chwilkę odsapnął.

Proszę sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Derę o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ta szczególna data przypomina agresję Związku Sowieckiego na Polskę, co zapoczątkowało okrutne represje wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy znaleźli się.

Jednym z podstawowych instrumentów polityki okupacyjnej władz sowieckich były masowe wywózki Polaków w głąb Związku Radzieckiego, przede wszystkim na Syberię. Polityka ta miała dwa podstawowe cele: eksterminację polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki etniczne. Deportacje zapoczątkowały gehennę kilkuset tysięcy polskich obywateli. Wywózki osób cywilnych, całych rodzin polskich to gehenna pokoleń, które traciły swoich bliskich w drodze na nieludzką ziemię. Męczeński szlak deportowanych zaczynał się już w chwili wejścia NKWD do ich domów, gdy dawano kilkanaście minut na spakowanie się.

Ludzie umierali z zimna, głodu, wyczerpania. Po dotarciu na miejsce zsyłki zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. Konsekwencje zesłań odczuwalne są do dzisiaj, choćby w przypadku żyjących jeszcze ofiar sowieckich prześladowań.

Dotychczasowe rekompensaty udzielane przez państwo polskie z tytułu prześladowań doznanych ze strony okupantów nie objęły wszystkich polskich zesłańców. Celem wniesionego przez pana prezydenta projektu ustawy jest zniwelowanie dotychczasowych nierówności i umożliwienie zaspokojenia słusznych roszczeń polskich obywateli zesłanych lub deportowanych do Związku Radzieckiego w latach 1939–1956, a którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia. Niniejsza inicjatywa opiera się na rozwiązaniach, które zostały przewidziane w projekcie ustawy śp. pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2009 r., inicjatywie ustawodawczej złożonej w Sejmie w 2013 r. przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, a także w prezydenckim projekcie ustawy, który został wniesiony w poprzedniej kadencji, w 2018 r. Proponowana ustawa przewiduje przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji w Związku Radzieckim. Projekt tej ustawy określa zasady przyznawania świadczenia pieniężnego, w tym krąg osób uprawnionych do jego otrzymania, wysokość świadczenia oraz tryb jego przyznania. Świadczenie pieniężne przysługiwać będzie osobom, które posiadały obywatelstwo polskie w chwili zesłania lub deportacji oraz posiadają obywatelstwo polskie w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego. Inicjatywa przewiduje przyznanie świadczenia pieniężnego jednorazowo w wysokości 200 zł za każdy pełen miesiąc okresu podlegającego represjom, jednak nie mniej niż 2400 zł. To świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej złożony do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przyznanie, ustalenie wysokości oraz ewentualna odmowa przyznania świadczenia następować będzie w drodze decyzji administracyjnej szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu. Świadczenie będzie też finansowane, wraz z kosztami jego obsługi, z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Te wypłaty będą wolne od egzekucji oraz nie będą podlegać wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Należy podkreślić, że ten projekt jest odpowiedzią na liczne postulaty otrzymywane przez prezydenta ze środowiska sybiraków, a rozwiązania były konsultowane zarówno z tym środowiskiem, jak i z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

I jeszcze druga prośba - o szybkie uchwalenie tego prawa, ponieważ oni żyją. Już kończę, panie marszałku.

Zdecydowana większość tych, którzy zostali deportowani, po prostu już nie żyje. Zostały tylko dzieci, które chyba, tzn. nie chyba, ale na pewno miały najtrudniejsze dzieciństwo ze wszystkich, którzy żyli w naszym kraju. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Myślę, że Wysoka Izba przychyli się do prośby pana ministra. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić państwu stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, druk nr 452.

Masowe wywózki Polaków w głąb Rosji, przede wszystkim na Syberię i do Kazachstanu, były podstawowym instrumentem polityki okupacyjnej władz sowieckich, których celem była eksterminacja polskich elit politycznych, intelektualnych oraz czystki etniczne.

Rosja - prawny następca Związku Sowieckiego - nigdy nie przyznała się, nie była sądzona i nie wypłaciła odszkodowań za eksterminację setek tysięcy Polaków. Taki stan utrzymuje się od lat, mimo że Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał przymusowe przesiedlenia za zbrodnię. Polska chce wypełnić zobowiązania, których nie wypełniła Rosja. Do chwili obecnej nie została rozwiązana kwestia odszkodowań dla Polaków. Dotychczasowe rekompensaty nie objęły wszystkich polskich zesłańców, dlatego nadrzędnym celem prezydenckiego projektu ustawy jest zniwelowanie występujących nierówności oraz zaspokojenie słusznych roszczeń polskich obywateli, którzy doznali ogromnego cierpienia. Zadośćuczynienie, o którym mówi projekt ustawy, będzie polegać na przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego, a jego wysokość będzie odpowiadać okresowi przebywania na zesłaniu lub deportacji do Związku Radzieckiego.

Jak wskazują dane Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, liczba osób, które mogłyby uzyskać świadczenie, wynosi ok. 22 tys. Z kolei średni czas przebywania na deportacji lub w obozie wynosił 66 miesięcy. Uwzględniając wysokość świadczenia za każdy miesiąc podlegania represjom, o którym mówi projekt ustawy, średnia wysokość świadczenia dla jednej osoby kształtowałaby się na poziomie 13 200 zł. Biorąc pod uwagę, że liczba osób, które skorzystałyby z wprowadzonej ustawy, wynosi ok. 22 tys., obciążenie dla budżetu państwa w związku z wprowadzeniem ustawy nie przekroczy kwoty 300 mln zł. Prezydencki projekt ustawy stanowiący uzupełnienie obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego sybiraków jest ważny ze względów społecznych, ale przede wszystkim godnościowych. Wielu sybiraków, którzy przeżyli to piekło, obecnie żyje w bardzo ubogich warunkach. Są to osoby starsze, najczęściej mocno schorowane. Prezydencki projekt ustawy ma na celu symboliczne uznanie krzywd oraz bólu zesłanych i deportowanych do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przyjęcie projektowanego rozwiązania podkreśli zasługi sybiraków, będzie wsparciem finansowym, ale także próbą zadośćuczynienia osobom zesłanym na Sybir za stracone lata życia. Dziękujemy panu prezydentowi za ten bardzo oczekiwany przez środowiska sybiraków projekt wspierający osoby starsze, które w swoim życiu doświadczyły tak wielkiego cierpienia. W związku z powyższym klub Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie opiniuje przedstawiony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy. Chcę powiedzieć, że posiedzenie komisji, które miało się odbyć dzisiaj, zostało przeniesione na wtorek z uwagi na to, że drugie czytanie odbędzie się w środę. Jestem pełna optymizmu, że zostanie jednogłośnie przyjęty. Bardzo dziękuję. Proszę panią poseł Joannę Frydrych, która przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

Wysoka Izbo!

Proponowane przepisy określają zasady przyznawania zadośćuczynienia, krąg osób uprawnionych do jego otrzymania oraz wysokość i tryb przyznawania świadczenia. Projekt ustawy określa, że będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne. Jego wysokość będzie obliczana na zasadzie proporcjonalności do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji w Związku Radzieckim. Za każdy pełny miesiąc okresu podlegania represjom będzie przysługiwać kwota 200 zł, jednak nie mniej niż 2400 zł. Projekt zakłada, że zadośćuczynienie będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej złożony szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. We wniosku powinno się znaleźć oświadczenie o nieuzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W uzasadnieniu projektu wskazano również, że średni czas przebywania na deportacji lub w obozie w Związku Radzieckim w przypadku sybiraków zamieszkałych na terytorium Polski wynosił 66 miesięcy, a co za tym idzie - średnia wysokość tego świadczenia pieniężnego dla jednej osoby może wynosić 13 200 zł. W uzasadnieniu projektu czytamy, że dotychczasowe rekompensaty udzielane przez państwo polskie z tytułu prześladowań doznanych ze strony okupantów nie objęły wszystkich zesłańców. Czytamy również, że projekt jest odpowiedzią na postulaty środowiska sybiraków, w których sygnalizowano, że dożywają oni swoich dni często w trudnych warunkach. Dlaczego więc tak długo czekacie na uchwalenie tej ustawy? Należy ją jak najszybciej uchwalić, ponieważ sybiracy na nią czekają. Przypomnę, że 13 listopada 2018 r. został złożony projekt ustawy mający na celu wypłatę odszkodowań za zesłanie lub deportację do Związku Radzieckiego. 6 grudnia 2018 r. podczas pierwszego czytania w Sejmie został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak państwo myślicie, co się stało? Utknął, został zamrożony, a w 2018 r. na to świadczenie czekało ok. 24 600 osób.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wejście w życie ustawy przewiduje pozytywny efekt społeczny w postaci długo oczekiwanego zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości. Jak długo osoby zesłane i deportowane do Związku Radzieckiego mają jeszcze czekać? Ten sam projekt ustawy prezydent wniósł tuż przed pierwszą turą wyborów. Czy prawdą jest, że była to wyłącznie oferta wyborcza? Szanowni Państwo! Jeżeli chcecie wypłacić odszkodowania sybirakom, to przejdźmy od razu do drugiego czytania, bez kierowania projektu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Składam taki wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Chcę podkreślić, że Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska będzie głosował za przyjęciem przedmiotowego projektu ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Jacka Czerniaka, który przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Koncepcja zadośćuczynienia w tej formie osobom niesłusznie zesłanym w głąb Związku Radzieckiego za swoją działalność zawodową, społeczną bądź polityczną jest z założenia koncepcją jak najbardziej słuszną.

Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym w tych latach w swoim założeniu miałby tę niesprawiedliwość, w jakimś stopniu oczywiście, zadośćuczynić. Teoretycznie można by bez zastrzeżeń poprzeć ten projekt, gdyż w założeniu jest on bardzo chwalebny, jednakże pojawiają się w nim pewne nieścisłości, a właściwie są do niego uwagi, kwestie, które należało wytłumaczyć i rozstrzygnąć przed głosowaniem za jego przyjęciem. Po pierwsze, mamy już następujące ustawy w tej materii, w systemie polskim są trzy ustawy: ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W tej ustawie znajduje się art. 8, który mówi o odszkodowaniach i zadośćuczynieniu.

Tutaj w art. 3 ust. 1 mówi się o świadczeniach przysługujących w wysokości ustalonej w wyniku podwyższenia wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent. Na podstawie tych przepisów są wypłacane comiesięczne świadczenia pieniężne: dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny, osobom, które z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych przebywały w więzieniach oraz obozach pracy albo na przymusowych zesłaniach w ZSRR. Kolejną kwestią jest szacunkowa liczba osób. Jak podaje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, liczbę tę szacuje się na 22 tys. Dlaczego właściwie - jest pytanie - te osoby nie skorzystały z tych trzech wcześniej wspomnianych ustaw, chociaż w uzasadnieniu jest napisane, w poszczególnych ustawach, jakie z tego tytułu są rekompensaty czy też zadośćuczynienia? Czy ta kwota. Na jakiej podstawie została wyliczona kwota 200 zł za pełny miesiąc i skąd minimum, które wynosi.

W związku z tym mam uwagę i pytanie: Jeżeli osoba nie jest w stanie udokumentować swojego pobytu i deportacji, zgodnie z ustawą o kombatantach ten okres przez kierownika zaliczany jest jako pełny miesiąc. To na jakiej podstawie ta osoba otrzyma.

Oczywiście to nie jest skierowane do pana ministra, ponieważ nie ma on wpływu na proces legislacyjny, ale 5 czy 4 lata VIII kadencji i nie można było tej ustawy przyjąć, to jest drobne, można powiedzieć, nieporozumienie, kieruję to pod adresem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawi pan poseł Mieczysław Kasprzak. Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Myślę, że ustawa jest bardzo ważna i winni jesteśmy tym ludziom jak najszybsze jej uchwalenie. Ale nie szukałbym w tej chwili winnego, bo to już jest kolejny projekt, myślę, że dobrze przygotowany.

Przechodzimy więc do drugiego czytania, panie marszałku, i na tym posiedzeniu załatwiamy temat.

Siedzący tutaj Marek Sawicki - rozmawialiśmy przed chwilą - był akurat posłem wnioskodawcą, przedstawiał ten projekt, uchwaliliśmy to i wszyscy sybiracy dostali to odznaczenie. Wielokrotnie uczestniczyłem w różnych uroczystościach, na których to odznaczenie było wręczane.

Jeżeli słucha się wspomnień tych, którzy.

Kilkadziesiąt dni jechali w tych wagonach bydlęcych. Część z nich nie dojechała na miejsce przeznaczenia, a część zginęła w warunkach ciężkiej pracy. To był dramat tych ludzi. Część wróciła później z armią Andersa czy z armią Wojska Polskiego, I Armią Wojska Polskiego.

Bo powiem państwu, że na każdym ze spotkań jest coraz mniej tych ludzi.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego, który przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja, wraz z panem posłem Grzegorzem Braunem - w drugiej kolejności. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Ponad 1 mln Polaków wywiezionych na nieludzką ziemię w latach 40. ubiegłego wieku i niestety kilkadziesiąt tysięcy tych, którzy doczekują się dzisiejszego dnia.

Cała rodzina babci Bronisławy z województwa wileńskiego - też wywieziona za Ural. Pradziadek Izydor przypłacił to swoim życiem, podobnie jak najstarszy brat dziadka. Dziękujemy za to, że ta inicjatywa się pojawiła.

To jest również bardzo ważne, że państwo polskie dzisiaj przypomina o tragedii górnośląskiej i przeprasza symbolicznie, stara się przeprosić symbolicznie Ślązaków, Polaków za tę krzywdę, jaką komuniści im wyrządzili po II wojnie światowej. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Panie Ministrze!

Szczęść Boże! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jest, chwila ulgi, kwestia dalece niekontrowersyjna tutaj, w Wysokiej Izbie, wprawdzie pustawej nieco, ale przecież nie będzie, mam nadzieję, żywiołowego sporu. Panie Ministrze! Nawet wrzutki w ostatniej chwili, na finiszu kampanii wyborczej, przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, bo rzeczywiście czas najwyższy. Tutaj różne szacunki są podawane, ale to już nie dotyczy ocalonych wraz z rodzinami, to już nie są setki tysięcy, to są dziesiątki tysięcy ocalonych z Sybiru, ocalonych z polskiego Holokaustu. Nie wiem, czy są jeszcze, czy zgłoszą się po to świadczenie ocaleni z białego Oświęcimia - z Kołymy. Dobrze byłoby, żeby następowało otrzeźwienie także w nomenklaturze.

Ci ludzie tam się znaleźli wedle cenzusu narodowościowego i byli przeznaczeni jeśli nie do pospiesznej eksterminacji - chociaż były takie przypadki, prawda, jak sowiecka akcja AB, czyli zbrodnia katyńska (Dzwonek) - to na pewno do eliminacji, eliminacji z życia publicznego, w ogóle z polskiego życia. Mam zatem nadzieję, że to jest rzutem na taśmę próba uczynienia zadość sprawiedliwości dziejowej, ale niech to nie będzie stawianie jakiejś kropki nad i, niech to nie będzie koniec, finał. Nie ciszej nad tą polską trumną Sybiru, tylko głośniej, więcej o tym opowiadajmy. Niech wreszcie wejdzie to do głównego nurtu polskiej świadomości i samoświadomości historycznej. Świeć, Panie, nad duszami tych, którzy stamtąd nie wrócili, i tych, którzy potem latami, ocaliwszy życie, dźwigali tutaj stygmat, byli na marginesie, lękali się opowiedzieć o swojej gehennie.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Do pytań zapisało się trzynaścioro państwa posłów. Proszę jako pierwszego pana posła Tadeusza Tomaszewskiego z klubu Lewica.

Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! To świadczenie od państwa polskiego w pełni tym osobom się należy. Nie ma potrzeby dzisiaj prowadzić sporu, czy to późno, czy za późno, bo każdy rząd, każdy prezydent mógł wcześniej z taką inicjatywą wystąpić.

Chciałbym zapytać przedstawiciela rządu o to, czy kiedykolwiek polski rząd zwracał się do następcy Związku Radzieckiego, czyli państwa rosyjskiego, z wnioskiem o odszkodowania dla obywateli polskich za tę pracę przymusową (Dzwonek), za deportacje do byłego Związku Radzieckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Marka Rutkę, klub Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W owym projekcie świadczenie miało przysługiwać w kwocie 400 zł za każdy miesiąc trwania represji, łącznie - nie więcej niż 30 tys. zł. Tymczasem w projekcie prezydenta Andrzeja Dudy wysokość świadczenia przysługującego za każdy miesiąc wynosi 200 zł. 11 lat temu prezydent Lech Kaczyński pragnął przeznaczyć w ramach zadośćuczynienia zesłańcom kwotę 966 mln zł, zaś 11 lat później prezydent Andrzej Duda - jedynie 290 mln.

Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Po pierwsze, to świadczenie warunkowane jest złożeniem pewnego oświadczenia i dokumentów, jednak nie ma w przepisach proponowanych przez Kancelarię Prezydenta żadnej formuły pomocy osobom represjonowanym w składaniu tego typu oświadczeń. W związku z tym pytanie: Czy to było analizowane? Są to często osoby starsze, schorowane, więc prawdopodobnie taka pomoc będzie potrzebna.

One uderzą w osoby represjonowane, de facto ograniczając być może czy podwyższając pulę środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Pawła Krutula, klub Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szkoda, że tak późno. Wszak prezydent Lech Kaczyński wnosił już taki projekt. Słuszną jest inicjatywą nagrodzenie czy też zadośćuczynienie krzywdom, jeżeli chodzi o wszystkich tych, którzy w wyniku agresji na Polskę byli represjonowani i zsyłani w głąb Związku Radzieckiego. Jak przewiduje ustawodawca, objętych dodatkowym świadczeniem może być nawet 22 tys. osób. Mają one być przyznawane na wniosek repatriantów po spełnieniu swego rodzaju trzech etapów składających się z szeregu skomplikowanych wniosków i zaświadczeń oraz skompletowaniu obszernej dokumentacji. Czy ustawodawca nie może zapewnić tej szczególnie zasłużonej i bardzo wąskiej grupie społecznej komfortu finansowego w postaci dodatkowych świadczeń w prostszej formule, ograniczając wymogi formalne oraz ilość zbędnej dokumentacji, która dla wielu osób starszych będzie dużą barierą, barierą nie do przejścia? Proszę państwa, uchwalmy w końcu tę ustawę, najlepiej na tym posiedzeniu Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Mieczysława Kasprzaka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Panie Marszałku! Kilka takich technicznych spraw. Czy państwo dysponujecie wykazami - wiem, że stowarzyszenia sybiraków posiadają takie wykazy - osób, które kwalifikują się, które ucierpiały wskutek wywózki na Sybir? To jest pierwsza sprawa. Czy w tym momencie są zagwarantowane środki finansowe, żeby dokonać wypłaty? Jeżeli tak, to w jakim terminie, panie ministrze, dokonalibyście tego? Bo to jest sprawa pilna. Dewaluacja następuje pod wieloma względami. Państwo też mówią, jak spada wartość nominalna tego świadczenia. Chodzi o to, żebyśmy nie odkładali tego w czasie i dalej nie dewaluowali, tylko jeszcze w najbliższych miesiącach dokonali wypłaty, ostatecznie obejmując wszystkich, którzy czekają na tego typu zadośćuczynienie. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pani poseł Paulina Matysiak, Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Pomoc sybirakom politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecywali już co najmniej dwukrotnie. Pierwszy projekt, zgłoszony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pochodził z 2009 r., drugi z 2013 r. Oba przewidywały wypłatę 400 zł za każdy miesiąc na zesłaniu. Jednak ustawy głosami posłów koalicji rządzącej PO-PSL przepadły. I powiem państwu, że mnie osobiście cieszy, że po tylu latach pojawiła się troska o sybiraków także wśród parlamentarzystów Platformy i PSL. Teraz, po 5 latach kadencji, Andrzej Duda spełnia swoją obietnicę, chociaż w skromniejszej wersji. I pozostaje pytanie: Dlaczego tyle czasu to trwało? Rządzą państwo 5 lat, projekt ten nie wymaga wielkich nakładów, a może być wielką ulgą, wielkim wsparciem dla tysięcy sybiraków, których od pierwszej obietnicy zmarło już ponad 10 tys. Jeśli chodzi o te zaprezentowane dzisiaj rozwiązania, to naprawdę liczy się każdy dzień. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pani poseł Wanda Nowicka, Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Świadczenia pieniężne dla osób represjonowanych poprzez deportację do Związku Radzieckiego należą się jak mało co mało komu. Jesteśmy tym ludziom to winni. Dlatego warto zadać sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz tym się zajmujemy, skoro każdego dnia osoby represjonowane, sybiracy od nas odchodzą. Można było tę sprawę już dawno załatwić. Czy naprawdę musieliśmy czekać, panie ministrze, na wybory prezydenckie, tak żeby prezydent Duda mógł wykazać się, że zrobił coś dla sybiraków?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu powiedziałem, że popieramy ten projekt ustawy. Mam konkretne pytanie.

Nie mogłaby być większa? Jeszcze raz podkreślam, że żadne pieniądze nie są w stanie temu cierpieniu zadośćuczynić.

Chciałam zapytać rząd, dlaczego od 2018 r. projekt utknął w Sejmie, nie był procedowany - rząd, ponieważ to jest decyzja większości rządowej, państwa z PiS-u.

Należy jak najszybciej uchwalić tę ustawę, bo ci Polacy zasłużyli sobie na tę pomoc, ci Polacy, jak żadni inni, potrzebują tej pomocy i ona im się należy. Pytanie zada pan poseł Edward Siarka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Osoby, które były deportowane, których nigdy do końca nie policzyliśmy, zasługują na to, aby takie świadczenie otrzymać.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Andrzej Grzyb, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Panie Ministrze! Myślę, że sprawa zadośćuczynienia, bo tak to trzeba nazwać, ludziom, którzy przeszli Sybir, nie powinna być przedmiotem sporu. Czy ona by była tydzień wcześniej, czy jest teraz, wydaje mi się, że. Pan poseł Marek Sawicki był wtedy wnioskodawcą w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby to odznaczenie przyznać, ponieważ sybiracy wtedy sami sobie ustanowili krzyż zesłańców.

Wydaje mi się, że ta myśl powinna nam wszystkim tutaj przyświecać. Myślę, że niewiele jest takich spraw, które ponad podziałami możemy w tej Izbie załatwić, dlatego wydaje mi się, że mimo że późno, to ci ludzie zasługują na to. bo przecież są Polacy, którzy byli deportowani do Kazachstanu z tzw. Marchlewszczyzny. Oni też w dalszym ciągu czują się Polakami, a Polskę zachowali, mimo że Polski nie było. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Paweł Szramka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Myślę, że wszyscy, jak jesteśmy na tej sali, uważamy, że jest to projekt potrzebny, i myślę, że również uważamy, że powinien jak najszybciej wejść w życie.

Bardzo proszę się nad tym zastanowić. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pani poseł Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, proszę przekazać panu prezydentowi wielkie podziękowania za ten projekt ustawy.

Powiem tylko tyle: moja ulubiona ciocia Zosieńka nie doczekała.

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W moim mieście co roku oddział Związku Sybiraków zbiera się pod pomnikiem Zesłańców Sybiru, aby w rocznicę pierwszej masowej deportacji oddać honor i pamięć tym, którym okrutny los w sybirskiej tajdze nie dał szans przeżycia i nie wrócili oni na ojczystą ziemię. Dzisiaj mamy uchwalić symboliczną pomoc.

Bardzo uprzejmie proszę przede wszystkim większość parlamentarną o to, aby nasze słowa nie były tylko [[Dzwonek]] słowami, aby dzisiaj przekształciły się w czyny. Pytanie zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panu prezydentowi Dudzie lepiej wychodzą rozmowy z rosyjskimi pranksterami aniżeli realizacja zobowiązań i obietnic. Panie Ministrze!

Komisja Zdrowia odwołuje posiedzenie dotyczące Funduszu Medycznego. Emerytury stażowe są za drogie dla rządu. Polski bon turystyczny będzie, ale nie dla seniorów.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szkoda, że niestety wiele z tych osób nie doczekało tego czasu, kiedy mogłyby zostać tym objęte. To taka nasza moralna odpowiedzialność wobec tych osób. Bardzo dziękuję, że dzisiaj rozmawiamy. Mam nadzieję, że rozmawiamy bez różnic, bo tym ludziom na pewno się to należy. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy również rozmawiali o ludziach, o dzieciach wojny, o których powinniśmy rozmawiać. Być może warto pomyśleć, że ci ludzie, dzisiaj już bardzo sędziwi, potrzebują bardziej rozległej pomocy, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj znaleźliśmy to porozumienie.

Lista posłów zapisanych do pytań została wyczerpana. Proszę teraz o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pana ministra Stanisława Szweda.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za tę inicjatywę dotyczącą bardzo ważnej kwestii społecznej, o której dyskutujemy przez wiele kadencji Sejmu.

Staramy się przez lata wolnej Polski ten system naprawiać, może za wolno, może czasami nieskutecznie, ale myślę, że ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom m.in. Związku Sybiraków i to jest dobra droga, którą zmierzamy.

Nie ma w tej chwili oczywiście jeszcze oficjalnego stanowiska rządu, ale mogę w imieniu naszego ministerstwa przekazać informację, że ten projekt ma poparcie naszego ministerstwa. Chcielibyśmy, aby jednak przepracować go na posiedzeniu komisji z różnych względów, m.in. tych głosów, które dzisiaj padły na posiedzeniu.

Nie ma odniesienia bezpośrednio do tego, że finansowane to będzie ze środków, które będą w ustawie budżetowej zapisane w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym najpierw bardzo serdecznie podziękować za poparcie przez wszystkie kluby parlamentarne tego projektu pana prezydenta Andrzeja Dudy.

Myślę, że w takich sprawach powinniśmy mówić wspólnym głosem, przede wszystkim oddając szacunek tym, którym się to należy. Niestety te piękne słowa zostały zaburzone przez posła Szczerbę. który chyba ma jakąś nienawiść w sercu, bo wszędzie widzi politykę, wszędzie widzi rzeczy, których nie powinien widzieć. Nigdy nie powinien powiedzieć w takiej sprawie, jak powiedział dzisiaj. To są słowa, które nie powinny padać.

Mam nadzieję, że pan poseł jakieś wnioski wyciągnie z tego, co pan w tej chwili słyszy. Każdy ma tę możliwość.

Dzisiaj rozmawiamy tutaj o sybirakach, rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach dla Polski i dla Polaków. Szanowni Państwo! Zacznę może od tego wątku.

Wtedy to świadczenie objęłoby zdecydowanie większą liczbę ludzi.

Tu padły też te słowa, za które dziękuję. Tu nie chodzi o pieniądze, bo nie da się przeliczyć tego cierpienia, tego wszystkiego, co ci ludzie przeszli, na jakąkolwiek złotówkę. Oni mówią: nie o pieniądze tu chodzi.

Rosja nie. Rosja tego w ogóle nie uznaje i żadnych pieniędzy. Polska bierze to tylko dlatego, żeby tym ludziom dać zadośćuczynienie.

I dlatego pan prezydent ten projekt złożył. Szanowni Państwo! 400, 200 zł. Tak się mówi: 200 zł.

Panie marszałku, jeszcze chwilę, bo było trochę tych pytań. Tu był pewien niepokój, że te osoby będą miały trudności w wypełnianiu wniosków. Nie, szanowni państwo, te osoby są zarejestrowane w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oni już to mają. Te osoby są policzone.

I dlatego ten wniosek powinien być złożony, ale to jest najprostszy wniosek, jaki może być.

W ciągu miesiąca zapada decyzja.

Otóż kwestia tego, czy świadczenie dla sybiraków będzie przedmiotem nowej ustawy, czy nowelizacji, w istniejącym już obrocie, jest kwestią wyboru konkretnego rozwiązania legislacyjnego. Myśmy uznali, że w tym momencie, chociażby przez to, że jest to ustawa dedykowana sybirakom, jest to podkreślenie tego, że to nie jest nowelizacja, dodanie gdzieś tam artykułu, wie pani poseł, jak to dokładnie wygląda. Ci ludzie mieliby kłopot, jak to odczytywać, gdybyśmy nowelizowali i dostosowywali te przepisy do istniejących innych ustaw. To jest ustawa dedykowana sybirakom, gdzie jasno i czytelnie jest napisane, co za co im się należy, co otrzymają.

Uważam, że jeżeli to we wtorek będzie na posiedzeniu komisji.

Reasumując, serdecznie dziękuję za wszystkie głosy, za bardzo mądre słowa, które tutaj padły, za głębokie poparcie tego projektu i za to, że wszystkie kluby poparły ten projekt, bo polityka polityką, partie partiami, ale oby nigdy w przyszłości żaden parlament nie rozpatrywał kwestii odszkodowań za jakiekolwiek deportacje, za jakiekolwiek przymusowe przesiedlenia, za jakiekolwiek represje, tylko dlatego że ktoś był Polakiem. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do drugiego czytania niezwłocznie po zakończeniu pierwszego czytania. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 430) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 430.

Postanowienia dyrektywy zmieniającej powinny być implementowane do krajowego porządku prawnego do dnia 30 lipca 2020 r. Na wstępie chciałbym przypomnieć tło prac nad zmianą dyrektywy o delegowaniu pracowników. Należy nadmienić, że w stosunku do tego projektu uruchomiono bardzo rzadko stosowaną w praktyce procedurę tzw. żółtej kartki, w której aż 11 parlamentów krajowych zgłosiło zastrzeżenia. Pomimo tego Komisja utrzymała swoją propozycję. Polska aktywnie uczestniczyła w negocjacjach unijnych, od początku sprzeciwiając się proponowanym zmianom, które w naszej ocenie naruszają zasadę swobody świadczenia usług, a co się z tym wiąże - ograniczają w praktyce możliwość delegowania pracowników.

Pierwsze dwa państwa sprzeciwiły się przyjęciu, pozostałe państwa wstrzymały się od głosu.

W szczególności wnieśliśmy o stwierdzenie nieważności przepisów dyrektywy, które bez wyraźnej poprawy warunków pracy pracowników wprowadzają znaczne utrudnienia w możliwości świadczenia usług i których stosowanie w praktyce może spowodować bardzo duże trudności. Skarga została oparta głównie na zarzucie ograniczenia przez zaskarżoną dyrektywę możliwości swobody świadczenia usług. Do dnia dzisiejszego nie ma niestety rozstrzygnięcia Trybunału w tej sprawie. Wysoka Izbo! Przejdę do zaprezentowania głównych rozwiązań zawartych w ustawie. Projekt zawiera modyfikację przepisów ogólnych w zakresie definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracodawcy delegującego pracownika z terytorium naszego kraju w zakresie dotyczącym delegowania pracowników tymczasowych. Należy podkreślić, że istotne zmiany w procedowanym projekcie ustawy dotyczą modyfikacji warunków zatrudnienia zapewnianym pracownikom delegowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co jest związane zwłaszcza z uzależnieniem zakresu ochrony pracowników od długości delegowania. Wyjaśniam: obecnie pracodawca delegujący pracownika na terytorium naszego kraju musi zapewnić pracownikowi delegowanemu określony ustawą zamknięty katalog warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż wynikające z Kodeksu pracy oraz z innych przepisów prawa pracy, które obejmują m.in. minimalne wynagrodzenie za pracę. Przedkładany projekt rozszerza ten obowiązek o konieczność zapewnienia takiemu pracownikowi pełnego, a nie tylko minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to konieczność wypłaty wynagrodzenia wraz ze wszystkimi jego obligatoryjnymi składnikami. Nowe przepisy nie ograniczają czasu delegowania pracowników do Polski, natomiast rozszerzają katalog warunków zatrudnienia, które trzeba zapewnić pracownikom delegowanym w przypadku wydłużenia okresu delegowania. Pracownik delegowany do Polski na okres do 12 miesięcy powinien mieć zapewniony zamknięty katalog warunków zatrudnienia. Po upływie 12 miesięcy pracodawca będzie mógł złożyć wniosek o przedłużenie stosowania zamkniętego katalogu o kolejne 6 miesięcy. Dopiero po tym okresie będzie musiał stosować wobec pracownika delegowanego co do zasady wszystkie warunki zatrudnienia wynikające z polskiego prawa.

Przedmiotowy projekt modyfikuje również zadania Państwowej Inspekcji Pracy, która już obecnie realizuje szereg zadań związanych z delegowaniem pracowników. Można tutaj przykładowo podać rozszerzenie zadań o charakterze informacyjnym, rozszerzenie w zakresie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z właściwymi organami innych państw członkowskich. Umożliwi on też występowanie Państwowej Inspekcji Pracy do pracodawcy delegującego pracownika z terytorium naszego kraju, do przedsiębiorcy, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów państwa członkowskiego.

Bardzo dziękuję panu ministrowi. Lista mówców w tym punkcie przedstawia się następująco. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Sylwester Tułajew, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

W opinii Komisji inicjatywa ta miała w szczególności na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego. Dodatkowo projekt ma na celu zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych, z akt podatkowych i tych, które są objęte tajemnicą skarbową. Ustawa składa się z siedmiu artykułów.

Szczegółowy opis proponowanych zmian jest przedstawiony w uzasadnieniu projektu ustawy. Rząd proponuje 17 zmian, które dotyczą przede wszystkim modyfikacji definicji, wprowadzają bardzo obszerne i bardzo potrzebne modyfikacje minimalnych warunków zatrudnienia, wprowadzają 12-miesięczny okres gwarancji stosowania minimalnych warunków zatrudnienia, wprowadzają również możliwość złożenia umotywowanego powiadomienia, rozszerzają poziom gwarancji warunków zatrudnienia w przypadku niezłożenia umotywowanego powiadomienia do upływu okresu 12 miesięcy delegowania lub gdy okres delegowania przekroczy 18 miesięcy w przypadku złożenia ww. powiadomienia. Wprowadza szereg różnych istotnych zmian, m.in. tę, o której wspomniałem, czyli modyfikacje zadań Państwowej Inspekcji Pracy, modyfikuje również uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadza przepisy karne, wprowadza zmiany redakcyjne. Jest propozycja dodania do Ordynacji podatkowej w art. 299 w § 3 ustawy pkt 15a, zgodnie z którym informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem niektórych wymienionych w tym przepisie informacji, udostępniane będą również organom Państwowej Pracy w zakresie niezbędnym do realizacji jej ustawowych zadań.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę o przyjęcie tego projektu ustawy i wyrażam pozytywne stanowisko w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Mariusz Witczak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest ważna ustawa. To jest ważna ustawa, dlatego że ona dotyczy w najszerszym ujęciu polskiej gospodarki, rynku pracy w Polsce i rozwoju wielu polskich przedsiębiorców, którzy zapraszają współpracowników na terytorium RP, zaprzyjaźnionych firm czy kooperantów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak jak pan minister powiedział, wdrożone przepisy tej dyrektywy muszą wejść w życie do końca lipca. Trzeba pamiętać o tym, że ta ustawa została napisana dla przedsiębiorców, a nie dla urzędników, a skoro dla przedsiębiorców, to powinna być dużo wcześniej przygotowana, przedsiębiorcy powinni mieć dużo więcej czasu na to, żeby się zapoznać z zasadami funkcjonowania tej ustawy, a tego czasu mieć nie będą. Niewypełnienie wymogów, które państwo nakładacie na przedsiębiorców, na firmy czy na pracowników delegowanych na własny rachunek czy przez oddziały, firmy państw członkowskich Unii Europejskiej, niewykonanie tych zapisów ustawy będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami prawnymi czy skarbowymi. Zatem z tego punktu widzenia należy państwa bardzo głęboko krytykować za to, że na ostatnią chwilę przygotowaliście tę ustawę. Ja muszę też powiedzieć, że skoro jest to ustawa dla przedsiębiorców, to powinna być przygotowana w sposób przejrzysty i komunikatywny. Zresztą zasady demokratycznego państwa prawnego wywodzone są z zasady prawidłowej legislacji. Natomiast rozmaite pojęcia, przepisy, które państwo formułujecie, nie mają charakteru jasnego i precyzyjnego. Ja tylko zwrócę państwu uwagę na dwie rzeczy. Tak naprawdę, jeśli precyzyjnie przeczyta się tę ustawę, nie ma się świadomości, o prawie którego państwa mówicie - czy państwa, które deleguje pracowników na terytorium RP, czy polskiego. Ja oczywiście rozumiem, jaka była intencja państwa przy pisaniu tej ustawy, ale to jest poważny kłopot. Przedsiębiorca będzie musiał radzić się poważnych kancelarii prawnych, żeby wiedzieć, jak dokładnie zinterpretować tę ustawę, i to jest wysoce naganne. Kolejny problem. Z przepisów projektu jasno wynika, że nie obejmujecie jego zakresem kwestii dotyczących transportu drogowego, ale mówicie o tym w uzasadnieniu. A przecież przedsiębiorca nie będzie czytał uzasadnienia, skoro nie zawarliście tych kwestii w sposób precyzyjny w tekście ustawy.

Już nie mówiąc o tym, a powtórzę to jeszcze raz, że przygotowaliście to w ostatniej chwili, co jest absolutnie naganne. Szanowni Państwo! Warto jeszcze przy tej okazji przypomnieć, że złożyliście państwo jakiś czas temu skargę do Trybunału. O tym też pan minister wspominał.

Prawda jest też taka, że skargę do TSUE przygotowaliście w sposób kiepski, powiem wprost, bo została ta skarga bardzo skrytykowana i prawdopodobnie nie będzie z tego tytułu żadnego skutku. Co do zasady dyrektywy jako państwo członkowskie przyjmujemy. Jeszcze moment i ta ustawa byłaby przeterminowana, zatem oczywiście należy tę ustawę doprecyzować, uczynić bardziej komunikatywną i przyjąć. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Macieja Koniecznego, który przedstawi stanowisko klubu Lewica. Wysoka Izbo! To jest dobry dzień dla Polski, bo robimy krok w stronę solidarnej Europy. Co prawda na ostatnią chwilę i ewidentnie wbrew woli zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej, ale robimy ten krok i to jest dobry krok. W świecie, któremu grozi kryzys klimatyczny, gospodarczy, szalejące nierówności, wciąż rosnąca potęga wielkich korporacji, silna, spójna i solidarna Europa to jest dokładnie to, czego potrzebujemy, bo żaden kraj samodzielnie sobie z wyzwaniami przyszłości nie poradzi. Kwestia pracowników delegowanych budzi ogromne emocje w całej Europie, bo dotyka sedna tego, jaka ta Europa ma być - czy Europa ma być jedynie wolnym rynkiem rządzonym bezwzględną, bezduszną zasadą zysku, czy może - i tego chciałaby Lewica - powinna być oparta na zasadach solidarności i współpracy i gwarantować, że każda Europejka i każdy Europejczyk będą mogli liczyć na uczciwą płacę i godne warunki życia. Dyskusja na temat pracowników delegowanych przez lata budziła takie emocje, bo to jest także dyskusja o tym, w czyim interesie będzie urządzona Europa. Chodzi o to, czy Europa będzie urządzona w interesie wielkich korporacji zalewających Brukselę armią lobbystów, czy Europa będzie urządzona w interesie pracującej większości, Europejek i Europejczyków, którzy żyjąc od pierwszego do pierwszego tak naprawdę ten kontynent utrzymują. Wielkie korporacje zrobią wszystko, wykorzystają każdy przepis, każdą lukę prawną, żeby płacić jak najmniej, omijać prawo pracy i unikać opodatkowania. Naszą odpowiedzią musi być właśnie solidarna Europa, która równa w górę, a nie w dół. Zmiana ustawy o delegowaniu pracowników - to brzmi bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę sprawa jest prosta. Chodzi o to, żeby pracownik, którego firma deleguje do pracy w innym kraju, mógł liczyć na takie same minimalne warunki płacy i pracy, jakie obowiązują pracowników w danym kraju. Brzmi uczciwie? Dla nas tak, ale zarówno Platforma, jak i PiS w Parlamencie Europejskim głosowały przeciwko tej zasadzie. Głosowały tak, bo chcą konkurować tanimi kosztami pracy, czyli chcą konkurować tym, że Polacy są tani, można płacić im mniej i gorzej ich traktować. Tyle, jeżeli chodzi o wstawanie z kolan. Lewica mówi jasno: polski pracownik nie może zarabiać mniej i być traktowany gorzej niż Francuz, Niemiec i Czech pracujący u jego boku. Mówimy coś więcej: brak solidarności i równanie do dołu na dłuższą metę nikomu w Europie się nie opłaca. Słaby to pomysł na rozwój kraju. Ale przyjmijmy, że tak jest, że prawica wygrała i Europa dalej rządzona jest przez wolnorynkowy dogmatyzm. Polscy pracownicy są tańsi i konkurują z nimi Niemcy, Francuzi. Na cholerę mi taka Europa, żaden to dla mnie interes. I stąd, z tej konkurencji do dołu właśnie biorą się napięcia, które rozsadzają Unię Europejską. Czy tego naprawdę chcemy? To zresztą nie wszystko. Załóżmy przez chwilę, że konkurowanie niskimi płacami się Polsce opłaca, tzn. panu premierowi się opłaca, firmom się opłaca, bo pracownikom to już niekoniecznie. Ale załóżmy, że tak jest. Otóż Holandii, Irlandii i Luksemburgowi opłaca się, żeby korporacje robiące biznesy w Polsce płaciły podatki u nich. Pan premier Morawiecki z tym walczy, i bardzo dobrze, że walczy z rajami podatkowymi w Europie. Ja mu w tej walce kibicuję, bo chcę, żeby wielkie korporacje uczciwie płaciły podatki w Polsce. Ale mam takie pytanie: Czy my możemy skutecznie upominać się o solidarność w kwestii podatkowej, jeżeli sami nie wykazujemy solidarności w kwestii pracowniczej? Oczywiście, że nie. Lewica jest za solidarną Europą, solidarną, czyli taką, w której umawiamy się, że pracownikowi nie można płacić mniej i traktować go gorzej dlatego, że przyjechał z innego kraju. Ale to nie wszystko. Chcemy Europy, w której obowiązuje płaca minimalna, poniżej której nie można zapłacić nikomu w żadnym kraju. Chcemy solidarnej Europy, w której korporacje uczciwie płacą podatki, bo nie ma rajów podatkowych, nie ma tych krajów-cwaniaków, które dorabiają się kosztem innych. Tylko taka Europa, solidarna i silna, jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości. Jednak idee to jedno, a wykonanie - drugie. Ta ustawa faktycznie jest niedopracowana, wymaga zmian i dlatego przedstawimy poprawki Lewicy, które zagwarantują, że to równe traktowanie pracowników nie pozostanie tylko na papierze. Po pierwsze, ustawa nakłada nowe obowiązki na i tak już skrajnie niedofinansowaną Państwową Inspekcję Pracy. Złożymy poprawki, które to naprawią, które to finansowanie zapewnią. Druga rzecz.

Dlatego będziemy składać poprawkę, która będzie sprawiała, że te kary będą proporcjonalne do realnej skali działalności firmy. Pan poseł Dariusz Klimczak przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo!

Historia tej dyrektywy jest dłuższa, ponieważ już raz kraje Unii Europejskiej planowały wprowadzić powyższe zmiany w przepisach, lecz wówczas pozycja Polski była na tyle silna, że obroniliśmy nasze firmy, dysponując tzw. mniejszością blokującą. Ministrem pracy i polityki społecznej w tym czasie był Władysław Kosiniak-Kamysz. To on rozmawiał w tej sprawie z liderami europejskich krajów. Pamiętam dokładnie, jak jeszcze w listopadzie 2013 r. Inicjatywa Mobilności Pracy, Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy, Polska Izba Handlu, Polskie Forum HR oraz Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia wyrażały głębokie zaniepokojenie kierunkiem prac nad projektem dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dlaczego tym razem to się nie udało? Przecież według propagandy Prawa i Sprawiedliwości Polska dopiero teraz zaczyna się liczyć w Europie. Jak się w takim razie liczy, skoro nowe unijne prawo to przede wszystkim bat na polskich przedsiębiorców, na polskie firmy? Dlatego warto przypomnieć tak ważny dla Polski i całej Unii Europejskiej kompromis osiągnięty w dyrektywie z 2014 r., po 2-letnich, bardzo trudnych negocjacjach, w których dużą skutecznością wykazał się minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednym z celów tamtego kompromisu było kluczowe dla tej sprawy zagwarantowanie przestrzegania praw pracowniczych. Nowa dyrektywa nie tylko regulowała kwestie monitorowania przestrzegania przepisów i współpracy administracyjnej, ale także nakładała obowiązki na państwa członkowskie w zakresie przejrzystości informowania o warunkach zatrudnienia i istniejących obowiązkach. Nigdy nie było naszej zgody na to, by pod szyldem ochrony praw pracowniczych i uczciwej konkurencji budować nowe mury w Europie. Dotychczas udawało nam się skutecznie przekonywać, że mobilność jest dla Unii szansą, a nie zagrożeniem - do czasu, kiedy stery rządów w Polsce objęło Prawo i Sprawiedliwość. Warto podkreślić, że Polska jest unijnym liderem w zakresie delegowania pracowników. Obrazuje to choćby liczba wydanych poświadczeń A1, czyli dokumentów określających, któremu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczenia społecznego podlega pracownik. Według najnowszych danych spośród prawie 3 mln wydanych poświadczeń na polskie firmy przypada ich ponad 605 tys., a więc to prawie 30% wszystkich wydanych dla pracowników delegowanych w obrębie całej Unii Europejskiej. Niestety inne kraje Unii Europejskiej, szczególnie tej tzw. starej Unii, inaczej postrzegają polską mobilność, nazywając to zjawiskiem dumpingu socjalnego, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ nasi pracownicy wypełniają w rzeczywistości lukę kompetencyjną, szczególnie w takich krajach jak Francja, Niemcy czy nawet Belgia. Co czeka naszych przedsiębiorców?

Każdy z przedsiębiorców, który zamierza kontynuować działalność, a raczej wyjścia nie ma, musi, po pierwsze, błyskawicznie zorientować się co do elementów charakterystycznych dla danego państwa przyjmującego, jeżeli chodzi o składowe wynagrodzenia, po drugie, trzeba będzie szczegółowo pilnować tzw. obliczeń w kwestii kumulatywnych okresów delegowania. Nowa dyrektywa wprowadza maksymalny okres delegowania, podczas gdy wcześniej tego typu określeń nie było. Wszystkiego tego można byłoby uniknąć, gdyby nasz rząd liczył się w Unii Europejskiej. Przykład tej dyrektywy pokazuje jak na dłoni, że rząd PiS ma dobrą pozycję w Europie, ale tylko wtedy, kiedy podają to „Wiadomości” TVP. Taka jest niestety smutna prawda. Nowe prawo ma według mnie i polskich przedsiębiorców charakter protekcjonistyczny i dyskryminacyjny w stosunku do naszego kraju. Obawiam się, że to może doprowadzić co najmniej do ogromnych strat dla 15 tys. polskich firm, a w konsekwencji do upadku wielu z nich, a co najmniej utraty przez pracowników miejsc pracy. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Krystiana Kamińskiego, który przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw to właśnie implementacja tejże dyrektywy unijnej, dyrektywy, o której wszyscy wiemy, że jest wyjątkowo niekorzystna dla Polski, a właściwie dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, której beneficjentem będą kraje Europy Zachodniej, dyrektywy, która w sposób jaskrawy przeczy zasadzie swobody świadczenia usług i przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej. Spójrzmy więc na to, jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie tej dyrektywy dla polskich firm delegujących, co nowego czeka polskich przedsiębiorców z powodu słabości Polski na arenie międzynarodowej. I tak: ograniczenie delegowania zasadniczo do 12 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach - do 18. Delegowanie długoterminowe oraz delegowanie stacjonarne, przy którym występuje zastępstwo, będzie de facto zabronione. Nastąpi praktyczny zakaz delegowania w branżach stacjonarnych: produkcja, logistyka, opieka i inne branże, w których usługi wykonywane są przez wiele miesięcy i lat w tym samym miejscu. Czekają nas nowe restrykcje i uciążliwe oraz kosztowne wymogi formalne. Nastąpi kategoryczny zakaz delegowania przez firmy nieprowadzące znacznej działalności krajowej zgodnie z działalnością eksportową. Nastąpi kategoryczny zakaz delegowania pracowników, którzy na terenie Polski nie świadczą zazwyczaj pracy. Nowe przepisy przewidują tzw. kontrole krzyżowe, czyli szerokie badanie przez zagraniczne instytucje i przez ZUS zdolności firmy do delegowania oraz zdolności pracowników do bycia delegowanymi. Kolejne kontrole ZUS-owskie - świetny pomysł, na pewno wszyscy się ucieszą. Ale dalej: po wejściu w życie nowych przepisów znacząco wzrosną wynagrodzenia pracowników delegowanych. Polskie firmy będą obciążone wyższymi kosztami z tytułu innych należności przysługujących zgodnie z przepisami krajów, do których delegowani są pracownicy. Ale to nie wszystko. Odpowiednie modyfikacje będą także obowiązywały wkrótce w zakresie poświadczenia A1. Większość polskich firm delegujących nie uzyska już formularzy A1 i nie będą one mogły delegować pracowników za granicę. W nowych przepisach zakłada się ograniczoną ważność dokumentu A1, ekspresowe weryfikowanie i uchylanie poświadczeń formularzy A1 przez ZUS i przez zagraniczne instytucje, a także automatyczną i błyskawiczną egzekucję zagranicznych składek. Czy Polska naprawdę jest tak małym państwem unijnym, że nasze zdanie, że nasze interesy nie mają dla reszty żadnego znaczenia? Wprowadzenie tej dyrektywy to ograniczenie swobody świadczenia usług i przepływu pracowników zagwarantowanej w traktatach Unii Europejskiej oraz działanie, którego głównym motywem jest właśnie zlikwidowanie przewagi konkurencyjnej Polski. Polacy to ok. 20% z ok. 3 mln delegowanych w Unii Europejskiej, czyli największa grupa narodowa. Delegowaniem zajmuje się w Polsce ok. 90 tys. firm - ogromny rynek, bardzo dużo polskich przedsiębiorców, którzy bez jakiejkolwiek pomocy zbudowali wielki biznes i sprowadzili miliardy złotych do Polski. W czyim interesie jest ta dyrektywa? Oczywiście w interesie Niemiec i Francji. Firmy delegujące, czyli polskie, przeniosą siedziby właśnie do tych państw albo się rozwiążą, a pracownicy będą zatrudnieni w Niemczech lub we Francji.

I to wszystko dzieje się w czasach kryzysu. Tego już niestety nie zatrzymamy. Nowe zasady dotyczące delegowania nie obowiązują na razie transportu drogowego, w dyrektywie zrobiono bowiem wyjątek od tego, ale wszyscy wiemy, że niedługo w życie wejdzie tzw. pakiet mobilności. To oznacza, że również nasz transport międzynarodowy bardzo mocno na tym straci. Walkę, aby zatrzymać dekret o delegowaniu pracowników, przegraliście, to mówię do rządu, z kretesem. Nie byliście w stanie obronić polskiego biznesu opierającego się na delegowaniu pracowników przed unijnymi ograniczeniami. Postarajcie się obronić chociaż nasz transport. W przeciwnym razie Polska, polscy przedsiębiorcy stracą na tych wszystkich sztucznych ograniczeniach, a wy będziecie za to odpowiedzialni, ponieważ nie stworzyliście odpowiedniej koalicji, aby temu zapobiec. I w tym wypadku Wuj Sam wam nie pomoże. Sami musicie zbudować dobre stosunki z innymi państwami Unii Europejskiej, aby mieć możliwość stworzenia koalicji, która uwzględni nasze polskie interesy.

Dziękuję bardzo. Przystępujemy do pytań.

Panie Ministrze! Klasyka gatunku partii rządzącej w postaci wrzucania w ostatniej chwili ustaw niezwykle ważnych dla pracodawców, przedsiębiorców, pracowników. Mieliście 2 lata, panie ministrze, na zaimplementowanie dyrektywy unijnej. Tak traktujecie przedsiębiorców. Tak ważna ustawa trzymana 2 lata, a dzisiaj jeden przedstawiciel rządu. Moje pytanie do pana ministra: Co będzie w momencie, kiedy tak skomplikowane zapisy ustawy nie zostaną na czas wdrożone przez przedsiębiorców? Czy tak wspieracie polską przedsiębiorczość (Dzwonek) i pracowników, że wrzucacie w ostatniej chwili, na 15 dni przed upływem terminu, niezwykle ważną ustawę, z której mogą skorzystać tysiące polskich pracowników i tysiące polskich firm? Dla mnie jako byłego przedsiębiorcy to jest po prostu skandal. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze!

Co prawda możliwe jest odstąpienie, gdyby było jakieś specjalne uzasadnienie.

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Dariusz Klimczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Mam pytanie. W uzasadnieniu do tej ustawy dowiadujemy się bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie: Państwowa Pracy obecnie napotyka bardzo duże trudności w pozyskiwaniu informacji od organów skarbowych na temat obrotów przedsiębiorcy, dlatego inspektorzy pracy mają mieć dostęp do dokumentów objętych tajemnicą skarbową. Mam pytanie o bardzo marną argumentację tego zapisu. Mianowicie chciałbym zapytać: Dlaczego projektodawca zmian nie wyjaśnił, w jaki sposób wiedza o obrotach pracodawcy delegującego pracownika ma pomóc w ustaleniu legalności zatrudnienia pracownika delegowanego? Pytanie zada pan poseł Robert Kwiatkowski, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Pierwsze dotyczy terminarza. Wszyscy już solidarnie, że tak powiem, skrytykowaliśmy rząd za opóźnienie. Nie będę wnikał w to, jakie są jego przyczyny, natomiast domniemywam, że w związku z tym, że państwo obsunęliście się, jeśli chodzi o harmonogram, to macie już przepisy wykonawcze do tej ustawy. Jeśli tak, to czy można by się z nimi ewentualnie zapoznać? Wiemy, że ta ustawa, podobnie jak ta dyrektywa, kabotażu nie dotyczy, ale w uzasadnieniu do ustawy znaleźliśmy informację, że toczone są prace regulujące sprawę kabotażu na gruncie prawodawstwa polskiego. Kto prowadzi te prace i na jakim one są etapie? Poproszę także o tę informację. Po trzecie wreszcie, chciałem zapytać o strategię negocjacyjną i prawną, zarówno jeśli chodzi o (Dzwonek) tę dyrektywę, jak i dyrektywę dotyczącą mobilności oraz skargi, jaką rząd polski złożył w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy istnieje jakiś zespół, który koordynuje kompleks tych problemów, czy też nie? Dziękuję bardzo. Pytanie zada pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Będziemy dziś deliberować także nad tym, czy mamy zaufanie do ministrów Ziobry i Kamińskiego. To pytam: Co robi polski rząd, by chronić polskich pracowników przed bandytami, którzy udając pośredników, kierują do niewolniczej pracy za granicą? Od lat Polacy pracują w ubojniach, na polach, na budowach, kierowani tam także przez pseudoagencje pracy. Czy ktoś się tym zajmuje?

Dlaczego to Niemcy ścigają naszych łobuzów, a nie panowie Ziobro i Kamiński? Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Mirosława Suchonia, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pewne wątpliwości dotyczące pracowników delegowanych, myślę, że każdy pracownik chciałby chyba być delegowany do zarządu partii Razem. Tam są rzeczywiście bardzo, powiedziałbym, godne zarobki. Pewnie rzeczywiście wielu pracowników delegowanych, ale także zwykłych polskich pracowników nie zarabia tyle, ile właśnie w tej najbardziej, powiedziałbym, lewicowej partii. To jest dosyć ciekawe. Oczywiście ta dyrektywa jest absolutnie protekcjonistyczna. Wszyscy możemy ubolewać nad tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w sposób beznadziejny po prostu przegrał tę walkę, zajął się rzeczami zupełnie pobocznymi, nie traktując poważnie interesów polskich firm i polskich pracowników. To jest bardzo wielkie zaniedbanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ten fragment dotyczy delegowania do Polski, ale mam pytanie do pana ministra dotyczące rosnących praktyk protekcjonistycznych stosowanych przez inne państwa w całej Europie. Co takiego zrobił rząd, żeby zatrzymać [[Dzwonek]] te praktyki, które w ostatnim czasie bardzo silnie uderzają w polskie firmy, zwłaszcza w branżę transportową? Wszyscy widzimy, że to się dzieje, a rząd milczy, skazując nasze firmy i pracowników tam pracujących po prostu na wyparcie z rynków zagranicznych. Pytanie zada pan poseł Paweł Krutul, Lewica. Wysoka Izbo! Ustawodawca wprowadza zmiany dotyczące delegowania pracowników, w nowym artykule zobowiązuje pracodawcę do składania swego rodzaju oświadczeń, zobowiązań. Czy ustawodawca planuje wydać stosowny druk, szablon, oświadczenie, które ułatwi pracodawcom spełnienie wymogów formalnych?

Jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, żeby to było jasne i klarowne. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania panią poseł Paulinę Matysiak, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie Posłowie! W ostatnim czasie głośno było o aroganckiej odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jaką dostały polskie opiekunki osób starszych pracujące w Niemczech. Szacuje się, że ok. 200 tys. opiekunek pracuje w Niemczech na czarno, dlatego poprosiły one polski rząd o podjęcie rozmów ze stroną niemiecką w celu objęcia ich niemiecką ochroną prawną. Że mają radzić sobie same, bo są w dobrej pozycji negocjacyjnej i jest wiele ofert pracy. Ministerstwo się zreflektowało i dzień później wysłało inną odpowiedź, ale z pewnością takie traktowanie Polek i Polaków, którzy proszą o pomoc, jest skandalem. Przyjęcie ustawy, o której dzisiaj dyskutujemy, jest konieczne i potrzebne. Jednak biorąc pod uwagę takie działania ministerstwa, obawiam się, że pozostanie ona martwym prawem. Dlatego mam pytania: Czy rządzący mają zamiar stawać po stronie polskich pracowników (Dzwonek) i po stronie polskich opiekunek? Czy każda polska opiekunka może być pewna, że wkrótce będzie traktowana tak samo jak jej niemiecka koleżanka? Czy może być pewna, że będzie miała pracę etatową i takie same stawki jak jej niemieckie koleżanki? Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Otóż mam takie pytanie: Czy była możliwość wprowadzenia do tej ustawy jednak zapisów, które dotyczyłyby warunków zamieszkania delegowanych pracowników? Media niejednokrotnie informowały o przypadkach naszych obywateli, którzy zamieszkiwali w różnego typu miejscach, w których na pewno nie były przestrzegane normy w zakresie zamieszkania, o których moglibyśmy powiedzieć, że lokale te nie były lokalami mieszkalnymi i nijak się miały do określenia, że są to lokale mieszkalne. Pytanie drugie. Otóż były 2 lata na przygotowanie tej ustawy. W związku z tym mam pytanie, gdzie są akty wykonawcze do tej ustawy. Nie dlatego pytam, że dobrą praktyką uchwałodawczą powinno być to, że te akty wykonawcze powinny nam tu dzisiaj towarzyszyć, tylko że o to po prostu pytają pracodawcy. Bo tam są różnego typu zapisy, których trzeba będzie przestrzegać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Krzysztof Bosak, koło Konfederacja.

Panie Marszałku! Szanowni Posłowie! Rząd po przegranej walce w Unii Europejskiej nie starał się odroczyć tej niekorzystnej dla nas dyrektywy. A przecież mógł. Są sytuacje, w których zalegamy latami z wdrożeniem dyrektyw, akurat w tych obszarach, w których Unia Europejska, o dziwo, ma bardziej liberalne prawo niż nasze państwo. To np. dyrektywa o handlu i posiadaniu broni. W tej chwili polskie prawo jest bardziej opresyjne, a w tajemnicy w ministerstwie jest szykowany podobno jeszcze bardziej opresyjny projekt. Państwowa Inspekcja Pracy dostanie nowe obowiązki. Będzie umożliwiony transfer danych. Nasze służby, nasi podatnicy sami będą finansowali opresje wobec polskich przedsiębiorców, wobec polskich firm, po to żeby zagraniczne firmy, które przestraszyły się polskiej konkurencji, mogły łatwiej ją wykończyć. Niemcy i Francja, które same zabiegały o tę dyrektywę, nie wdrożyły jej. Polscy przedsiębiorcy nie wiedzą, co będzie po 30 lipca, a grozić im mogą podwójne kontrole [[Dzwonek]] ze strony i zagranicznych, i naszych inspekcji. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Najwyższy czas i ostatni dzwonek, żeby ta ustawa, tak ważna z punktu widzenia pracowników delegowanych, została przyjęta. Słuchając dzisiaj dyskusji na sali, mogłam odnieść wrażenie, że tak naprawdę ta ustawa służy po to, żeby szykanować i prześladować przedsiębiorców, a nie po to, żeby wspomóc pracowników, tych pracowników polskich, którzy wciąż jeszcze są traktowani jak pracownicy drugiej czy trzeciej kategorii po blisko 20 latach bycia częścią Unii Europejskiej. A zatem trzeba było wreszcie wprowadzić takie ustawodawstwo, dzięki któremu pracownicy mogą być traktowani na równi z pracownikami w innych krajach Unii Europejskiej. Pytanie, jakie mam, dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy.

Czy ministerstwo nie przewiduje wzmocnienia instrumentów dla Państwowej Inspekcji Pracy w taki sposób, żeby inspekcja mogła również proaktywnie monitorować, jak ta ustawa jest przestrzegana, w szczególności z perspektywy pracowników wykonujących pracę tymczasową, którzy są szczególnie dyskryminowani? Teraz pytanie zada pan poseł Killion Munyama, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zauważam, że dyrektywa musi być przyjęta właśnie w krajach członkowskich do 30 lipca, czyli za 15 dni. Stąd pytanie: Dlaczego akurat dopiero w ostatniej chwili po prostu dyskutujemy nad tym projektem? Co się stanie w momencie, kiedy akurat tej dyrektywy nie uda się nam przyjąć?

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Roberta Winnickiego, Konfederacja.

Wysoka Izbo! Zdrowo rozumiana ochrona praw pracowniczych w XXI w. to oczywiście pewien standard cywilizacyjny, ale to, co państwo tutaj, zwłaszcza ze strony Lewicy, proponują i do czego nawołują, to po prostu nic innego jak eurokomunizm. To jest po prostu realne urzeczywistnienie eurokomuny. Oczywiście jest to eurokomunizm taki za 200 tys. na rok, państwo z zarządu partii Razem, wiemy o tym już z oświadczeń majątkowych. Natomiast mam pytanie do przedstawicieli rządu. Jest niestety rażąca nieskuteczność w zabieganiu o polskie interesy na forum Unii Europejskiej. Wiemy, że Unia Europejska jest forum starcia tak naprawdę interesów narodowych. Niemcy prą do realizacji swoich interesów, jeśli chodzi o usługi transportowe, prą w przypadku Nord Streamu i w innych przypadkach. Skończmy wreszcie z tą frazeologią (Dzwonek) jakichś wspólnych interesów i zacznijmy mówić otwartym tekstem, o co toczy się gra w Brukseli, w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. I jeszcze pytanie zada pan poseł Dobromir Sośnierz z koła Konfederacja. Ja mam taką propozycję, żeby państwo z lewej i z prawej strony przestali się za każdym razem przerzucać odpowiedzialnością za to, że przegraliśmy w Unii kolejne głosowania, bo przegrywamy tam wszystkie od lat. Nie ma przykładów odwrotnych. Ja też tam byłem, gorycz porażki piłem, widziałem posłów Platformy Obywatelskiej bezsilnie protestujących, proszących o powtórzenie głosowania, w którym się pomylili z powodu nadmiernego tempa narzuconego przez przewodniczącego, i nawet takiego gestu grzecznościowego nie mogli się doprosić. W Unii Europejskiej bawimy się w wolny rynek zawsze tylko wtedy, tylko do tego momentu, do którego opłaca się to Niemcom i Francuzom. Jak przestaje się opłacać, kiedy okazuje się, że oni nie umieją znaleźć się na wolnym rynku, kiedy przegrywają na wolnym rynku, to mówią: A, zaraz, zaraz, tak się nie będziemy bawić, tutaj musimy sobie wdrożyć jakieś regulacje. Ubolewam nad tym, że rząd polski nie dość, że bierze na siebie rolę nakładającego kaganiec na własnych obywateli, to jeszcze okazuje się w tym tak gorliwy, bo mam wrażenie, że moglibyśmy tę dyrektywę nie tylko wdrażać później, ale i w sposób nieco bardziej dziurawy, żeby nie być aż tak gorliwym strażnikiem kagańca nakładanego na własnych obywateli. Głos teraz zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan Stanisław Szwed. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyrektywa faktycznie jest skomplikowana. Ona zupełnie czego innego dotyczy.

W drugą stronę, tak, faktycznie, jeśli chodzi o delegowanie polskich pracowników, ponad 648 tys. do krajów Unii Europejskiej, ale w naszą stronę jest zupełnie inaczej.

Negocjacje prowadził pan minister Mleczko z PSL-u. To jest początek tego, o czym dzisiaj mówimy. Dyrektywa wdrożeniowa została wdrożona za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ważną kwestią przy tej dyrektywie zmieniającej jest to, że w pierwszym okresie udało nam się wprowadzić tzw. procedurę żółtej kartki, czyli 11 państw, które były przeciwne tym wdrożeniom, ale dalej też nie mieliśmy wsparcia.

O tym mówił były eurodeputowany pan poseł Sośnierz. Jeśli chodzi o terminy, to projekt został przygotowany na koniec ubiegłego roku.

Jednym z powodów tego, że ten temat był trochę dłużej procedowany, było to, że czekaliśmy na rozstrzygnięcie trybunału europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości.

Jeśli chodzi o państwa, które dzisiaj są też na etapie wdrożenia, to są Belgia, Czechy, Francja, Malta, Litwa, Słowacja i Niemcy, czyli te państwa mają wdrożoną w tej chwili dyrektywę. Austria, Dania i Finlandia są na podobnym etapie jak my, czyli też w tej chwili. Padały pytania o Państwową Inspekcję Pracy.

Jeśli chodzi o kwestię związaną z tymi decyzjami, które wynikają z decyzji Trybunału Sprawiedliwości, ten prace koordynuje KPRM, pan minister Szymański, jego przedstawiciel bezpośrednio uczestniczy w posiedzeniach Trybunału Sprawiedliwości, reprezentując nasz kraj.

Liczymy, że ta procedura będzie szybko przebiegać i że jeszcze uda się to na następnym posiedzeniu Sejmu przyjąć. Dziękuję bardzo. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 430, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 420 i 451) Proszę teraz pana posła Marka Asta o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, druki nr 420 i 451.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 18 czerwca i 8 lipca 2020 r. wnosi: Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. Jednocześnie komisja zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu przedstawia na żądanie wnioskodawców trzy wnioski mniejszości zgłoszone przez klub Lewicy, które nie zyskały akceptacji komisji. Warto jednak podkreślić, że komisja w uzgodnieniu z wnioskodawcami i stroną rządową zaakceptowała trzy inne wnioski Lewicy, co pokazuje, że projekt był procedowany ponad partyjnymi podziałami, co daje naprawdę dużą satysfakcję. Komisja nad projektem, tak jak już wspomniałem, pracowała na dwóch posiedzeniach. Rzeczywiście projekt zyskał poparcie praktycznie wszystkich klubów Wysokiej Izby, więc to bardzo dobrze rokuje dla funkcjonowania tej ustawy. Wobec powyższego w imieniu komisji wnoszę jak na wstępie. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Marek Ast w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu co do sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Myślę, że po tym procedowaniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka warto przypomnieć główne założenia tego projektu właśnie z uwagi na to, że pierwsze czytanie odbywało się nie tutaj, na sali plenarnej, tylko w komisji. Projekt, o czym już jako sprawozdawca komisji wspominałem, ma poparcie rzeczywiście szerokie, jeżeli chodzi o wszystkie strony zasiadające w Sejmie. Wynika to z tego, że on powstał w celu zapewnienia sprawniejszego działania komisji na rzecz realizacji jej ustawowych zadań. Analiza przepisów ustawy doprowadziła wnioskodawców do przekonania, że jest jednak uzasadnione na tym etapie wprowadzenie zmian legislacyjnych, które będą przeciwdziałały przewlekłości postępowań toczących się przed komisją oraz służyły zwiększeniu zaufania obywateli do komisji. Główne kierunki zmian, które zostały zaproponowane, dotyczyły udzielenia pełnomocnictwa, chodzi o adwokata lub radcę prawnego, do reprezentowania komisji czy poszerzenia dotychczasowego katalogu przesłanek będących podstawą do nałożenia obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia. Ponadto w celu usprawnienia i przyspieszenia procedury przyznawania przez komisję na rzecz pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich odszkodowań oraz zadośćuczynień zaproponowano również w przedmiotowym projekcie regulację, zgodnie z którą sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom nieruchomości warszawskich. Z uwagi na wyłączenie możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez miasto stołeczne Warszawę logiczną konsekwencją takiego kierunku zmian legislacyjnych jest przyjęcie, że zaskarżone decyzje w trybie dotychczasowych przepisów przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie uważa się za ostateczne i prawomocne, zaś odszkodowanie oraz zadośćuczynienie zostaną wypłacone uprawnionym osobom w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy. Te zmiany, te propozycje spotkały się ze zdecydowanym poparciem ze strony stowarzyszeń lokatorskich. To pokazuje, że zmiany idą w dobrym kierunku i zasługują na poparcie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem dzisiaj procedowanej ustawy. Teraz w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska pan poseł Michał Szczerba. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po 5 latach rządów PiS Warszawa i inne miasta czekają na dużą ustawę reprywatyzacyjną, ustawę, która była obiecana, a której założenia 3 lata temu na konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości przedstawiał Patryk Jaki z panem dr. Zaradkiewiczem. Minęły 3 lata, ustawy dużej jak nie było, tak nie ma. Wysoka Izbo! Cały czas jedyną ustawą, która zadziałała, ustawą, która nie wyczerpuje potrzeb miasta stołecznego Warszawy, jest mała ustawa reprywatyzacyjna. Ale gdy była uchwalana, PiS wstrzymał się od głosu. Chroni ona dzisiaj instytucje kultury, szkoły, parki, obiekty sportowe. Ta nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych zaproponowana przez Klub Parlamentarny PiS to próba naprawiania własnych błędów. Od początku mówiliśmy, jakie to są błędy. Mówiliśmy, że ustawa o komisji weryfikacyjnej była pisana pospiesznie i na kolanie. Jej celem nie było wcale powołanie instytucji, która rozwiąże kompleksowo problemy dzikiej reprywatyzacji i naprawi krzywdy lokatorów. Chodziło o coś innego. Widzieliśmy to doskonale w kampanii warszawskiej Patryka Jakiego. Wtedy temat komisji weryfikacyjnej, temat reprywatyzacji stał się jakby dla PiS-u mniej istotny. Szanowni Państwo! Co jest w tej sprawie najważniejsze? W tej sprawie najważniejsze są kompleksowe rozwiązania, żeby nigdy więcej nie dochodziło do krzywd ludzkich, do dramatów, do tragedii. Nie może być tak, że pisane na kolanie ustawy, pospiesznie, bez refleksji powodują tylko kłopoty i chaos prawny. Ta ustawa już raz była nowelizowana. Teraz jest nowelizowana po raz drugi. Tę złą ustawę trzeba oczywiście naprawić. Obietnica wypłaty odszkodowań była bez pokrycia, a one są potrzebne. Trzeba tę sprawę załatwić. Takie od dawna było stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej, takie było stanowisko prezydenta Warszawy i warszawskiego ratusza. Dlatego jeszcze w poprzedniej kadencji złożyliśmy projekt osobnej ustawy o odszkodowaniach dla każdego lokatora, któremu pomoc się należała, a nie otrzymał jej, a nie tylko dla tych, których wybierze sobie sama komisja. Ale PiS ten projekt odrzucił. Również miasto Warszawa od roku wskazywało, jak tę ustawę trzeba poprawić, żeby można było wypłacać odszkodowania. Uchwalenie proponowanych teraz zmian otwiera drogę do ich wypłaty przynajmniej dla części osób. Ale to nie zmienia faktu, że to w ogóle nie załatwia sprawy. To tylko mały krok odsuwający w czasie konieczność zmierzenia się z największymi problemami. Projekt nie rozwiązuje problemów związanych z roszczeniami dawnych właścicieli nieruchomości przejętych na mocy dekretu o reformie rolnej, ustawy o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej czy wielu innych obowiązujących do 1989 r. W dalszym ciągu polskie miasta zmagają się ze skutkami eliminowania z obrotu prawnego starych decyzji stanowiących podstawę nabycia gruntów przez Skarb Państwa. Problem reprywatyzacji dotyczy całej Polski, a propozycje PiS dotyczą wyłącznie problemów wybranej grupy warszawskich lokatorów, bez szerszego spojrzenia na problem, z którym zmagają się w szczególności duże miasta w kraju. Wysoka Izbo! Bez rozwiązań systemowych, kompleksowych, znajdujących równowagę pomiędzy prawami byłych właścicieli, interesem miast, prawem lokatorów a wartościami społecznymi ta ustawa będzie wyłącznie kolejną małą ustawą. Gdzie zatem jest obiecana duża ustawa, o której mówimy od 5 lat, a która była obiecana 3 lata temu? Bez niej duch reprywatyzacji nadal będzie straszył i będzie ona jak smok, któremu odcina się kolejne głowy, a na ich miejscu ciągle wyrastają nowe. Klub Koalicji Obywatelskiej popiera projekt, ale wymaga on przyjęcia kilku zmian i doprecyzowania części zapisów, aby zapewnić trwałość i pewność orzeczeń reprywatyzacyjnych, które będą skarżone przez dawnych właścicieli do sądów administracyjnych. Na konieczność tych zmian wskazuje również Prokuratoria Generalna. Nie mogą znaleźć poparcia zapisy, które de facto pozbawiają byłych właścicieli jakichkolwiek praw do zwrotu utraconego mienia bez jakiejkolwiek rekompensaty. Uregulowania wymaga też kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Skarbu Państwa. Przyjęcie zaproponowanych przepisów bez zmian wskazanych przez miasto (Dzwonek) naraża miasto na znaczną odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz dawnych właścicieli nieruchomości. Popierając ten projekt ustawy, składamy poprawki do tego projektu. Tych poprawek jest 13.

Proszę, teraz pani poseł Magdalena Biejat w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy. Wysoka Izbo! Dom jest miejscem, do którego wracamy zmęczeni, by odpocząć, w którym spędzamy czas z rodziną. To fundament równowagi w innych obszarach życia: zawodowym, zdrowotnym, rodzinnym. Posiadanie domu, własnego miejsca, w którym możemy się schronić i zregenerować, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i obywatela. Ta potrzeba znajduje swoje odzwierciedlenie w polskiej konstytucji. Art. 75 mówi: władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Ochronę praw lokatorów określa ustawa. Niestety, od 30 lat kolejne ekipy rządzące nie wywiązywały się należycie z tego konstytucyjnego obowiązku. Podstawowe potrzeby tysięcy lokatorów, polskich obywateli okazywały się mniej ważne od interesów właścicieli, osób z roszczeniami. Były tak mało istotne dla urzędników, sędziów, biznesmenów zajmujących się reprywatyzacją, że nie dokładano starań, aby dokumenty należycie sprawdzić, potwierdzić ich autentyczność, odszukać faktycznych spadkobierców lub stwierdzić ich brak. Kwitły przestępcze procedery i korupcja, a lokatorzy byli bestialsko nękani przez firmy wyspecjalizowane w czyszczeniu kamienic. Postępowania reprywatyzacyjne toczyły się ponad głowami skazanych na niepewność mieszkańców, którym odmawiano prawa do wglądu w dokumentacje czy choćby rzetelnej informacji co do zaawansowania procesu reprywatyzacyjnego, a co za tym idzie - do informacji o ich sytuacji i ich przyszłości. W efekcie lokatorzy - często osoby starsze, z niepełnosprawnościami, niezamożne - latami żyli w niepewności i stresie. Przez 30 lat lokatorzy kamienic oraz władze samorządowe prosili o uregulowanie kwestii roszczeń reprywatyzacyjnych, o stworzenie systemowych rozwiązań, które zagwarantowałyby cywilizowane, humanitarne rozstrzygnięcia w sporze pomiędzy prawami mieszkaniowymi obywateli a prawem własności. Po dzikiej reprywatyzacji, która w szczególnym stopniu dotknęła Warszawę, apelowali o sprawiedliwość i jak dotąd jej nie otrzymali. To problem Krakowa, to problem Poznania, Lublina i innych miast. Wnioski reprywatyzacyjne pojawiają się także na wsiach.

W rzeczywistości problem reprywatyzacji dotyka więc milionów Polek i Polaków. Zarówno mała ustawa reprywatyzacyjna, jak i komisja reprywatyzacyjna nie rozwiązały skutecznie problemów natury prawnej, nie zakończyły dramatów ponad 100 tys. ludzi bezpośrednio dotkniętych problemem roszczeń. Szacuje się, że komisja reprywatyzacyjna, która zajmuje się jedynie sprawami warszawskimi, musiałaby pracować do 2050 r., aby zweryfikować wszystkie 4 tys. postępowań toczących się w stolicy. Wadą dotychczasowych rozwiązań, źródłem ich nieskuteczności jest przede wszystkim ich niekompletność. Poszczególne rozwiązania obejmują jedynie wycinek problemu, skupiają się tylko na stolicy i nie uwzględniają wszystkich kategorii reprywatyzowanych nieruchomości ze względu na sposób ich przejęcia przez państwo. Nowelizacja, o której dziś rozmawiamy, po raz kolejny jedynie koryguje z gruntu wadliwe i nieskuteczne przepisy. Lewica zagłosuje za jej przyjęciem. Doceniamy dobre intencje. Poprzemy każde rozwiązanie, które choć w niewielkim stopniu poprawi sytuację obywateli.

Część z tych poprawek została przyjęta w czasie prac komisji, a dziś zgłaszamy kolejne. Liczymy na ich poparcie przez obóz rządzący i przez opozycję. Ale Lewica nie zamierza na tym poprzestać. Zawsze broniliśmy i będziemy bronić podstawowego, konstytucyjnego prawa obywateli do bezpieczeństwa mieszkalnego. Broniliśmy lokatorów przed eksmisjami, byliśmy z nimi podczas ulicznych demonstracji, a dziś bronimy ich praw i zabiegamy o sprawiedliwość dla nich tutaj, w Sejmie.

Doceniamy dobre intencje obozu rządzącego oraz podjęcie trudnego tematu reprywatyzacji.

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania komisji sprawiedliwości o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dla ścisłości, projekt jest opatrzony drukami nr 420 i 451. W omawianym projekcie zaproponowano regulację, zgodnie z którą sprzeciw wobec decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom nieruchomości warszawskich.

Oznacza to, że przyznane na ich podstawie odszkodowania oraz zadośćuczynienia miałyby zostać wypłacone uprawnionym osobom w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ww. przepisów.

Projekt zakłada również odmowę reprywatyzacji na rzecz osoby, która nabyła prawo lub roszczenie od kuratora spadku lub kuratora ustanowionego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, jeżeli nie było podstaw do jego ustanowienia.

Natomiast w imieniu Koalicji Polskiej, jeśli chodzi o ten projekt, deklaruję wolę (Dzwonek) udziału w dalszych pracach nad nim. Pan poseł Grzegorz Braun w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kilka spraw naraz, w telegraficznym skrócie. Nie żadna reprywatyzacja, tylko po prostu zwrot mienia zagrabionego. Albo jest prawo własności, albo go nie ma. Lewica nigdy nie przestanie nas zadziwiać swoją inwencją językową. Bezpieczeństwo mieszkaniowe. My przebijamy to i mówimy: sprawiedliwość dziejowa mieszkaniowa. Przebijamy i mówimy: sprawdzam. Popieramy rzecz jasna wszystkie działania, które zmierzają do zwrócenia tego, co się komu należy, ale zrobiliście do tego taką specustawę, tak jak kolega to przed chwilą stwierdził, wycinkowe rozwiązywanie problemu, m.st. Warszawa, pod publikę działania komisji. Chcielibyśmy uniknąć tej fikcji. Bardzo proszę w dalszej pracy wziąć tę poprawkę pod uwagę. Poseł Konrad Berkowicz, koło Konfederacja. Szanowni Państwo! Przewodniczący Ast przed chwilą powiedział, że doszło do porozumienia ponad partyjnymi podziałami, i rzeczywiście partyjne podziały zostały przezwyciężone przez wspólnotę idei. A ideą, która połączyła m.in. Prawo i Sprawiedliwość ze zjednoczoną Lewicą, jest idea socjalistyczna. Prawo własności - święte dla każdego konserwatysty, oczywiste dla każdego wolnościowca - ma według członków komisji zostać wyrzucone na śmietnik.

A więc tradycyjne, naturalne prawo własności ma być zastąpione nowotworem ideologicznym, wykwitem rewolucji komunistycznej. Ja rozumiem, że mieć gdzie mieszkać to jest ważna sprawa, ale dlatego rząd powinien przestać przeszkadzać się bogacić, przestać przeszkadzać biurokracją, wysokimi podatkami i przestać dawać sygnał ludziom, że nie warto się bogacić, bo w każdej chwili majątek, który zgromadzą, w imię tej idei komunistycznej mogą stracić na rzecz tych, którzy się wzbogacili mniej, żeby było równo. Ja powiedziałem tu mocne słowa, bo rzeczywiście twierdzę, że jesteście komunistami, czy to bezbożnymi, [[Wesołość na sali]] czy to z krzyżem w zębach - jesteście komunistami. To jest kontrowersyjne stwierdzenie, więc podeprę się waszym autorytetem. Słowa premiera Morawieckiego sprzed kilku miesięcy brzmią: Możemy sobie tak szczerze powiedzieć: ta myśl, robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Na to można odpowiedzieć tylko słowami Czesława Miłosza: „Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, / nie zajrzeli do dupy - tam miałem socjalizm”

Całe szczęście obyło się bez. O czym my tutaj dzisiaj mówimy? Mówimy o negatywnych skutkach ogromnego problemu, a państwo te negatywne skutki chcą łatać jakimiś wyborczymi komisjami, które powstały na użytek kampanii wyborczej samorządowej w Warszawie, a nie patrzą państwo na źródło problemu. Co jest źródłem problemu? Oczywiście komunizm, który zagrabił prywatne mienie, doprowadził do tego, że gros nieruchomości, tysiące nieruchomości w Polsce, nie mając swojego właściciela, niszczeją i w zasadzie niedługo nie będą miały wartości. Oczywiście na tym zyskały mafie poprzez różne przekręty, ale głównym winowajcą są te wszystkie ugrupowania zasiadające w Sejmie, poza Konfederacją, które przez lata nie doprowadziły do uchwalenia w Polsce ustawy reprywatyzacyjnej czy ustawy Polska jest jedynym krajem w bloku postkomunistycznym, w którym nie uchwalono takiej ustawy. Ostatnia taka ustawa została zablokowana przez prezydenta Kwaśniewskiego. Szanowni Państwo! Ja bym chciał, żebyśmy wreszcie zlikwidowali problem nieuregulowanego stosunku własnościowego i przystąpili do prac może nie nad ustawą reprywatyzacyjną, ale przynajmniej nad ustawą o odszkodowaniach, ustawą, która także ureguluje stosunek własnościowy, bo państwo zrzucili to na sądy. Sądy działają tak, jak działają, mamy problemy wtórne, które państwo chcą teraz łatać kolejnymi regulacjami, kolejnym zagmatwaniem. Mamy kolejną nowelizację tej ustawy o komisji, a komisja ma też kolejne problemy, bo państwo np. wyłączają kolejne przesłanki zwrotu nieruchomości, także wykraczają poza warunek dotyczący nieruchomości, która ma służyć użyteczności publicznej. My na to się nie godzimy. Uważamy, że jeżeli chcemy, rozwiązać problem i też sprawić, by własność w Polsce miała właściciela, a nie niszczała [[Dzwonek]] nie była niszczona przez brak nadzoru właścicielskiego, trzeba uchwalić odpowiednią ustawę. Jako pierwsza pani poseł Hanna Gill-Piątek, klub Lewicy. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wybrzmiał głos oprawców, teraz może coś głosem pokrzywdzonych. Targowa 47 - grzywna dla lokatorów za transparent w obronie ich praw. Kilińskiego 89 - kamienica, którą podpalili tzw. nieznani sprawcy, razem z lokatorami w środku. Odcinanie wody, niszczenie klatek - tak dziś wygląda rzeczywistość w przypadku lokatorów w reprywatyzowanych kamienicach w Łodzi, a problem dotyczy miast w całej Polsce. Kupcy roszczeń i mafia reprywatyzacyjna mają się doskonale, bo ani PO, ani PiS nie zależało przez lata, aby ten problem rozwiązać, czego przykładem jest przedstawiany projekt. To ponad 100 procesów dotyczących 300 nieruchomości, w których opieramy się nawet na Kodeksie Napoleona. W tym czasie PiS woli lansować się w nieskutecznej komisji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa to z pewnością krok w dobrą stronę, gdyż ograniczy to patologię reprywatyzacji. Pozbywanie się z kamienic lokatorów jest jednym z najbardziej haniebnych epizodów w naszej najnowszej historii. Żałuję jednak, że nie wykorzystano tej okazji do podjęcia jeszcze bardziej skutecznych działań. Zaproponowane przepisy nie określają jednoznacznie sposobu wyceny nieruchomości, co oznacza, że wciąż utrzymany może zostać reprywatyzacyjny biznes. W związku z tym chciałbym zapytać, jakie działania zamierza podjąć rząd, żeby rekompensaty za nieruchomości były naliczane od wartości w dniu nacjonalizacji, a nie wartości obecnej. To byłaby prawdziwa zmiana, która doprowadziłaby do zakończenia tej haniebnej procedury. Po drugie, problem nie dotyczy tylko Warszawy. Kiedy możemy się spodziewać rozwiązań także dla innych miast, dla Poznania, Wrocławia itd. Z tego miejsca dziękuję Beacie Siemieniako, Katarzynie Czarnociej, wszystkim innym, którzy walczą o prawa lokatorów. To dzięki wam ta ustawa jest dzisiaj procedowana.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa, o której dyskutujemy, to nie jest ustawa reprywatyzacyjna, tylko ustawa odszkodowawcza dla lokatorów warszawskich. Odszkodowania to ważne kwestie, ale niewystarczające i nie można uciekać od tego problemu, jeśli chodzi o resztę kraju. Sprawy związane z własnością gruntów czy kamienic w całej Polsce należy raz na zawsze uregulować i nie może być tak, że jedynie decyzje administracyjne i wyroki sądowe rozstrzygają te kwestie. Nie może również być tak, że nie bierze się pod uwagę zasiedzenia, przedawnienia roszczeń czy nakładów na nieruchomości przy rozliczaniu z właścicielami. Problemem jest również brak właściwych wpisów do ksiąg wieczystych, co miało miejsce np. w Gliwicach, gdzie spadkobiercy właścicieli gruntów rolnych odsprzedali swoje ziemie biznesmenowi jako grunt rolny, mimo że wiedzieli, że to nie jest grunt rolny. Gmina musiała to odkupić za wiele milionów złotych, co obciążyło mieszkańców miasta. Na Śląsku z roszczeniami ciągle (Dzwonek) występują właściciele kamienic i gruntów.

Wysoka Izbo! W ustawie przyznają państwo dodatkowe uprawnienia komisji, którą wcześniej kierował Patryk Jaki, ale nie ma podstaw prawnych do tego, by te przyznane przywileje miały moc prawną. Brak podstaw prawnych do przydzielania odszkodowań, szacowania obowiązujących kwot do zwrotu lub wywłaszczenia. O ile trzeba było już dawno stworzyć dużą ustawę reprywatyzacyjną, i to jest oczywiste, o tyle teraz nie ma powodów do dawania kolejnych martwych w świetle prawa kompetencji komisji, która będzie służyła do atakowania przeciwników politycznych. Dlaczego ustawodawca świadomie uchwala słabej jakości prawo i przyznaje komisji przywileje, które nie mają żadnych podstaw i umocowania prawnego? Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, klub Lewicy.

Wysoka Izbo! Niniejsze przedłożenie w części nawiązuje również do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w której odnajdziemy katalog celów publicznych, a wśród nich odnajdziemy budowę i utrzymanie dróg, lotnisk, budynków dla organów władzy, sądownictwa czy szkolnictwa, opiekę nad zabytkami i pomnikami, ale nie znajdziemy tego, co powinno być równie ważne, jeśli nie najważniejsze, czyli zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób przez zarządzających publicznym zasobem mieszkaniowym. Lewica złożyła stosowną poprawkę, która tę lukę wypełnia. Niestety, została ona odrzucona w trakcie prac komisji.

Wysoki Sejmie! Mam dwie uwagi i jedno pytanie. Pierwsza uwaga. Trzeba mieć świadomość, że po wojnie wielu właścicieli, również spadkobierców, po prostu nie żyło.

Druga uwaga. Doceniam fakt, iż znajduje się w tej ustawie zapis, który rozszerza nieco kompetencje, by odbierać i nakładać odpowiednie kary na spółki córki handlarzy roszczeń.

Bo my to traktujemy. Patrzę na to trochę jak na wywieszenie białej flagi wobec mafii reprywatyzacyjnej.

Wysoka Izbo! To jest bardzo ważny i potrzebny projekt ustawy. Jeden z tych projektów, które pomimo że były tak potrzebne, kazały na siebie czekać ponad 20 lat. Chcę jednak zwrócić uwagę na jedną prostą sprawę. Choć komisja weryfikacyjna zasadniczo zazwyczaj staje po stronie lokatorów, to sami lokatorzy w postępowaniach przed komisją mają jednak ograniczoną podmiotowość. Można by to zmienić, gdyby na wniosek lokatorów przewodniczący komisji mógł dopuścić ich do udziału w postępowaniu na prawach strony. I tu pytanie: Czy ewentualnie możemy liczyć na poparcie takiej poprawki? Ona po prostu bardzo ułatwiłaby sytuację lokatorom i byłaby dowodem na to, że traktujemy ich jako stronę, bo de facto w tych postępowaniach powinni mieć taki status. Dziękuję. Pani poseł Karolina Pawliczak, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niniejsza ustawa pozwoli oczywiście zabezpieczyć prawa lokatorów i faktycznie przerwać dziką reprywatyzację nieruchomości wraz z jej lokatorami. Ten fakt oczywiście cieszy, choć ta ustawa nie jest wolna od ułomności. Pytam bowiem: Co z resztą kraju? Warszawa to przecież nie wszystko. W moim rodzinnym Kaliszu taki sam los spotkał kilkadziesiąt kamienic i ich lokatorów. Mamy te same problemy. Proces czyścicieli kamienic kosztem uboższej części społeczeństwa trwa bowiem od lat i dotyczy wielu miast w naszym kraju. Lewica złoży kompleksowy projekt ustawy, przedstawiliśmy już publicznie jej wstępne założenia i mam nadzieję, że spotka się to z taką samą życzliwością. O tę życzliwość i wsparcie będziemy zabiegać. Dużo słyszeliśmy tutaj o świętym prawie własności, ale jeśli spojrzymy chociażby na historię Warszawy i przyjrzymy się konkretom, to zobaczymy, że to jest historia, w której miasto było w gruzach, ludzie pracą społeczną i własnym wysiłkiem odbudowali kamienice, mieszkali w nich i po kilkudziesięciu latach przychodzi jakiś cwaniak i chce im tę kamienicę zabrać. Dla mnie to jest święte prawo złodziejstwa, a nie święte prawo własności. Czas, żeby w końcu prawo do złodziejstwa przestało być święte. Dlatego potrzebujemy dużej ustawy reprywatyzacyjnej, i Lewica ją złoży.

Panie Ministrze! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Powstrzymanie zwrotów nieruchomości zamieszkałych przez lokatorów w naturze powinno być priorytetem i tutaj projekt ustawy wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Natomiast odmowa zwrotu nieuchronnie wiąże się z koniecznością wypłacenia odszkodowania. Te odszkodowania są dzisiaj często zawyżone. Nieruchomości przejęte w 1945 r. często były kupą gruzów, i to kupą gruzów z zadłużeniem. Na tych gruntach odbudowano budynki, dokonano oddłużenia, ich wartość znacząco wzrosła. I tutaj pytanie: Czy Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę przyjęcia takich zapisów, które urealnią wycenę nieruchomości, tak by odpowiadała ona stanowi, w jakim nieruchomości rzeczywiście znajdowały się po II wojnie światowej? Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przy okazji procedowania nad tym punktem obrad chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inną niesprawiedliwość, dotyczącą tzw. polityki mieszkaniowej, a mianowicie dotyczącą Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Wielu lokatorów mieszkań zakładowych zarządzanych przez tę spółkę od nawet kilkunastu lat zabiega o wykup swoich mieszkań zgodnie z ustawą. Mieszkańcy, którzy do tej pory żyją w budynkach od lat nieremontowanych, zwykle płacąc wysoki czynsz, chcą wreszcie sami zadbać o siebie, tworząc wspólnoty, aby ich warunki mieszkaniowe i życiowe uległy znaczącej poprawie. Niestety spółka, zapewniając w kolejnych pismach, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najemców, postępuje w tej sprawie zbyt powoli, robi za mało. Dlatego chciałbym zapytać: Kiedy rząd zamierza zająć się tą kwestią, która również narusza zasady sprawiedliwości społecznej? Wysoka Izbo! Chciałbym kontynuować myśl rozpoczętą przez przewodniczącego Asta. Dziękuję za wyjątkowo dobrą atmosferę podczas pracy w komisji. Od Lewicy, przez Platformę, po Prawo i Sprawiedliwość mamy tę świadomość dziejową, że ta ustawa jest potrzebna. Nie słuchamy pohukiwań społecznych darwinistów z Konfederacji i pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami. Lewica proponowała i będzie proponować - i będziemy za tym obstawać - aby do ustawy wpisać jak najszerszy katalog sytuacji, na podstawie których będzie można składać wnioski o zadośćuczynienie i odszkodowanie, ponieważ katalog tych sytuacji, stosowany przez tych, którzy chcą odzyskiwać w sposób nielegalny kamienice, jest bardzo duży. Te sytuacje są obrzydliwe i ohydne - zastraszanie, dokwaterowywanie lokatorów, zajmowanie lokali. Te sytuacje trzeba wpisać do katalogu przesłanek, na podstawie których lokatorzy, mieszkańcy będą mogli [[Dzwonek]] wnosić te wnioski. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy prawdą jest, że w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, a więc pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydenta Marcina Święcickiego, pana Pawła Piskorskiego, na ogólną liczbę 4200 decyzji zwrotowych ponad 80% to decyzje właśnie tej trójki prezydentów, a więc pani prezydent Waltz, panów Piskorskiego i Święcickiego? Czy prawdą jest, że komisja zbadała ponad 3 tys. decyzji, wykazując że m.st.

Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście sprawa reprywatyzacji stała się sprawą bardzo polityczną.

Prawda jest taka, że ten problem nie dotyczy tylko Warszawy, ale również innych miast w Polsce. Kolejne pytanie to kwestia zapisu w tej ustawie, dotyczącego tego, że sprzeciwy, które dzisiaj złożyło miasto Warszawa, wobec tych decyzji, które już zostały wydane, mówiąc krótko, są tą ustawą odrzucane, w związku z czym decyzje w tej sprawie stają się prawomocne.

Wysoka Izbo! Panie ministrze, moje pytanie dotyczy innych miast. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy na temat pierwotnego projektu ustawy, to oczywiście zgłaszaliśmy szereg wątpliwości. Pamiętam też, że wnosiliśmy czy informowaliśmy, że tego rodzaju, różnego rodzaju wydarzenia spójne z tym, co miało miejsce w Warszawie, mają miejsce i w innych miastach w Polsce. Do dzisiaj nie przedstawili państwo żadnej inicjatywy w tym zakresie.

Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Sebastian Kaleta. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mówimy o sprawie warszawiaków, którzy przez lata w zaciszu swoich kamienic musieli znosić wielkie krzywdy i cierpienia. Pukali oni do wielu drzwi, ale te drzwi nie były przed nimi otwierane.

Powstała komisja weryfikacyjna, która wyciągnęła na światło dzienne, zaprezentowała oblicze tej wielkiej afery, ale też oddała głos tym, którzy przez lata byli pomijani. Dzięki Wysokiej Izbie w poprzedniej kadencji parlamentu udało się przyjąć prawo, na podstawie którego te krzywdy z odzyskanych przez komisję środków powinny być naprawione w formie zadośćuczynień. Niestety politycy Platformy Obywatelskiej konsekwentnie odmawiają uznania tych krzywd.

Władze Warszawy ciągają swoich mieszkańców przed sądy. W imię czego?

Ustawa, nad którą procedujemy, zagwarantuje, że te krzywdy zostaną w końcu zadośćuczynione - to jest podstawowa rzecz, którą ta ustawa realizuje - i zabezpieczy inne osoby, które mieszkają w budynkach objętych roszczeniami i które boją się o dach nad głową, ponieważ były zapowiedzi, że w najbliższym czasie Warszawa przystąpi do zwrotów budynków w naturze.

Przez 30 lat problem reprywatyzacji nie został rozwiązany. Dlatego też ta propozycja, która znajduje się obecnie w Sejmie, jest kolejnym krokiem naprzód. Widzimy, że niestety nasze państwo nie uregulowało kwestii własnościowych. Podejmowanie kolejnych kroków, takich kroków jak ten, jest konieczne, by chronić poszczególne grupy osób, które mogą odczuwać negatywne skutki tego stanu prawnego. Tak jest z mieszkańcami Warszawy, dlatego ten projekt jest procedowany, dlatego ten projekt, mam nadzieję, zyska uznanie Wysokiej Izby. Natomiast oczywiście dyskusja nie jest zamknięta.

Natomiast dzisiaj rozwiązujemy problem tysięcy warszawiaków, którzy boją się o dach nad głową, setek ludzi, których Rafał Trzaskowski i Hanna Gronkiewicz-Waltz ciągają po warszawskich sądach, mając naprawdę na niskim poziomie priorytetów ich cierpienia. Dlatego też sprawę powinny załatwić parlament i rząd, a ci ludzie w końcu powinni móc o tych krzywdach zapomnieć i powiedzieć, że polskie państwo tym krzywdom zadośćuczyniło. Głos zabierze przedstawiciel wnioskodawców pan poseł Paweł Lisiecki.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Padło tutaj wiele różnego rodzaju deklaracji i oświadczeń, natomiast trzeba pewne rzeczy wyprostować. Ten projekt nie jest ustawą reprywatyzacyjną, żebyście mieli państwo tego świadomość. To nie jest ustawa, która ma na celu zwracać nieruchomości, natomiast ma na celu doprowadzić do tego, żeby pewne prawa osób mieszkających w tych budynkach były zapewnione.

Komuniści sami tych praw nie chcieli przestrzegać.

Trzeba jasno powiedzieć, że ta sytuacja jest zarówno problemem dla lokatorów, jak i prawowitych właścicieli. Z jednej strony dla lokatorów, jeżeli chodzi o wysoki czynsz, a z drugiej strony dla właścicieli, ponieważ często dochód z czynszu nie pozwala tak naprawdę naprawić strat czy nie pozwala doprowadzić takich budynków do stanu, który pozwalałby na ich użytkowanie.

Dzisiaj często dochodzi do sytuacji, w której roszczenia są zbywane przez prawowitych właścicieli na rzecz ludzi z mafii reprywatyzacyjnej, handlarzy roszczeń, którzy nabywają te roszczenia od tych właścicieli za ułamek wartości. I rzeczywiście, dobrze by było, aby również państwo wypłacało odszkodowania tymże prawowitym właścicielom. Natomiast sytuacja w tej chwili w mieście stołecznym Warszawa jest taka, że w tych zwróconych nieruchomościach znalazło się ok. 40 tys. ludzi, którzy podpisywali umowy najmu z miastem stołecznym Warszawa, z przedstawicielami władzy publicznej. Tymczasem zostali zwróceni razem z tymi lokalami, a ich umowy były rozwiązywane przez osoby, które przejmowały kamienice. Nie jest natomiast prawdą, że te nieruchomości w Warszawie otrzymywali wyłącznie złodzieje, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że w ok. 80% te decyzje dotyczące zwrotów były kierowane do prawowitych właścicieli. Natomiast szacujemy, że w ok. 20% były to budynki przejmowane przez mafię reprywatyzacyjną, handlarzy roszczeń, czyścicieli kamienic, którzy później dokonywali tego, czego dokonywali. Jedna to jest taka, aby te odszkodowania, które miało wypłacać miasto stołeczne Warszawa, przenieść do budżetu państwa. Za tym miałyby pójść pieniądze, które w mieście stołecznym Warszawa na ten cel były wpłacane, właściwie zabierane złodziejom i mafii reprywatyzacyjnej. Druga kwestia to jest doprowadzenie do sytuacji, w której zwrot nieruchomości nie byłby możliwy, dopóki miasto stołeczne Warszawa tak naprawdę nie zabierze ostatnich lokatorów z danej kamienicy. Chodzi de facto o doprowadzenie do tego, aby nie zwracać nieruchomości razem z lokatorami. Jako przedstawiciel wnioskodawców chciałbym jeszcze złożyć kilka poprawek do tego projektu, tak aby uporządkować pewne rzeczy. I tu, panie marszałku, na pana ręce te poprawki składam. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu sprawdzenia kworum. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek formalny o przerwanie posiedzenia i rozszerzenie porządku dziennego o punkt obejmujący przedstawienie przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli informacji na temat sytuacji w Najwyższej Izbie Kontroli w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa [[Oklaski]] złożonym przez prezesa NIK oraz wnioskiem o odwołanie wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wysoka Izbo! NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, kontroluje działalność NBP i państwowych osób prawnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli musi być jak żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami. Szanowni Państwo! Media donoszą o przekroczeniu uprawnień przez wiceprezesa NIK. Media donoszą o tym, że próbowano zastraszyć kontrolerów oraz wywierać nielegalny nacisk, jeśli chodzi o treść raportu kontroli doraźnej dotyczącej pomocy humanitarnej realizowanej przez rząd PiS. To sytuacja skandaliczna. Składam wniosek o przerwę i o umożliwienie prezesowi NIK. Nie ma tego w porządku obrad, panie pośle, tego posiedzenia Sejmu. W związku z tym. Odnoszę się, panie pośle. Mówię panu, że wniosek jest nieformalny, dlatego że nie dotyczy porządku dziennego posiedzenia Sejmu, który został uchwalony, panie pośle. Dziękuję bardzo. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw, - o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Sprawozdania to druki nr 478 i 472. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, - o Polskim Bonie Turystycznym, - o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to druki nr 476, 477 i 473. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 446 i 478) Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu powyższej uchwały wnosi, aby Sejm odrzucił obydwie poprawki. Dziękuję, pani poseł. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druki nr 443 i 472) Proszę pana posła Cezarego Grabarczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, które odbyło się w dniu wczorajszym, komisja rozpatrzyła dwie poprawki zgłoszone do ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie obydwu poprawek. Dziękuję. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy.

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 450 i 476) Proszę panią poseł Annę Milczanowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 r. wnosi: Dziękuję, pani poseł. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wniosek formalny, pan poseł Marek Sowa. Proszę. Mam nadzieję, panie pośle, że to będzie wniosek formalny dotyczący porządku dziennego tego posiedzenia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Dziękuję, panie pośle. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druki nr 449 i 477) Proszę panią poseł Teresę Wargocką o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zawarte w druku nr 477, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, druk nr 449. Marszałek Sejmu zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 7 lipca 2020 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu na posiedzeniu w dniu 14 lipca. Senat zgłosił do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym 65 poprawek, przy czym aż 36 poprawek miało charakter legislacyjno-redakcyjny. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu uchwały na posiedzeniu w dniu 14 lipca rekomenduje, aby Wysoka Izba 37 poprawek przyjęła i 27 poprawek odrzuciła. Wysoka Izbo! Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym złożona do laski marszałkowskiej przez pana prezydenta

dziecko niepełnosprawne to jest ogromne wsparcie.

Pani poseł, bardzo dziękuję. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw?

1 - za, przeciw - 436, 10 się wstrzymało. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Z poprawką tą łączą się poprawki 29., 50. i 56. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 27. i 28., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 30. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 65. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 445 i 473) Proszę panią poseł Annę Kwiecień o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury, druk nr 473, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, druk nr 445. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 19 czerwca 2020 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Senat zgłosił do art. 1 zawierającego zmiany do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Senat proponuje ujednolicenie terminologii. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nikt nie był za, 443 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Z poprawką tą łączy się poprawka 7. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 5. i 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Powołanie 3 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (druki nr 416 i 428)

Lista kandydatów na członków komisji została paniom i panom posłom doręczona w druku nr 416. Proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Milczanowską w celu przedstawienia opinii komisji.

Wysoka Izbo! Przedstawiam kandydatów na członków komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, którzy zostali zarekomendowani przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Są to: pani Karolina Bućko, pani Barbara Chrobak, pan Adam Czarnecki, pani Hanna Elżanowska, pan Marek Konopczyński, pani Teresa Barbara Matthews-Brzozowska, pan Andrzej Nowarski, pan Bartłomiej Tkacz, pan Tadeusz Bohdan Zaleski. Dziękuję, pani poseł. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur? Nikt się nie zgłasza. W takim razie proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem. Panie pośle, proszę nie pokrzykiwać, bo słyszę. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Aby możliwe było osiągnięcie celów stawianych przed komisją, potrzeba ludzi o odpowiednich kompetencjach wynikających z posiadanej wiedzy i życiowego doświadczenia, ludzi wrażliwych, odważnych i zaangażowanych. Od składu tej komisji zależeć będzie jej rzeczywisty bądź fikcyjny, pozorny charakter. Od konkretnych ludzi podejmujących się tego ogromnie trudnego zadania i ogromnej odpowiedzialności zależeć będzie zdolność komisji do przełamania bezradności i bezsilności państwa w zwalczaniu pedofilii. Takim członkiem komisji będzie prof. Marek Konopczyński - profesor zwyczajny, ekspert od patologii społecznych, nauczyciel akademicki, autor licznych analiz i opracowań z tego obszaru spraw społecznych, zaangażowany w wiele działań i inicjatyw społecznych, absolwent Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie prof. Marek Konopczyński kieruje katedrą pedagogiki specjalnej na uniwersytecie białostockim. Wcześniej był m.in. rektorem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Współpracował także z Akademią Ignatianum ojców jezuitów w Krakowie. Jest redaktorem naczelnym periodyku „Resocjalizacja Polska” oraz zastępcą przewodniczącego rady naukowej miesięcznika „Policja 997” Jest założycielem fundacji Pedagogium, która pracuje z ofiarami i sprawcami przestępstw. Prof. Konopczyński uważa, iż pedofilia jest jak rak. Trzeba ją właściwie diagnozować, aby skutecznie leczyć. Jeśli nie będzie prawidłowej diagnozy i właściwego leczenia, skutki mogą być katastrofalne, o czym świadczą losy ofiar. Prof. Marek Konopczyński podkreśla, iż do skutecznej walki z tą ciężką chorobą społeczną potrzeba szerokiej, stałej i intensywnej współpracy, trzeba szerokiej i mocnej koalicji w obronie krzywdzonych i zagrożonych skrzywdzeniem dzieci. Potrzeba zwłaszcza starannie przemyślanej i szeroko akceptowanej oraz konsekwentnie realizowanej profilaktyki i edukacji, kierowanych przede wszystkim do dzieci i ich rodziców lub opiekunów. Dlatego też z głębokim przekonaniem zgłaszamy prof. Marka Konopczyńskiego na członka komisji do spraw zwalczania nadużyć seksualnych wobec dzieci. O ocenie kandydatury prof. Konopczyńskiego dobitnie świadczy wynik głosowania na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 19 czerwca 2020 r., gdzie prof. Marek Konopczyński uzyskał najwięcej, bo 21, głosów za, a nikt nie głosował przeciw. Proszę.

Szczęść Boże! Rzadka to okazja dla posłów Konfederacji nie tylko popierać kandydatury przez innych wysunięte, ale także mieć swój skromny udział w wysuwaniu kandydatur do tego gremium, które oczywiście jest jakąś formą działania zastępczego, leczenia objawowego. Jest to wbrew pozorom, które z lewa i z prawa państwo staracie się stwarzać, budowanie wyższego piętra hipokryzji w naszym życiu publicznym, bo chcecie państwo - i słusznie - tropić, ścigać i, mam nadzieję, przykładnie karać. Przecież to jest tylko szczególnie ohydny przypadek, ale na szerszym tle, to szersze zjawisko. Państwo jesteście z lewa i z prawa podporządkowani poprawności politycznej. W waszym języku, którego używacie wobec rewolucyjnej inwazji dewiacji i promocji dewiacji w naszym życiu publicznym, i temu nie jesteście się w stanie sprzeciwić.

Mam nadzieję, że procedowanie w tej komisji, w której z radością zobaczymy przynajmniej jednego sprawiedliwego, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, będzie prowadzić do rzeczywistej naprawy stanu Rzeczypospolitej, tak że do aresztów pakować się będzie dewiantów i promotorów dewiacji, nie zaś tych, którzy próbują się przeciwstawić tej rewolucyjnej inwazji. Nie ważcie się używać tej komisji, do której, owszem, delegujemy naszego przedstawiciela, ale nie będziemy tam mieli większości, nie ważcie się używać tego narzędzia do walki z typowanymi przez was arbitralnie, selektywnie winowajcami.

Panie pośle, dziękuję bardzo.

Nic panu nie radzę, panie pośle, dziękuję panu. Pan poseł Jarosław Sachajko, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Proszę. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 oraz Koła Poselskiego Konfederacja mam zaszczyt przedstawić kandydaturę ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego jako kandydata na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaświadczył swoim życiem, iż dla niego ważne są dwie rzeczy: dobro dzieci oraz sprawa oczyszczenia i transparentności Kościoła. Jest on najbardziej wyrazistym duchownym, który otwarcie mówi i pisze o zmowie milczenia na temat pedofilii w Kościele. Ze wszystkich kandydatów najlepiej zna środowisko kościelne i otwarcie mówi, gdzie jest patologia i jak można jej zaradzić. Jeszcze w czasie studiów jako uczestnik międzynarodowego ruchu Wiara i Światło zakładał w Krakowie i Chrzanowie wspólnoty osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców i opiekunów. W 1987 r. był współzałożycielem ogólnopolskiej Fundacji im. Brata Alberta i schroniska dla niepełnosprawnych w Radwanowicach. Fundacja ta prowadzi na terenie całego kraju 35 placówek dla 1200 podopiecznych.

Należy również podkreślić, iż wobec ks. Isakowicza-Zaleskiego jako opozycjonisty w okresie PRL-u były prowadzone działania operacyjne przez ówczesne tajne służby. Nie były to jedynie działania inwigilacyjne, ale były podejmowane wobec niego prowokacje.

Spośród licznych książek napisanych przez księdza należy wymienić książkę pt. „Chodzi mi tylko o prawdę”, poruszającą tematy niedokończonej lustracji w polskim Kościele, homoseksualizmu wśród części duchowieństwa, zaangażowania politycznego duszpasterzy czy ludobójstwa na Kresach Wschodnich. W czerwcu obecnego roku ukazała się kolejna książka, pod dużo mówiącym tytułem „Kościół ma być przezroczysty” Wysoka Izbo! Uzyskanie większości sejmowej dla tej kandydatury będzie testem, na ile poważnie parlamentarzyści, politycy podchodzą do tematu pedofilii i czy nie powstanie kolejna komisja strachu, która będzie miała za zadanie polityczne wykorzystanie krzywdy dzieci.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 to bardzo ważne gremium, którego ideą działania będzie troska o dobro dziecka, a także wyjaśnianie przypadków takich haniebnych i nikczemnych działań. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje dwóch kandydatów na członków państwowej komisji. Tymi kandydatami są pani dr Hanna Elżanowska oraz pan mecenas Andrzej Nowarski. Współpracuje z uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Jest absolwentką 5-letniego kursu psychoterapii i terapii rodzin organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką psychologiczną, poradnictwem, psychoterapią indywidualną i terapią rodzin. Pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci. Pan mecenas Andrzej Nowarski jest radcą prawnym z 15-letnim doświadczeniem zawodowym.

Został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Mecenas Andrzej Nowarski zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach w Krakowie i Warszawie. Zajmował się szerokim spektrum spraw z wielu dziedzin prawa. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Od 2014 r. świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. Od 2018 r. współpracuje z ministerstwem kultury. Zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie zawodowe pani dr Hanny Elżanowskiej oraz pana mecenasa Nowarskiego dają pewność, że są oni dobrymi kandydatami na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Dziękuję, pani poseł.

Wysoka Izbo! Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma zajmować się wszystkimi przestępstwami, nie tylko tymi popełnianymi przez Kościół, choć to właśnie Kościół systemowo chronił sprawców, nie rozliczył się z tego i nie chce nawet wypłacać ofiarom odszkodowań. Komisja, potocznie nazywana komisją do spraw pedofilii, dostała ogromny budżet, jest to 12 mln zł. Nie będzie przyznawać odszkodowań, będzie za to wpisywać sprawcę do specjalnego rejestru, co budzi wątpliwości, bo w rejestrze można się znaleźć bez wyroku sądowego, a o winie orzekną członkowie komisji. W komisji ma zasiadać siedem osób. Pierwotnie mieli być to tylko lekarze, psychologowie, prawnicy, ale po zmianie do ustawy COVID-owej wystarczy teraz np. odznaczenie otrzymane od prezydenta. Dziesięć osób - tyle liczyła lista przedstawiona nam w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wśród tych kandydatur szczególnie wyróżnia się kandydatka zgłoszona przez klub parlamentarny Lewicy. Jako jedyna. Pani mecenas Karolina Bućko to nie tylko prawniczka, adwokatka aktywna zawodowo od 2005 r., prowadząca własną kancelarię, ale również osoba z szerokim wykształceniem prawniczym.

Mamy nadzieję, że to nie jest kolejny sposób na uwłaszczenie partii rządzącej i że ten skład będzie w miarę obiektywny, merytoryczny i rzeczowy. Zamykam dyskusję. Powołanie członków komisji przez Sejm odbywa się zgodnie z następującymi zasadami. Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdego z trzech powołań. Jeżeli w pierwszym głosowaniu kandydat nie uzyskał większości 3/5 głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, a Sejm powołuje członka komisji zwykłą większością głosów. Pod głosowanie poddam kandydatury w kolejności alfabetycznej. Pozostałe kandydatury będą poddane pod głosowanie w procedurze powołania kolejnego członka komisji. Przypominam, że zgłoszone zostały kandydatury: - pani Karoliny Bućko, zgłoszonej przez grupę posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia), - pani Barbary Chrobak, zgłoszonej przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, - pana Adama Czarneckiego, zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie, - pani Hanny Elżanowskiej, zgłoszonej przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, - pana Marka Konopoczyńskiego, zgłoszonego przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, - pani Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej, zgłoszonej przez Naczelną Izbę Lekarską, - pana Andrzeja Nowarskiego, zgłoszonego przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, - pana Bartłomieja Tkacza, zgłoszonego przez Krajową Radę Radców Prawnych, - pana Tadeusza Bohdana Zaleskiego, zgłoszonego przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 oraz Koła Poselskiego Konfederacja. Ponadto informuję, że pan Radosław Krajewski, zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wycofał swoją zgodę na kandydowanie na członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad powołaniem pierwszego członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani Karoliny Bućko. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Karoliny Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć

Większość 3/5 wynosi 270 głosów. Za było 178, przeciw - 244, wstrzymało się 28. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Karoliny Bućko na członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani Barbary Chrobak. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Barbary Chrobak na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Barbary Chrobak na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Adama Czarneckiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Adama Czarneckiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Hanny Elżanowskiej na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Hanny Elżanowskiej na członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pana Marka Konopczyńskiego. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Marka Konopczyńskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Marka Konopczyńskiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Andrzeja Nowarskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Andrzeja Nowarskiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Bartłomieja Tkacza na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Bartłomieja Tkacza na członka komisji. Przepraszam bardzo. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem ks. Tadeusza Bohdana Zaleskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał ks. Tadeusza Bohdana Zaleskiego na członka komisji. Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów przez żadnego z kandydatów przystąpimy do ponownego głosowania w tej sprawie. Przypominam, że w tym przypadku Sejm powołuje członka komisji zwykłą większością głosów. Pod głosowanie poddam ponownie kandydatury w kolejności alfabetycznej. Uzyskanie zwykłej większości głosów przez jednego z kandydatów oznaczało będzie zakończenie procedury powołania pierwszego członka komisji. Pozostałe kandydatury będą poddane pod głosowanie w procedurze powołania kolejnego członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani Karoliny Bućko. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Karoliny Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosowało 449 posłów. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Karoliny Bućko na członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani Barbary Chrobak. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Barbary Chrobak na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Przepraszam, źle zostały wyświetlone wyniki. Sejm większością głosów powołał panią Barbarę Chrobak na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, a tym samym powołał pierwszego członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad powołaniem drugiego członka komisji. Pod głosowanie poddam kandydatury w kolejności alfabetycznej. Pozostałe kandydatury będą poddane pod głosowanie w procedurze powołania kolejnego członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani Karoliny Bućko. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Karoliny Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę państwa, to jest procedura wynikająca z ustawy. Państwo nie słuchaliście, co czytałam na początku. Musimy tak głosować, musimy.

To jest procedura ustawowa.

I proszę się nie oburzać, bo to jest procedura ustawowa. Głosujemy. Jeszcze raz pytam. Kto jest za? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Karoliny Bućko na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Adama Czarneckiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Adama Czarneckiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Hanny Elżanowskiej na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Hanny Elżanowskiej na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Marka Konopczyńskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Za - 180, przeciw - 232, 31 wstrzymało się. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Marka Konopczyńskiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad kandydaturą pana Andrzeja Nowarskiego. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Andrzeja Nowarskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Andrzeja Nowarskiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Bartłomieja Tkacza na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Bartłomieja Tkacza na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem ks. Tadeusza Bohdana Zaleskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

to jest większość 3/5. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał ks. Tadeusza Bohdana Zaleskiego na członka komisji. Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów przez wszystkich kandydatów przystąpimy do ponownego głosowania w tej sprawie. Przypominam, że w tym przypadku Sejm powołuje członka komisji zwykłą większością głosów. Uzyskanie zwykłej większości głosów przez jednego z kandydatów oznaczało będzie zakończenie procedury powołania drugiego członka komisji. Pozostałe kandydatury będą poddane pod głosowanie w procedurze powołania kolejnego członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad powołaniem drugiego członka komisji zwykłą większością głosów. Głosujemy nad kandydaturą pani Karoliny Bućko. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Karoliny Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Karoliny Bućko na członka komisji. Głosujemy nad kandydaturą pana Adama Czarneckiego. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Adama Czarneckiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Adama Czarneckiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Hanny Elżanowskiej na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm większością głosów powołał panią Hannę Elżanowską na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, a tym samym powołał drugiego członka komisji.

Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Karoliny Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Karoliny Bućko na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Adama Czarneckiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Adama Czarneckiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Marka Konopczyńskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Marka Konopczyńskiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Andrzeja Nowarskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Andrzeja Nowarskiego na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Bartłomieja Tkacza na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pana Bartłomieja Tkacza na członka komisji.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał ks. Tadeusza Bohdana Zaleskiego na członka komisji. Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów przez wszystkich kandydatów przystąpimy do ponownego głosowania w tej sprawie. Przypominam, że w tym przypadku Sejm powołuje członka komisji zwykłą większością głosów. Uzyskanie zwykłej większości głosów przez jednego z kandydatów oznaczało będzie zakończenie procedury powołania trzeciego członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad powołaniem trzeciego członka komisji zwykłą większością głosów. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani Karoliny Bućko. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Karoliny Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Karoliny Bućko na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Adama Czarneckiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał pani Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka komisji. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Andrzeja Nowarskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm większością głosów powołał pana Andrzeja Nowarskiego na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, a tym samym powołał trzeciego członka komisji. Proszę państwa, na tym zakończyliśmy procedurę wyboru trzech członków komisji. Ogłaszam 10 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego (druki nr 453 i 474) Proszę przedstawiciela wnioskodawców pana posła Tomasza Szymańskiego o przedstawienie uzasadnienia wniosku. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czas wyznaczony na uzasadnienie wniosku jest zdecydowanie za krótki. Przez 5 minut nie da się przedstawić Wysokiej Izbie oraz milionom Polek i Polaków całej listy zaniechań i nadużyć, których dopuścił się minister Mariusz Kamiński. Ba, przez 5 minut nie uda się ugotować jajek na twardo. A tyle właśnie czasu dajecie państwo opozycji na uzasadnienie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec konstytucyjnego ministra. Składając wniosek o wotum nieufności, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec nienależytego wypełniania obowiązków służbowych oraz nadużywania władzy, a tym samym nieprzestrzegania obowiązującego prawa, w tym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego chcemy odwołania pana ministra Mariusza Kamińskiego? Powodów jest wiele, czasu mało, wymienię więc siedem grzechów głównych pana ministra Mariusza Kamińskiego. Grzech pierwszy - zaangażowanie służb w bezwzględne tłumienie protestów obywateli. Zgodnie z konstytucją każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Tymczasem służby podległe ministrowi Kamińskiemu zostały zaangażowane w bezwzględne tłumienie protestów obywateli. Doskonale pamiętamy protest przedsiębiorców, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec nieudolnej polityki rządu Mateusza Morawieckiego, a w szczególności w zakresie braku pomocy państwa w związku z panującą epidemią koronawirusa. Doskonale wiemy, że wielu przedsiębiorcom do dziś nie zapewniono oczekiwanego przez nich wsparcia. Ludzie ci spontanicznie wyszli na ulicę, by ratować miejsca pracy, by nadal móc uczciwie pracować i zarabiać pieniądze. Jak ich potraktowano? Zaangażowano do tego podległą ministrowi Kamińskiemu Policję. Policję, w której szeregach są porządni obywatele, ludzie, którzy zakładają mundur nie po to, by być wykorzystywanymi do tłumienia pokojowych protestów obywateli, lecz po to, by bronić najsłabszych i dbać o ich bezpieczeństwo. Tymczasem w ostatnich latach wykorzystuje się ich do zupełnie innych celów. I tu jest drugi grzech ministra Kamińskiego - wykorzystywanie służb do zadań, do których nie zostały powołane. Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi. Tymczasem ze względu na ogromne zaangażowanie polityczne Mariusza Kamińskiego oraz budowanie przez niego swojej pozycji w obozie władzy służby mu podległe wykorzystywane są do zadań, do których nie zostały powołane. Jednym z przykładów najlepiej obrazujących ten proceder jest wykorzystanie podległej ministrowi Kamińskiemu Policji do patrolowania okolic domu jego partyjnego szefa, pana posła Jarosława Kaczyńskiego.

polska Policja to nie partyjny folwark. Polska Policja została utworzona po to, aby służyć społeczeństwu, a nie waszej partii. Grzech trzeci - działanie bez podstawy prawnej. Zgodnie z konstytucją organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tymczasem Mariusz Kamiński podjął się przygotowań do przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pomijając w tym procesie najwyższy i najważniejszy organ państwowy, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza. Doskonale pamiętamy, z jakim uporem PiS dążyło do przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 10 maja. Pamiętamy o pakietach wyborczych wydrukowanych za 70 mln zł, o tym, że taki pakiet trafił do jednego z kandydatów. Panie ministrze, profesjonalizm na miarę San Escobar. Grzech czwarty - totalny brak profesjonalizmu. Good afternoon, mister president - brzmi to śmiesznie, banalnie, ale niestety jest na pozór bardzo niebezpieczne. Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów pan Mariusz Kamiński sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością służb specjalnych i koordynuje ich działania. Tymczasem służby podległe panu ministrowi nie potrafiły zapobiec rozmowie pana prezydenta z rosyjskim youtuberem, który przedstawił się jako sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Służby, które powinny dbać o bezpieczeństwo Polski, dopuściły do tego, że prezydent przez ponad 11 minut rozmawiał z jakimś rosyjskim youtuberem, który następnie wrzucił nagraną rozmowę do sieci. Czy dociera do pana, panie ministrze, co się tak naprawdę stało? Tłumaczenia, że nagrany został również premier Boris Johnson, są słabe. W Wielkiej Brytanii państwo zadziałało. Pragnę przypomnieć, że połączenie to zostało przerwane. W Polsce prezydent rozmawiał ponad 11 minut łamaną angielszczyzną. Ośmieszyliście państwo urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ośmieszyliście Polskę. Pokazaliście, że każdy ot tak może zadzwonić do głowy państwa i urządzić sobie pogawędkę. Już dziś ludzie drwią, że szybciej można dodzwonić się do prezydenta Polski niż na infolinię ZUS albo urzędu skarbowego. Grzech piąty - inwigilacja. Zgodnie z konstytucją władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie. Tymczasem minister Kamiński pozostaje odpowiedzialny za wysoce prawdopodobne funkcjonowanie w Polsce systemu Pegasus, zakupionego za 35 mln zł (Dzwonek), służącego do nieograniczonego podsłuchiwania obywateli. Dziękuję. Szanowni Państwo! Oczywiście ten czas, o którym na początku wspomniałem, jest niewspółmiernie krótki do zarzutów, które możemy. Bardzo proszę, pani marszałek, o umożliwienie mi spuentowania zasadnego wniosku. Złożony przeze mnie, przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego stanowi próbę zahamowania działań rządu zmierzających do pogłębienia kryzysu demokratycznego w Polsce. Jest także próbą obrony praw człowieka, które w arogancki sposób łamane są przez służby podległe ministrowi Kamińskiemu. oraz działaniem mającym na celu zaprzestanie dalszego wykorzystania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych do celów, do których nie zostały powołane. Szanowna Pani Marszałek! Proszę pana posła Jerzego Polaczka o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, która wczoraj rozpatrywała ten wniosek, w sposób jednoznaczny opowiedziała się za odrzuceniem propozycji ze strony wnioskodawców i rekomenduje odrzucenie propozycji, aby minister spraw wewnętrznych miał być w tej materii oceniony negatywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Przypominam, że zgodnie z art. 116 ust. 1a regulaminu Sejmu po wyczerpaniu listy mówców głos może zabrać tylko prezes Rady Ministrów oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Zdzisław Sipiera - ze stanowiskiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Reszta - omawiana w lutym, kiedy był pierwszy wniosek o odwołanie ministra, ale jako koordynatora służb specjalnych - w tym wniosku tak naprawdę omawiana nie jest, dlatego że nie dotyczy tego ministra, którego państwo wywołaliście. To jest pierwsza uwaga formalna, ale moim zdaniem bardzo istotna, bo sygnuje to, że ten wniosek nie jest wnioskiem literalnie formalnoprawnym, tylko jest po prostu politycznym wnioskiem, który ma zrobić pewnego rodzaju entourage, który mówi o tym, że jeżeli jest wniosek o odwołanie ministra, to kompetencje bierze się z kogoś innego. Oczywiście to jest ta sama osoba, ale jednak inne kompetencje. W tym wniosku są literalnie dwa zarzuty wobec ministra. Pierwszy wniosek zakłada nieadekwatność zachowań, działań Policji, a drugi wniosek, który jest w tym zawarty, to sformułowanie, że premier polskiego rządu wydał polecenie panu ministrowi. To naprawdę są dwie bardzo ciekawe konstrukcje, które mogą służyć do tego, żeby ten wniosek miał powagę formalnoprawną. A jakie są pozostałe zarzuty, szanowni państwo?

No naprawdę sama merytoryka, głęboka merytoryka zawarta jest w tym wniosku. Żadnych konkretów, tylko ogólny entourage, który ma powiedzieć: coś się dzieje. We wniosku, proszę państwa, są też daleko idące insynuacje, które mówią o wykorzystywaniu funkcji czy braku działań ministra w celu zabezpieczenia interesów polskich. Powiem tak, proszę państwa, w imieniu klubu: dziwimy się, bo tutaj mamy dwoistość postępowania. Z jednej strony wnioskodawcy mówią: minister powinien działać tak, że nic się w państwie nie zdarzy bez jego zgody, a z drugiej strony padają w tym wnioski sformułowane w ten sposób, że minister tak naprawdę używa wszystkiego, co ma, do tego, żeby stłumić wolność w Polsce. Albo jedno, albo drugie. Albo jest tak, że faktycznie pan minister jest tak wielki, że wszystko się dzieje, czyli nic się nie dzieje bez jego zgody, albo faktycznie jest państwo prawa, które działa formalnie i normalnie i jest następstwo tych działań. A państwo zarzucacie we wniosku, że coś się dzieje przed, a nie po - to jest niekonsekwencja.

Ale jeżeli mówimy o poważnym państwie, to powinny być wobec tak poważnego ministra poważne zarzuty, a ich nie ma w ogóle. Minister Mariusz Kamiński w opinii naszego klubu bardzo dobrze wypełnia swoją funkcję, jest bardzo dobrym ministrem, świetnie koordynuje prace komisji i innych służb, które są mu podległe jako ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Absolutnie zasługuje na pełne wsparcie, a nawet więcej.

To takie twórcze, bardzo artystyczne podejście. Ale podstawowa sprawa, proszę państwa, która dotyka powagi tego wniosku, jest chyba zawarta w cytacie i pozwolą państwo, że go odczytam na końcu. Wnioskodawcy: „Ponadto dymisja ministra Mariusza Kamińskiego w sposób znaczący mogłaby przysłużyć się ograniczeniu możliwości korupcji w administracji państwowej”

No ale można powiedzieć tak: jaki jest wniosek, tak też działa opozycja, taka właśnie jest siła tej opozycji. Ta wielka armata, którą państwo wytoczyliście, jest właśnie dokładnie ujęta w tym wniosku, miałkim, żadnym.

Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak, będziemy głosować za odwołaniem pana ministra, tak naprawdę z trzech powodów. Po pierwsze, pan minister użył Policji państwowej na gruncie ustaw COVID-owskich sprzecznie z prawem i z konstytucją. Otóż zapisy ustawy o Policji nierozszerzone o działania w zakresie prawa administracyjnego nie pozwalały panu wypuszczać policjantów i nakazywać im łamanie praw i wolności obywatelskich [[Oklaski]] inaczej niż poprzez ustawy o stanie wyjątkowym. Otóż prawda jest taka, że to, że policja jest używana do zaganiania ludzi na rowerach, do ścigania ludzi, którzy wychodzą na spacer z niepełnosprawnymi, to jest pana odpowiedzialność, nie policjantów, pana. Pan złamał ustawę, pan nie ma prawa używać policji na gruncie ustaw, które są wadliwe, jeśli chodzi o prawa i obowiązki obywatelskie. I ten zarzut jest zarzutem bardzo poważnym.

Czy 160 mln wróciło do państwa polskiego, czy nie? Czy nadal można, będąc żoną instruktora narciarskiego pana kolegi w rządzie, jednego dnia założyć firmę, a drugiego dnia dostać 5 mln od państwa, od podatników, od nas na rachunek tej firmy? Nagle się okazuje, że nic w tej sprawie nie można zrobić, że służby i Policja są bezczynne. Pan się broni w ten sposób, że to są służby, a pan tu odpowiada jako minister. Chciałbym powiedzieć, panie ministrze, jedną rzecz. Ma pan pod sobą potężny pion kryminalny. Otóż gdyby młodszy aspirant z tego pionu dostał materiały tej sprawy, to za 2 dni byłyby aresztowania, byłyby zajęte materiały, wszystko by się potoczyło idealnie, tylko że on ich nie dostał. Jak to kontrastuje z tą niezwykłą skutecznością podległych panu funkcjonariuszy, kiedy np. trzeba ścigać marszałka Senatu, ponieważ jest waszym przeciwnikiem politycznym. Pan jest bezradny wobec tego bagna, które się odbywa w pańskim rządzie, a równocześnie jest pan niezwykle sprawny i okrutny wobec przeciwników politycznych. I to jest prawda o panu jako szeryfie walczącym z korupcją. Ostatnia sprawa, moim zdaniem, niezwykle obciążająca, panie ministrze. Otóż pan w ostatnich dniach, w dniach kampanii wyborczej, handlował bezpieczeństwem Polski, [[Oklaski]] handlował pan w ordynarnych politycznych dealach. Czym innym jest komunikat RCB wysłany SMS-em wbrew wyraźnym zapisom ustawy - art. 21a pkt 1 mówi, że takie komunikaty się wysyła wyłącznie w sytuacji zagrożenia, a pan wziął udział w kampanii wyborczej Andrzeja Duda, pan grał na frekwencję, która była korzystna dla tego kandydata. Panie ministrze, czy tak pan spłaca długi wobec prezydenta za ułaskawienie, które umożliwiło panu bycie ministrem? Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Już zbliża się koniec. Pan się bardzo chętnie chowa za policjantów i mówi, że atak na pana jest atakiem na ciężko pracujących policjantów.

To nie ma nic wspólnego z obrażaniem Policji. Niech pan się nie chowa tchórzliwie za mundurami policjantów, bo pan nie jest jednym z nich. Pan jest ich politycznym nadzorcą i ponosi pan pełną odpowiedzialność za to, co się w niej dzieje. Jest jedno usprawiedliwienie, które można by od pana ministra usłyszeć. Otóż to usprawiedliwienie jest takie: tak jak Policja jest ślepym mieczem w pana rękach, tak pan jest ślepym mieczem w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Pan tworzy państwo policyjne, państwo stanu wyjątkowego bez ustaw o stanie wyjątkowym. To jest państwo, które Jarosław Kaczyński zaprojektował dla nas wszystkich, a pan jest jego wykonawcą.

Pan poseł Andrzej Rozenek w imieniu klubu parlamentarnego Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny panie ministrze, nie da się rozdzielić funkcji ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Nie da się, bo obydwie funkcje sprawuje jedna osoba, konkretnie pan. Stąd musi pan być w tej chwili, jak ta znana żaba z pewnej anegdoty, i piękny, i mądry. Nie da rady inaczej, panie ministrze. Zacznijmy od tej drugiej funkcji. Komicy z Rosji nagrali i ośmieszyli prezydenta Polski. Gdzie były służby? Chciałem zapytać, jak sprawdzono kontrahenta przy transakcji na respiratory, która kosztowała budżet państwa prawie 200 mln? Czy wiedzieliście o tym, że jest to handlarz bronią o szemranej przeszłości? Czy w ogóle jakakolwiek podległa panu służba rzeczywiście dała ministrowi zdrowia zielone światło na tę transakcję? Powiem szczerze, nie chce mi się w to wierzyć. Niech pan ma odwagę i powie, jak było naprawdę, że nikt służb o to nie pytał, bo gdyby było inaczej, to jest to ogromna kompromitacja polskich służb. Maseczki bez certyfikatów kupione od instruktora narciarstwa, przyłbice kupione od handlarza oscypków. Szanowny panie ministrze, w sytuacji gdy z powodu epidemii pozwala się na zakupy poza rygorami ustawy - Prawo zamówień publicznych, rola służ specjalnych jest szczególnie istotna. Czy może pan powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że zrobiono w tej sprawie wszystko, co należało zrobić? Czy podległe panu służby wykazały się profesjonalizmem i czujnością, czy też może przymknęły oko na deale, które robiono w Ministerstwie Zdrowia? Chwalę tu pana ministra. Zapowiedziane dodatki dla policjantów, żeby pozostawali w służbie pomimo nabycia praw emerytalnych, również chwalebne, popieram, bo doświadczeni policjanci są bardzo potrzebni w służbie, o tym wszyscy wiemy. Czy nie można było o tym pomyśleć znacznie wcześniej? Czy potrzebne były ślepe czystki pod hasłem: święto Policji bez milicji? Pozbyliście się wtedy znakomitych fachowców. Wielu z nich mogłoby nadal służyć społeczeństwu i przekazywać swoje doświadczenie młodszym kolegom.

Pilnujecie skrzynki pocztowej na płocie prezesa, zamiast pilnować bezpieczeństwa zwykłych obywateli. Niestety, rośnie fala przestępstw. Coraz więcej jest włamań do domów, coraz częściej kradzione są samochody. A Policja? Policja musi walczyć z obywatelami, którzy protestują, zamiast walczyć z przestępcami. Nakaz zachowania dystansu społecznego był pretekstem do brutalnych interwencji Policji. Gdzie jest równość wobec prawa? W czasie protestu pod siedzibą Trójki policjanci wręczali mandaty za trzymanie kartek z hasłami: 50 zł za hasło „Murem za Niedźwiedziem”, ale już stówa za hasło „Wolne media” Panie ministrze, co to jest za taryfikator? Doszło do tego, że policjanci w dniach protestów antyrządowych szli na urlopy, bo nie chcieli konfrontacji z obywatelami, nie chcieli brać w tym udziału. Policjanci wykazali się większym rozsądkiem niż rządzący nimi politycy, bo Policja jest państwowa, a nie pana Kamińskiego ani nawet pana Kaczyńskiego. I na koniec sprawa dla mnie szczególnie bolesna. Do pana należy przywilej skorzystania z art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Nie słyszałem jednak, żeby skorzystał pan z tego artykułu i przywrócił komukolwiek ukradzioną emeryturę. Nie skorzystał pan z tego prawa w przypadku tak zasłużonych osób, jak Grażyna Biskupska, Piotr Wróbel czy gen. Gromosław Czempiński. Nie skorzystał pan z tego prawa nawet wobec inwalidów, wdów i sierot po funkcjonariuszach. Za to podległy panu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA kieruje do kolejnych osób informacje o odebraniu znaczącej części emerytury. Tym razem haniebna ustawa represyjna jest wykorzystywana przeciwko emerytom z pionu paszportowego i pionu łączności MSW. Wiem, że macie zamiar obniżyć emerytury następnym grupom społecznym. To zemsta polityczna oparta na odpowiedzialności zbiorowej, która nie jest znana w demokratycznych systemach, [[Dzwonek]] za to bywa często stosowana w dyktaturach. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata, w której mam honor reprezentować klub poselski Koalicja Polska - PSL - Kukiz15, dotyczy wyrażenia wotum nieufności wobec ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, a tym samym stanowi doskonałą okazję do dyskusji, oceny przygotowania oraz reakcji państwa polskiego na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Wiemy dobrze, że rząd polski został zaskoczony pandemią. Rząd polski nie był przygotowany na wybuch pandemii, natomiast w samej sferze zarządzania kryzysowego działania były pełne chaosu, pozbawione szerszego planu. Przepraszam, jeden plan był - wygrać wybory prezydenckie. Wysoka Izbo! W ustawach marcowych, słynnych ustawach COVID-owskich, rząd wprowadził zmiany w systemie zarządzania kryzysowego, tworząc de facto alternatywny system zarządzania kryzysowego, podważając aktualny stan prawny, który dobrze funkcjonował. System ten, obowiązujący od marca, zmodyfikował czasowo bądź też zdublował istniejący system, wprowadzając nowy, który działa wyłącznie po linii administracji rządowej, czyli prezesa Rady Ministrów, właściwego ministra lub głównego inspektora sanitarnego i wojewody. Patrząc na działania rządu, dostrzec można, że w KPRM-ie zorganizowano quasi-nieformalne centrum antykryzysowe premiera złożone z Centrum Analiz Strategicznych - CAS i Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pojawiło się nagle tylko raz. RCB objawiło się w momencie wyborów, ogłaszając sławetny alert. Wysoka Izbo! Teraz skupię się na straży pożarnej. Chciałbym zacytować pewien list związkowców do komendanta głównego. Związki zawodowe działające w PSP, mając na uwadze bezpieczeństwo strażaków, wystąpiły 11 marca do komendanta głównego z wnioskiem, cytuję: o opracowanie lub przedstawienie procedur obowiązujących strażaków podczas prowadzenia działań związanych z wirusem. Wskazano również, żeby do czasu ustalenia i opracowania tych wszystkich uregulowań powyższych kwestii, jak również do czasu zapewnienia niezbędnych indywidualnych środków ochronnych oraz zapoznania funkcjonariuszy z procedurami postepowania z wirusem SARS-CoV-2, ograniczono się do niezbędnych działań.

Co więcej, podobnie wygląda sytuacja w kwestii ochrony ludności, obrony cywilnej kraju. Jej szef, komendant główny PSP, jak można się dowiedzieć z publicznych i dostępnych danych, nawet nie podjął próby koordynacji działań szefów obrony cywilnej województw i wojewodów. Dlaczego nastąpiło zdublowanie tego systemu i budowanie systemu centralistycznego? Zdaję sobie sprawę, że elity Prawa i Sprawiedliwości robią wszystko na rozkaz, że chcą stworzyć system ratowniczy, który będzie działał według rozkazu, ale jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może za tym iść coś kolejnego. Może doprowadzić to do zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy, która się wykluła w ciężkiej pracy, za sprawą której ratowano życie ludzkie. I ta ustawa może zostać zakwestionowana. A może z tego tylko powodu, że to jest system zdecentralizowany, zdecentralizowany system, który funkcjonuje najlepiej, gdy nie ma polityków z Warszawy w terenie. Kolejna sprawa, krótko już. Teraz jest to temat najistotniejszy, najbardziej trudny, o którym musimy powiedzieć. To jest to, że każdy zakup, który organizował rząd - maseczka, przyłbica, testy, tarcza, wydano prawie miliard złotych - te wszystkie zakupy były zakupami nieskutecznymi, a przecież minister dysponuje Policją, innymi służbami, i powinna być kontrola.

Służby powinny działać jeszcze o wiele bardziej skutecznie. tego typu transakcji, po to żeby chronić urzędników państwowych. Jak sami widzimy, afera goni aferę. Widzimy brak przygotowania do zagrożenia, którego można było się spodziewać. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Krzysztof Tuduj. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności względem ministra Kamińskiego jest niemerytoryczny, słaby i chaotyczny.

Przechodziłem koło tej budki, kiedy ona płonęła. Z tymi złymi również dla polskiej Policji czasami nie chcemy mieć nic wspólnego. Nie jesteśmy jako Konfederacja opozycją totalną i widzimy, że obecnie w resorcie dzieją się również pozytywne i długo oczekiwane przez środowiska mundurowe rzeczy. Mam nadzieję, że uda się w najbliższym czasie skutecznie rozwiązać szalenie palący problem braków kadrowych, szczególnie w Policji, bo niełatwa służba dla państwa polskiego powinna być zawsze należycie dowartościowana, a funkcjonariusze powinni mieć zapewniony możliwy komfort jej pełnienia. Do pracy pana ministra Kamińskiego Konfederacja ma jednak własne zastrzeżenia, choćby takie jak brak prac nad łatwiejszym dostępem do broni palnej dla odpowiedzialnych Polaków, cicha próba odebrania prawa do broni czarnoprochowej, brak współpracy z MON w zakresie przygotowania projektu kodyfikacji szeroko rozumianego prawa obronnego i bezpieczeństwa, wreszcie brutalne pacyfikacje środowisk narodowych protestujących przeciwko marszom LGBT, m.in. w Rzeszowie. Ponadto prokuratura umorzyła właśnie dochodzenie w sprawie mężczyzny, który został zatrzymany na zeszłorocznym Marszu Niepodległości we Wrocławiu, tego z dzieckiem na rękach, który otrzymał liczne ciosy pałkami teleskopowymi od dwóch funkcjonariuszy. Nie wiem, czy ustalono już, czy doszło tam do przekroczenia uprawnień, czy nie ustalono tego jeszcze.

Gdzie były służby? Potrzebna jest poselska kontrola nad służbami również z naszej strony, ale konsekwentnie, pomimo silnego mandatu posłów Konfederacji, dostęp do Komisji do Spraw Służb Specjalnych jest dla nas ciągle zamknięty, co jest dużym błędem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi na tę interpelację. 3 lipca zwróciłem się w związku z tym z interwencją do wiceministra Wąsika o ujawnienie tych dokumentów, które ministerstwo przygotowuje, i do dzisiaj tych dokumentów nie dostałem. Pańscy ludzie na to nie reagują. Pan minister Wąsik obiecał mi ten projekt ustawy, obiecał mi potem jakąś notatkę na jej temat. Powiedział, że zaraz wróci z ustawą, po czym przyszedł z jakąś teczką, w której była nic niewnosząca notatka udająca odpowiedź na moją interpelację, na którą de facto nie odpowiadała, albo to, co tam było napisane, było nieprawdą. Czy państwu posłom tutaj, również z Prawa i Sprawiedliwości, to nie przeszkadza, że daliście się zdegradować do roli jakichś botów prezesa, którzy tylko naciskają guziki?

Dlaczego zatajacie prace legislacyjne przed Izbą legislacyjną? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Nie, nie, dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie pośle. Składam go na ręce przedstawiciela Prezydium Sejmu. Tak jest, my mamy swoje zastrzeżenia do ministra.

Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

Dziękuję, pani marszałek. panie premierze.

W takim razie w pierwszej kolejności - pan minister Mariusz Kamiński. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Minister jest zawsze w dyspozycji premiera i zawsze w dyspozycji parlamentu. Nie przesądzam, jaki będzie wynik głosowania. Zakładam, że może być pozytywny dla mnie, bo jak widać po dzisiejszych głosowaniach, jest stabilna większość w parlamencie, ale nie o to chodzi, proszę państwa.

To nie jest seans nienawiści dotyczący Mariusza Kamińskiego. Zgodnie z procedurą odpowiadam jako minister spraw wewnętrznych na zarzuty, które formułujecie wobec mnie.

Szanowni Państwo! Czytałem uważnie wniosek i jego uzasadnienie. Odnalazłem tam osiem zarzutów wobec mojej osoby, z czego tak naprawdę jeden dotyczy mnie jako ministra spraw wewnętrznych. Mówię o zarzutach, a nie faktach, tak naprawdę można powiedzieć: o insynuacjach, które tam są zawarte, często dementowanych, oczywistych. Słusznie pan poseł Sipiera wskazał na znamiennie sformułowania z tego wniosku, takie jak „z dużą dozą prawdopodobieństwa można domniemywać” To jest cytat z waszego uzasadnienia. W opinii publicznej panuje przekonanie” - takie są uzasadnienia insynuacji, które wobec mnie formułujecie. Ale odpowiem na zarzuty, bo tu pada jeden zasadniczy zarzut: brutalne tłumienie prawa, fundamentalnego dla obywateli prawa do swobodnego gromadzenia się i artykułowania swoich poglądów. Tak, uważam, że jest to prawo fundamentalne, prawo święte. Mówicie o brutalnym tłumieniu legalnych manifestacji. W uzasadnieniu znajduje się zdanie: „Tłumienie pokojowych i legalnych protestów obywateli przeciwko działaniom władzy przywodzi na myśl najczarniejsze karty historii PRL” To jest zdanie z waszego uzasadnienia.

Jakie? O jakie czarne karty w kontekście dławienia zgromadzeń publicznych chodzi?

Teraz ja, panie pośle, mówię. Bo nie mnie obrażacie. Obrażacie ofiary komunistycznych zbrodni, banalizując zło, banalizując zbrodnie, porównując happeningi jednego z kandydatów na prezydenta do zbrodni komunistycznych. A dodatkowo obrażacie 100 tys. polskich policjantów, porównując ich do komunistycznych zbrodniarzy.

Mówicie, że to były legalne protesty. Na mocy obowiązującego prawa, w związku z pandemią w całej Europie, we wszystkich niemalże państwach europejskich, wprowadzono zakazy gromadzenia się w celu zachowania dystansu społecznego, bo to jest najskuteczniejsza forma ograniczania pandemii. W niektórych państwach te zakazy istnieją do tej pory.

Półtora miesiąca. Dziękuję za poprawienie.

Teraz chciał stanąć na czele fali jakichś protestów. Czy naprawdę ktokolwiek jest w stanie uwierzyć, że mieliśmy do czynienia ze strajkiem przedsiębiorców? Mieliśmy do czynienia z politycznym happeningiem. Rozumiem, że też mam ograniczony czas, tak jak i państwo, więc rzeczywiście nie będę mógł tutaj szczegółowo i długo uzasadniać tych rzeczy. Ale zwracam państwa uwagę na słowa, jakie padają w parlamencie, na ich wagę, na to, że obrażacie ludzi, obrażacie pamięć o tych, którzy zginęli w PRL za wolność, za wolną Polskę i za chleb. To są rzeczy nieadekwatne.

Co robiły służby podległe MSW w ostatnich miesiącach? Robiły bardzo wiele i z tej trybuny moim obowiązkiem jest podziękowanie im... A Szumowski? ...niezasłanianie się nikim, ale podziękowanie. Opinia publiczna musi o tym wiedzieć. 10 mln wizyt związanych z kwarantanną zostało wykonanych przez funkcjonariuszy Policji. Już 10 mln, bo cały czas trwają te sprawdzania. I to nie chodzi tylko o to, żeby egzekwować ważne wymogi epidemiczne, ale chodzi również o to, żeby zapytać tego obywatela, który przestrzega przepisów i jest w domu: Tak, oskarżacie policjantów o to, że są bezmyślnym narzędziem w rękach nowego Kiszczaka, bo takie jest wasze myślenie.

W ciągu kilku dni powstały realne granice, żeby chronić naszych obywateli przed transmisją wirusa. Wszystkie te namioty, które widzieliście przed polskimi szpitalami, które były tymczasowymi izbami przyjęć, to były namioty strażackie, strażacy je rozstawiali. Strażacy wspierali służby na granicach, a jednocześnie wykonywali w skrajnie trudnych sytuacjach swoje obowiązki. Podtopienia, które miały miejsce, gwałtowne, zaskakujące wszystkich, w wielu regionach kraju. Czy ktoś został bez pomocy? Mówię o tym, czym się zajmował minister spraw wewnętrznych w ostatnich miesiącach i jemu podległe służby, za co chcę im z tego miejsca podziękować. Wojewodowie, którzy podlegają ministrowi spraw wewnętrznych, to rzeczywiści gospodarze w czasach bardzo trudnej walki z koronawirusem. 7 dni w tygodniu, w sobotę, w niedzielę również, odbywały się sztaby kryzysowe. Tak pracowały służby i administracja podległe ministrowi spraw wewnętrznych. I nikt im nie odbierze prawa do satysfakcji z tego, co zrobili, bo zrobili bardzo wiele dobrych rzeczy dla wszystkich obywateli. Mówicie o brutalności Policji, o tym, że doszło do rozruchów na miarę tego, co się działo w tragicznych sytuacjach w PRL. Spójrzcie, co się działo w tym czasie w innych państwach w Europie. Czy widzieliście te obrazki ze Stanów Zjednoczonych, te bójki z Policją, te napaści na policjantów, na sklepy, również na pomniki? Czy chcecie takich scen w Polsce? Nie, takich scen w Polsce nie będzie, nie będzie żadnych autonomicznych stref bez Policji, bo Policja to jest jeden z elementów funkcjonowania państwa. Każdy, kto rozumie, jak państwo funkcjonuje, wie, że służby podległe MSW muszą działać sprawnie.

Ja się tym nie przejmuję, mnie nie jesteście w stanie obrazić, jestem do tego przyzwyczajony, ale pośrednio atakujecie funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy służą wszystkim obywatelom. I to jest niedopuszczalne, to jest nieakceptowalne. I chcę z tego miejsca jeszcze raz bardzo gorąco podziękować wszystkim funkcjonariuszom służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i wszystkim urzędnikom podległym ministrowi. I na koniec jeszcze krótko odniosę się do tych tematów dnia.

No na Boga, służby specjalne, które mają kontrolować rozmowy międzynarodowe prezydenta czy premiera? No nie, szanowni państwo, tak nigdy nie było, nie jest i nie będzie. Są odpowiednie biura w Kancelarii Prezydenta, w kancelarii premiera, biura współpracy międzynarodowej, które na co dzień, codziennie organizują tego typu rzeczy, gdzie weryfikuje się pewne sprawy. Rzeczywiście ktoś zawiódł i wiemy, kto. Znamy z imienia i z nazwiska osobę, do której zwróciła się Kancelaria Prezydenta w przedstawicielstwie polskim w ONZ, którą poproszono o sprawdzenie wiarygodności tego telefonu i która potwierdziła, że to jest wiarygodne, że ta sytuacja jest wiarygodna. Będą wyciągnięte konsekwencje wobec konkretnej osoby, która zawiodła, która miała obowiązek jako pracownik polskiego przedstawicielstwa przy ONZ. Mówię to dla opinii publicznej, nie dlatego że minister spraw wewnętrznych czy koordynator służb specjalnych ma coś do rozmów międzynarodowych prowadzonych przez najważniejsze osoby w państwie. W sensie zabezpieczenia ich - tak, żeby nie były podsłuchane, ale nie w sensie kontaktowania się głów państw.

Jeżeli ktoś formułuje taki zarzut, to powinien przynajmniej sprawdzić podstawowe rzeczy. Naprawdę uważacie, że poinformowanie, że kobiety w ciąży, że osoby niepełnosprawne i seniorzy. mogą podchodzić bez kolejki do głosowania, jest nadużyciem? Nie, to jest w interesie tych osób, bo trzeba zachować środki bezpieczeństwa, a te osoby powinny być szczególnie chronione. RCB wielokrotnie tego typu alarmy wysyłało.

Tak że, kończąc swoje wystąpienie, jeszcze raz chcę podkreślić, że te emocje, które rozbudzacie, ta fala niechęci, nienawiści muszą mieć swój koniec. Mam nadzieję, że jednak troszkę te emocje opadną po wyborach. Następne wybory za 3 lata, więc pracujcie jako parlamentarzyści dla dobra państwa polskiego i obywateli. Śledztwo w tej sprawie trwa, szanowna pani, śledztwo w tej sprawie trwa z zawiadomienia ministra Szumowskiego. To są wasze insynuacje, wy przesądzacie o winie. Odpowie na to śledztwo, w którym funkcje wykonuje również Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pozwólcie, że też w ciągu kilku minut opowiem o osiągnięciach pana ministra, bo o tym należałoby mówić, i złożę podziękowania panu ministrowi za jego działanie w tym wyjątkowo trudnym czasie. Ten czas, czas COVID-19, jak słusznie ktoś tutaj zauważył, pandemii, której żaden kraj na świecie nie był w stanie przewidzieć, stawiał przed służbami specjalnymi i służbami mundurowymi wyjątkowe oczekiwania i wyjątkowe wymagania. I w tym czasie, kiedy z jednej strony służby mundurowe podległe panu ministrowi, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, musiały wypełniać swoje zadania dotychczasowe, a jednocześnie w dwójnasób spełniać oczekiwania społeczne co do nowych zadań nałożonych na nie, w tym samym czasie wykryto ogromne nieprawidłowości finansowe, a także takie, które są na ustach właściwie całego Europolu, związane z wykryciem gigantycznego przemytu narkotykowego, i to nie jednego, a trzech takich prób przemytu. Kiedy sobie uświadomiłem, jak wielka tkwi wartość we współpracy poszczególnych służb, którą zorganizował pan minister Kamiński, a jednocześnie jak bardzo brakowało tego wcześniej, to jednocześnie stało mi się bardzo przykro w związku z myślą o tym, jak wiele nieprawidłowości musiało umykać we wcześniejszych czasach, w czasach naszych poprzedników, przed tego typu kontrolami. Otóż przez ostatnie 6 miesięcy, 7 miesięcy, ale w czasie, który zahaczał o COVID-19, rozbite zostały gangi narkotykowe o międzynarodowym zasięgu i ocalone zostało życie i zdrowie dziesiątek tysięcy, może setek tysięcy młodych ludzi w całej Europie - nie tylko w Polsce, również w całej Europie. Dlatego premierzy innych państw dziękowali mi za te akcje, które w tak skuteczny sposób udaremniły import narkotyków na terytorium Unii Europejskiej. Te akcje stały się znane opinii publicznej. Zachęcam wszystkich do przyglądnięcia się temu, w jaki sposób od strony praktycznej współdziałały służby mundurowe i jakie były w związku z tym deficyty wcześniej. Kolejne obszary, na które chciałem zwrócić uwagę - o tych kolejnych obszarach mówił pan minister Kamiński, więc tylko krótko. Policja oprócz swoich normalnych działań przeprowadziła znakomite działania w obszarze kontroli kwarantann, ale także zaspokajania potrzeb, które można nazwać codziennymi potrzebami ludzi najbardziej tego wymagających, czyli wsparcia w zakresie dostarczenia żywności, pójścia po lekarstwa, pomocy w codziennych bytowych potrzebach. Tutaj policjanci byli zawsze dostępni i za to wszystkim policjantom chciałem podziękować. To ponad 9 mln, pan minister powiedział: 10 mln wizyt [[Oklaski]] - 10 mln wizyt. To też dzięki wam, drodzy policjanci, tę chorobę udało się ograniczyć w sposób skuteczny. Państwowa Straż Pożarna. Również pan minister o tym mówił. W czasie, kiedy pomagała przy podtopieniach, powodziach, pożarach wielkich, jednocześnie pełniła swoje obowiązki na różnych liniach frontu związanych właśnie z COVID-19.

To też jest wielka zasługa służb mundurowych pana ministra.

To było w lutym 2015 r., wtedy policjanci zostali zmuszeni, tak trzeba powiedzieć, przez dowództwo do strzelania do górników gumowymi kulami. Podobnie akcja „Widelec” - kilkuset kibiców aresztowanych, przetrzymywanych długo w aresztach. To pana śmieszy, panie pośle? Proszę się nie śmiać, proszę sięgnąć do zeznań tych kibiców. To wreszcie akcja AntyKomor, gdzie ośmiu antyterrorystów skierowaliście przeciwko jednemu studentowi bodaj o 6 rano, jeśli mnie pamięć nie myli, który założył stronę przeciwko ówczesnemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.

Tymczasem chcę podkreślić wyraźnie jedną cechę, bo to tutaj nie padło, pana ministra Kamińskiego. My równo traktujemy ludzi związanych z obozem rządzącym i z opozycją, ponieważ zatrzymywane są osoby również związane z obozem rządzącym, bo miecz prawa złemu tylko srogi, powinien być rzeczywiście zupełnie obiektywny i niepatrzący na to, kto skąd pochodzi. I dlatego właśnie pan minister Kamiński jest najlepszym ministrem w czasach III Rzeczypospolitej, który zapobiega korupcji, który w możliwie maksymalny sposób stara się odzyskać te zasoby, te pieniądze, które wpadły w ręce grup przestępczych. Chcecie dowody?

To są służby podległe panu ministrowi. Nie byłoby też tego sukcesu w ograniczeniu roli mafii VAT-owskiej, w ograniczeniu przestępstw podatkowych związanych z mafiami VAT-owskimi, tych przestępstw, w przypadku których tak udajecie, że patrzycie w ziemię w tym momencie, jak to mówię, ponieważ one was najbardziej bolą. Bo to jest kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie potwierdzonych przez Komisję Europejską. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. Dlatego, pani marszałek, Wysoka Izbo, pan minister Kamiński we wcześniejszych miesiącach, co do których przecież się wypowiadałem niedawno we wniosku składanym przez państwa, jak również, a może zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach, kiedy do normalnych zadań służb specjalnych, służb mundurowych doszły rozliczne wyzwania o charakterze hybrydowym związane z cyberbezpieczeństwem. W tym czasie nastąpiły różnego rodzaju aresztowania szpiegów, aresztowania i wydalenia osób, które w ewidentny sposób zagrażały bezpieczeństwu państwa, 48 osób, które miały zamiary terrorystyczne, a więc nasze grupy antyterrorystyczne świetnie zdały egzamin, ponieważ zidentyfikowały źródło ryzyka i dokonały wydalenia takich osób oraz niewpuszczenia dwudziestu kilku osób związanych z międzynarodowymi grupami terrorystycznymi. Nie widać tego, co dobrze działa. I zamiast podziękować panu ministrowi Kamińskiemu, kierujecie wobec niego doprawdy absurdalne zarzuty, zarzuty nijak się mające do rzeczywistości, bo oprócz normalnej roli, którą służby mundurowe i służby specjalne wypełniały w tym czasie, owszem, również roli związanej z pozyskiwaniem zasobów medycznych, środków medycznych, bo udajecie dzisiaj, że zapominacie o tych nagłówkach gazet sprzed 3 miesięcy: Skąd wziąć maseczki? Skąd wziąć respiratory? Skąd wziąć. Nieprawidłowości, które zostały wykryte w państwach Unii Europejskiej, przekraczają wielokrotnie te nieprawidłowości, które my sami wykryliśmy i co do których wyjaśnienia oczywiście dążymy. Ale za to, że pan minister Kamiński razem z panem ministrem Szumowskim wtedy szukali materiałów po całym świecie i ocalili życie dziesiątków milionów, dziesiątków tysięcy Polaków, tysięcy, dziesiątków tysięcy Polaków, należą im się słowa podziękowania, a nie absurdalne wnioski, które kierujecie. Dlatego podsumowując, szanowni państwo, mam krótki apel: Bądźcie opozycją Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a nie opozycją totalną, bo wnioskami, które kierujecie, i sformułowaniami. też haniebnymi sformułowaniami, które się znalazły w waszym wniosku, obrażacie majestat Rzeczypospolitej i wielu Polaków, którzy, jak powiedział tu słusznie pan minister Kamiński, pamiętają dobrze czasy PRL-u. Ale my i tak będziemy starali się cały czas modernizować służby mundurowe i usprawniać działanie służb państwa tak, żeby one służyły dobru wspólnemu, żeby one służyły także wam, bo państwo polskie to jest nasza przyszłość, to jest nasze dobro wspólne. Zamykam dyskusję. W jakim trybie, panie pośle?

Bardzo proszę. Jedno zdanie, panie pośle. Wysoka Izbo! Ja w trybie ad vocem. Oczywiście nie będę polemizował z panem premierem, to nie ta ranga, ale chciałam się odnieść w jednej sprawie do tego, co mówił pan minister Kamiński. Szanowny panie ministrze, specjalnie podkreślałem w czasie tego przemówienia, podobnie jak mój kolega, że jesteśmy pełni szacunku dla służb mundurowych, które wykonują swoją pracę znakomicie, tak jak wykonywały ją wcześniej, zanim pan był ministrem, i tak jak będą wykonywały tę pracę, jak pana dawno nie będzie. I to nie jest pana zasługa, że mamy dobrych policjantów. To niech się pan za nimi nie chowa i niech pan nam nie wciska, że my tak naprawdę poniżamy policjantów, bo jest dokładnie odwrotnie. Zamykam dyskusję. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.

Niech fakty przemówią. Coroczne badania opinii publicznej dotyczące oceny instytucji publicznych pokazują, jaki postęp zrobiliśmy jako państwo polskie, jako ministerstwo spraw wewnętrznych.

Dużo. W 2020 r., po kilku latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, po raz pierwszy w historii polska Policja została oceniona najwyżej przez obywateli, a poparcie dla niej i dobra ocena jej pracy sięga 80%.

Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (druki nr 454 i 475)

Wysoka Izbo!

Trefne maseczki, trefne testy, trefne karty wyborcze, niewidzialne respiratory i niewyobrażalna bezczynność resortu podległego Zbigniewowi Ziobrze, prokuratury w tych kwestiach właśnie. Czas spojrzeć w oczy i zapytać się, czy my przypadkiem nie żyjemy w trefnym państwie PiS. W państwie PiS afera goni aferę, tylko wszyscy mamy wrażenie, że nikt aferzystów w państwie PiS nie ściga. Wczoraj na posiedzeniu komisji sprawiedliwości nie dopuściliście nawet do zadawania pytań, dzisiaj wniosek jest raptem 5-minutowy. To są standardy jak w putinowskiej Rosji, jak w rosyjskiej Dumie, a nie w polskim Sejmie. Pani poseł... Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Oto najprostsze pytania, jakie możemy sformułować w odniesieniu do trzech ostatnich afer. Afera z maseczkami. Wiemy, kto na nim zarobił. Jakby był pan minister Ziobro, zadałabym mu pytanie, czy jest w stanie w jakikolwiek racjonalny sposób wyjaśnić, dlaczego nikt w tej sprawie nie siedzi jeszcze w areszcie. Państwo polskie zostało okradzione, [[Oklaski]] zrobiono naprawdę gruby wał, a winni chodzą na wolności. Kolejna sprawa: respiratory. Kontrolowane przez PiS Ministerstwo Zdrowia, zamiast dołączyć do unijnego przetargu, podpisało umowę z jakąś firemką, przelewając jej w kwietniu w klika godzin po podpisaniu kontraktu 160 mln zł. Miało być 1200 respiratorów, a jest drobny ułamek tej liczby. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Gdzie w państwie PiS jest prokuratura? To jest pytanie, które ciśnie się na usta. Udajecie najuczciwszych na świecie, a gdy trudne pytania zaczynają dotyczyć osób, które obecnie mają władzę, to nagle stajecie się osobami, które nic nie słyszały, które nic nie widziały. Myślałam, że jakkolwiek będziecie rządzić, to przynajmniej złodziei będziecie łapać. Wiecie co, nawet tego nie potraficie robić. Kolejna bulwersująca sprawa. Jacek Sasin i jego ludzie przygotowali wybory kopertowe, które przecież nie miały szans się odbyć. Wszyscy o tym wiedzieli. Epidemia, nic nie działało normalnie. Policja rozdawała mandaty wychodzącym z domu, dziesiątki tysięcy osób na kwarantannie. Straty dla państwa, dla każdego z nas, dla tych, którzy ciężko pracują i płacą podatki, sięgnęły, jak oszacowali dziennikarze, 70 mln zł. W czasie, gdy każdy publiczny grosz jest ważny, mógłby ratować miejsca pracy. Czy ktokolwiek miał postawione zarzuty w tej sprawie? Dlaczego na pytania prokuratury nie odpowiadał Jacek Sasin? Panie Ministrze! Listę pańskich błędów, pańskich zaniechań mogłabym wymieniać w nieskończoność, ale daliście mi tylko 5 minut. Powiem wprost: jest pan najgorszym ministrem sprawiedliwości w historii Polski.

To jest zwolnienie dyscyplinarne, które panu przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość przymykania oczu na afery z udziałem ludzi PiS. Przekazuje je panu w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość upolityczniania sądów. Przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość upolityczniania prokuratury i wykorzystywania jej do partyjnych celów. Przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość niszczenia europejskich standardów i wprowadzania tu, w Polsce, standardów znanych dotychczas tylko z Rosji i Białorusi. Przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość paraliżu Trybunału Konstytucyjnego.

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Pani poseł, proszę wrócić na miejsce i zachowywać się godnie. Bardzo proszę, panie pośle. Pani poseł, narusza pani powagę Sejmu. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, druku nr 454. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 116 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 7 lipca 2020 r. powyższy wniosek do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu zaopiniowania.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Przypominam, że zgodnie z art. 116 ust. 1a regulaminu Sejmu po wyczerpaniu listy mówców głos może zabrać tylko prezes Rady Ministrów oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Piotr Sak. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Generalnie wnioski tego typu są takimi swoistymi, specyficznymi aktami oskarżenia. Państwa wniosek, ten wyrób wnioskopodobny, nie powinien w ogóle trafić pod obrady Sejmu, tylko co najwyżej do konkursu im. Ignacego Krasickiego i Stanisława Lema, bo tyle w nim jest bajkopisarstwa i fantastyki, fantazji politycznej.

bo siła państwa argumentów jest porównywalna do zdolności bojowej plastikowych żołnierzyków. Wielu ministrów działa bardzo aktywnie i prężnie. Na tym tle wyróżnia się pan minister Zbigniew Ziobro, podobnie jak minister aktywów państwowych pan Jacek Sasin, minister zdrowia pan Łukasz Szumowski i minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Kamiński. Wszystkich potraktowaliście wnioskami o wotum nieufności. Co ich łączy? Są ludźmi ciężkiej, tytanicznej pracy, [[Oklaski]] a wy takich ludzi nie lubicie. Przecież lata waszych rządów to czas bylejakości, nastrojów niemożności, czas kranologii stosowanej, tej ciepłej wody w kranie, która jest synonimem waszego nieróbstwa i intelektualnego lenistwa. Wasza filozofia i doktryna to były ucieczka od rządzenia, zachowawczość działań, a wręcz nanibyzm i symulacja. Zamiast harować woleliście haratać w gałę. Stąd zagrożenie dla was ze strony naszego rządu, który jest bardzo pracowity i skuteczny. Nie potraficie urzeczywistniać zamierzeń i obietnic. Od 5 lat na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stoi pan minister Zbigniew Ziobro. Lista osiągnięć i sukcesów jest spora. Nie oczekuję oczywiście siłą rzeczy od państwa bezkrytycznych zachwytów, ale wasza ocena nijak ma się do rzeczywistości. Ostatnie lata to czas bezwzględnej walki, wojny z aferzystami. Odbierany jest majątek kartelom narkotykowym i mafiom, wprowadzano zbrodnię VAT-owską, zaostrzono kary dla pijanych kierowców, wprowadzono rejestr pedofilów. To jest podstawowa różnica. Wyciągnęliście ich samoloty, ich interesy, a my odbieramy im majątki, wsadzamy ich za kratki. Ministerstwo wspiera także osoby słabe i pokrzywdzone, z drugiej strony. Zbigniew Ziobro jest protektorem i strażnikiem interesów osób słabych i pokrzywdzonych. W ostatnich latach zwiększono ochronę ofiar przemocy domowej, uskuteczniono ściąganie alimentów, wprowadzono ogólnopolską sieć bezpłatnej pomocy prawnej. Wreszcie zatrzymano panoszenie się czyścicieli kamienic. Przerwano tę gehennę najemców. Skończono z nadużyciami komorników. Skończono z odbieraniem dzieci za biedę.

Zatem są podejmowane wielokierunkowe działania i dotyczą one także reformy wymiaru sprawiedliwości. Państwa autorytety zdiagnozowały kiedyś bardzo dobrze sytuację odnośnie do KRS-u. Andrzej Rzepliński w 2004 r. mówił: KRS to państwowy związek zawodowy konserwujący interesy źle służące polskiemu sądownictwu.

Szanowni Państwo! Fakty mówią przeciwko państwa wnioskowi i trwanie w złudzeniu, że jest inaczej, nie zmienia obiektywnego stanu rzeczy. O osiągnięciach, a lista jest coraz dłuższa, możemy mówić z zasłużoną satysfakcją (Dzwonek), bez naciąganych zachwytów. Nie chodzi o wystawianie laurki, ale chodzi o realizm oceny, którego wam niestety zabrakło. Szanowni Państwo!

W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Arkadiusz Myrcha.

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska pragnę jednoznacznie oświadczyć, że popieramy wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry. Popieramy wniosek o odwołanie najgorszego ministra sprawiedliwości. Popieramy wniosek o odwołanie ministra, który zbudował politykę resortu na kłamstwie, manipulacji i taniej propagandzie sukcesu, czego zresztą wczorajsze posiedzenie komisji sprawiedliwości było najlepszym potwierdzeniem. To nie jest kwestia naszej jakiejś subiektywnej politycznej oceny. Przeciwko panu ministrowi Ziobrze przemawiają fakty, statystyki, ale przede wszystkim ocena Polaków. To jest pierwszy minister sprawiedliwości w historii, który przez cały okres swojego urzędowania ma nieprzerwanie negatywne oceny działalności i prokuratury, i sądów. Proszę zerknąć do badań CBOS. Przecież to jest nokaut i wstyd, panie ministrze. Za chwilkę pewnie usłyszymy o innych badaniach CBOS, że teraz Polacy jakoby wyjątkowo bezpiecznie czuli się w Polsce. Ale, panie ministrze, odsyłam do lektury tego badania CBOS. Zauważy pan, że Polacy jako bezpieczne swoje miejsce zamieszkania oceniają w ok. 90% nieprzerwanie od 2008 r., więc proszę nie przypisywać sobie cudzych sukcesów. To jest wybitne osiągnięcie przede wszystkim policji, straży municypalnych, samorządowców, ale na pewno nie pana. Kolejny mit pana ministra Ziobry obalony. Ale chciałbym wrócić do wczorajszych obrad komisji sprawiedliwości. Pan minister Ziobro, pan minister Warchoł w sposób absolutnie haniebny zarzucali nam, jakobyśmy wspierali przestępców, jakobyśmy prowadzili bierną politykę w stosunku do sprawców przestępstw na tle seksualnym, pedofilii. To jest ustawa z kwietnia 2014 r., przyjęta przez Sejm. Ta ustawa ochroniła polskie dzieci przed zjawiskiem prostytucji. Ta ustawa wprost uderzała w zwyrodnialców, którzy promowali pornografię dziecięcą. Cała nowa regulacja art. 202 Kodeksu karnego. Tą ustawą policja uzyskała większe uprawnienia operacyjne w zwalczaniu przestępstw na tle seksualnym, w szczególności przeciwko małoletnim. I dzisiaj osiąga dzięki temu sukcesy, którymi pan się chwali. Wczoraj w komisji sprawiedliwości pan minister Ziobro i pan minister Warchoł ordynarnie okłamali Polaków. I gdyby mieli poczucie honoru, to za same te kłamstwa podaliby się po prostu do dymisji. Ale a propos pana ministra Warchoła.

Ale przypomnę: pan wtedy nie zasiadał w szeregach PiS, pan wtedy tutaj, w polskim Sejmie, był doradcą prawnym klubu Ruch Palikota. Ruch Palikota większość tych inicjatyw popierał. Tę nowelizację Kodeksu karnego z 2015 r., którą pan tak ostro krytykuje, pana ówczesny mocodawca Janusz Palikot poparł. To albo pan był miernym doradcą, albo pan jest dzisiaj zwykłym karierowiczem i hipokrytą.

Panie ministrze, zaskoczę pana. Pracowali wcześniej. Pracowali, zanim powstała Platforma i PiS, ba, do 2010 r. pracowało więźniów odpłatnie więcej niż teraz. Macie wynik 17 tys. Proszę sobie zerknąć - przed 2010 r. pracowało 20 tys. więźniów odpłatnie. Tylko taka różnica jest między nami, że my mu podziękowaliśmy, a wy go wzięliście na wicepremiera. Fundusz Sprawiedliwości - przez lata wspierał ofiary przestępstw, nikt nie miał do niego zarzutów. Pieniądze bez konkursów, miliony dla imperium o. Rydzyka, 25 mln na CBA, z których prawdopodobnie zakupiono program Pegasus, i dzisiaj słyszymy, że CBA inwigiluje dwa razy więcej osób niż ABW. Przecież to jest hańba. 5 lat ministra Ziobry to jest kompletna zapaść wymiaru sprawiedliwości i utrata zaufania do tego wymiaru przez Polaków. Polacy czekają rekordowo na wyroki sądowe. Sytuacja w prokuraturze jest jeszcze gorsza. Spraw długotrwałych jest w tej chwili ponad 21 tys., przy czym w 2015 r. ta liczba sięgała ledwie 6 tys. Państwo polskie płaci coraz więcej odszkodowań za przewlekłe postępowania. Dyscyplinarki dla prokuratorów, którzy mają odwagę być niezależni (Dzwonek) i mieć swoje zdanie. Tarcza, ochrona dla spraw, w których zaangażowani są ludzie PiS, czego symbolem na zawsze pozostanie całkowita bierność w sprawie tzw. łapówki prezesa Kaczyńskiego. Spada liczba spraw sądowych z udziałem prokuratura.

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Zawsze trudno przechodzi mi to przez usta: minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bo pan ma tyle wspólnego ze sprawiedliwością, co prezydent Andrzej Duda z konstytucją. Coś tam pan liznął, ale nic pan nie skumał. Ale przejdźmy do pana grzechów. Prokuratura. Prokuratura jest w pełni na pana usługach i prowadzi coraz więcej postępowań z powodów politycznych. Potraficie błyskawicznie wystosować akt oskarżenia wobec aktywistki za naklejki z tęczową Matką Boską. Potraficie ekspresowo wszczynać postępowanie wobec studentów z Uniwersytetu Śląskiego i przesłuchiwać ich tak, jakby byli mordercami. Potraficie wywlec z domu i wsadzić do aresztu bez jakiegokolwiek wyjaśnienia aktywistów za wieszanie plakatów, a do tej pory nie sformułowaliście aktu oskarżenia wobec Jarosława Kaczyńskiego za sprawę dwóch wież, a są na to taśmy. Drugi grzech, pedofilii. Wczoraj w komisji odwalił pan niezły teatr. Żadne pana machanie rękoma nie zmyje wstydu i blamażu pana i prezydenta Dudy, który ułaskawił pedofila.

Powiedzieliście, że to będzie obligatoryjnie. Czy zajął się pan 382 przypadkami księży pedofilów, o których na swojej konferencji w marcu 2019 r. mówił Episkopat Polski? 56% tych przypadków według Episkopatu Polski nigdy nie trafiło do prokuratury. Czy wysłał pan chociaż jeden wniosek do Watykanu o dostęp do dokumentacji o księżach pedofilach z Polski? Od grudnia macie taką możliwość, bo papież Franciszek zniósł tajemnicę papieską. Jedyne, co pan zrobił, to rozesłał pismo do regionalnych prokuratur, w których nakazał pan, aby organy państwa w relacjach z Kościołem opierały się na współdziałaniu i zrezygnowały z wykorzystywania swoich uprawnień. Pan, panie ministrze, cynicznie wykorzystuje kwestię pedofilii, bo chodzi tylko i wyłącznie o to, aby bronić biskupów, którzy kryją i przenoszą pedofilów w sutannach. Kolejny grzech, grzech Funduszu Sprawiedliwości. NIK po kontroli zmiażdżył ten fundusz. Wykazał, że fundusz nie zapewnia skutecznej pomocy ofiarom przestępstw. Zamiast pomagać ofiarom, pomagacie politykom Solidarnej Polski i organizacjom religijnym. Mało tego, zaczął pan ścigać organizacje pozarządowe, które zbuntowały się przeciw tym praktykom. Nasłał pan na organizacje pozarządowe Policję, która rekwirowała im komputery z danymi ofiar. Aktywistki zamęczaliście śledztwami po to, żeby później te śledztwa umorzyć, bo nic nie Ziobro, zamiast ścigać przestępców, ściga pan niewinne kobiety. Kolejny grzech, kadry. Wystawia pan, gdzie pan chce, swoich kolegów na eksponowanych stanowiskach w sądach w całym kraju, a tych, którzy są niezawiśli, stara się pan upodlić, zdegradować, przenosić i zastraszać. Oczywiście zadbał też pan o swoją żonę i swojego brata. Jest pan również głównym wykonawcą demontażu państwa prawa, szczucia na sędziów i nazywania ich uprzywilejowaną kastą. I zastanawiam się, czy podobne działania podejmie pan wobec uprzywilejowanej kasty klubu milionerów z PiS, którzy dorobili się milionów na szkodliwych transakcjach, szemranych interesach albo dorobili się w spółkach Skarbu Państwa. To za pana władzy również w instytucjach państwowych zatrudnienie dostają ludzie z fundamentalistycznej organizacji Ordo Iuris, która jawnie głosi poglądy odejścia od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To pana wiceminister Piebiak był głową układu, którego celem było szukanie haków na sędziów i prokuratorów. To pana człowiek Matecki prowadzi kilkadziesiąt stron, które mieszczą rasistowskie treści. Jarosław Kaczyński szukał kiedyś układu, ale ten układ urósł mu dzięki panu. W 2015 r. został pan ministrem sprawiedliwości, a swoimi ministrami mianował pana Dudę i panią Manowską. W 2018 r. rękoma niekonstytucyjnej KRS wysłał pan panią Manowską do Sądu Najwyższego, a w 2020 r. pani Manowska została kandydatką na pierwszą prezes Sądu Najwyższego i przypadkowo Andrzej Duda właśnie ją wybrał na to stanowisko. Mówiąc w skrócie, były wiceminister sprawiedliwości u Ziobry powołał byłą wiceministrę sprawiedliwości u Ziobry na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Panie Ministrze! Mój znajomy, kolega powiedział o panu kiedyś, że jest pan zerem. Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Dokonał pan rzeczy wręcz niewiarygodnej i w ciągu kilkunastu lat zjechał pan na poziom mniej niż zero.

Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Premierze! Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, który mam przyjemność reprezentować, nie widzi żadnych powodów, by dzisiaj bronić pana ministra Zbigniewa Ziobrę przed odwołaniem. Traktujemy jednak to wotum nieufności jako doskonałą okazję, by ocenić, przeanalizować pańską pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, albowiem, panie ministrze, jest pan najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości w naszym kraju w ciągu ostatnich 30 lat. W listopadzie minie już 5 lat, odkąd kieruje pan resortem. I w tym kontekście, panie ministrze, słabo prezentuje się pańska linia, która wczoraj została zaprezentowana w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, by odpowiadać na kłopotliwe pytania recenzowaniem poprzedników sprzed wielu, wielu lat. To naprawdę niezwykle słabo. 16 listopada 2015 r., obejmując urząd ministra sprawiedliwości, mówił pan, cytuję: Będziemy konsekwentnie zmierzać do tego, aby wymiar sprawiedliwości służył wszystkim ludziom, również tym słabym, niemającym grubych portfeli. Trzeba pamiętać, że sądy są dla ludzi, a nie ludzie dla sądów. Trzeba przyznać: niezwykle zacne i słuszne słowa. Wielu Polaków wtedy panu zawierzyło, licząc na naprawę systemu sprawiedliwości w Polsce. Jak się dzisiaj czują, najlepiej, myślę, świadczy pełna sala kolumnowa w styczniu tego roku przedstawicieli stowarzyszeń gromadzących ludzi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości, którzy tu przybyli, do Sejmu, na zaproszenie klubu Koalicji Polskiej, by wyżalić się z tego, jak są od wielu lat, kiedy zarządza pan resortem i prokuraturą, traktowani. Najlepiej świadczy o tym, jak rozgoryczeni są dzisiaj pańską postawą ludzie, osoba pana Marka Kubali, którego wniosek o rozpoznanie skargi nadzwyczajnej czeka na to rozpoznanie już ponad 830 dni. Przypomnijmy, skarga nadzwyczajna w założeniu miała pomagać obywatelom poszkodowanym przez wymiar sprawiedliwości. Pan Marek pyta, czy to są standardy działania pana ministra Ziobry. Za to wszyscy widzą zamiast tej poprawy, panie ministrze, Wysoka Izbo, parasol ochronny dla polityków Zjednoczonej Prawicy, dla ministrów Zjednoczonej Prawicy, dla liderów Zjednoczonej Prawicy, dla urzędników Zjednoczonej Prawicy. Wedle zapowiedzi Zbigniewa Ziobry wymiar sprawiedliwości miał być bardziej przyjazny dla obywateli. Dwa przykłady tylko.

Drugi przykład: wniosek o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela - wzrost opłaty o 400%. I tak dalej, i tak dalej, panie ministrze.

Wzrost ten, co istotne, szczególnie jest widoczny w sądach rejonowych. Wiele było deklaracji, panie ministrze, na temat skutecznego zwalczania przestępczości.

Było to o 48 tys. przestępstw więcej. Zapewniał pan o lepszej ochronie prawnej dzieci.

Naprawdę czas przestać uprawiać cyniczną politykę kosztem wymiaru sprawiedliwości, a wziąć się za jego naprawianie. Stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Krystian Kamiński. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Debatujemy teraz nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Argumenty, które słyszymy z obu stron, nie robią na mnie wrażenia. Przecież z góry wiadomo, że minister Ziobro nie ruszy nikogo z PiS-u, tak samo jak wcześniej było wiadomo, że minister z Platformy nie ruszy nikogo z Platformy. A przydałoby się. Przypomnę tutaj słowa z rozmowy pana Wojtunika z panią Bieńkowską o tym, kto według nich stoi za spaleniem budki przy rosyjskiej ambasadzie w czasie Marszu Niepodległości. Nie widzę ministra spraw wewnętrznych Platformy, a chciałbym go spytać, czy też jest zainteresowany dogłębnym śledztwem w tym temacie, bo powinien chyba być. Tak że tych państwa argumentów nie traktuję poważnie. Ale argument o braku zmian systemowych już uważam za słuszny. Dotychczasowe zmiany to tylko i wyłącznie walka o wpływy. Nie ma zgody na dalsze trwanie w tak niewydolnym systemie sądowniczym, w którym zwykli obywatele nie mają poczucia sprawiedliwości, a przedsiębiorcy na wyrok muszą czekać latami. Wszyscy widzimy, że potrzebna jest dziś gruntowna reforma systemowa, tak aby usprawnić nasze sądy, aby uczynić je przyjaznymi dla obywateli. Sądy powinny być przede wszystkim szybkie i sprawiedliwe. Sędziów trzeba uwolnić od wykonywania niemerytorycznych, biurokratycznych zadań. Właśnie dlatego jako Konfederacja proponujemy parametryzację sądów, przypisywanie asystentów na stałe do każdego sędziego, wprowadzenie zasady, że zostanie sędzią powinno być zwieńczeniem kariery prawniczej, a nie jej początkiem, w końcu uporządkowanie tematu współpracy sądów z biegłymi, który przysparza wiele problemów, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, a docelowo - proces w 1 miesiąc.

Walka pomiędzy waszymi kadrami naprawdę w tym przypadku jest kompletnie nieistotna, ponieważ żadna ze stron nic nie zrobiła, aby sprawy były rozstrzygane szybko i sprawiedliwie. Dziękuję, panie pośle.

Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję panu ministrowi, że zaszczycił nas swoją obecnością, bo na początku tej debaty go nie było, a wydawało mi się, że debata jest dosyć ważna.

Zacznę od tej strony. Wniosek o Trybunał Stanu dla pana Zbigniewa Ziobry. Nieobecni: Andrzej Biernat, Ewa Kopacz, Piotr Tomański, Leszek Blanik, Cezary Kucharski, Irena Tomaszak-Zesiuk, Marek Hok, Radosław Sikorski i Norbert Wojnarowski. Dziewięcioro członków Platformy Obywatelskiej zabrakło na sali, nie wypełniło swojego obowiązku poselskiego.

Ale to dzięki wam, przez was, przez nieobecność tej dziewiątki pan Zbigniew Ziobro przez ostatnie lata był ministrem i prokuratorem generalnym. To jest wasza sprawka, sobie podziękujcie. Szanowni Państwo! Trybunał Konstytucyjny - wasz. Sąd Najwyższy też już praktycznie przejęliście. Jeżeli macie wszystkie te mechanizmy, macie takiego genialnego ministra sprawiedliwości, dlaczego Platforma Obywatelska siedzi tutaj, a nie na Białołęce? Przecież szliście do wyborów, mówiąc, że wy tych wszystkich złodziei rozliczycie, że ich wszystkich powsadzacie. Gdzie oni siedzą?

Szanowni Państwo! Nieudolność, kolesiostwo, ustawy pisane na kolanie - to jest wizytówka Zbigniewa Ziobry, dlatego będziemy. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę o zabranie głosu ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobrę. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Mianowicie te fakty to działanie prokuratury, tak bardzo krytykowane i atakowane przez moich przedmówców, w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w okresie pandemii, w związku ze sprawą maseczek, respiratorów.

A jak było za czasów przedstawicieli totalnej opozycji, która chce wyznaczać szczególne standardy działania prokuratury i krytykuje rzetelnie i uczciwie wywiązujących się ze swoich zadań śledczych? Otóż przypomnę państwu, bo pamięć to rzecz krótka i warto ją odświeżać. Otóż materiał dowodowy został zebrany w tej sprawie przez organa ścigania w okresie rządów Platformy w 2014 r.

Czy widzicie różnicę? Mieliście jakieś problemy ze ściganiem swoich nie tylko w tej sprawie. To popatrzmy na inny fakt. Sprawa Amber Gold. Od momentu, kiedy wpłynęło pierwsze zawiadomienie do prokuratury za waszych czasów, do wszczęcia śledztwa minęły przeszło 2 lata, przeszło 600 dni, a w tym czasie ludziom rozkradano majątek i dorobek całego życia. W tym czasie działy się ludzkie dramaty, w tym czasie niektórzy ludzie odbierali sobie życie. Co zrobiliście dla tych ludzi? Tutaj macie problem, że my wszczęliśmy następnego dnia. Czego wy chcecie? Macie odrobinę honoru? To nie jest rzeka, to nie jest morze, to jest ocean hipokryzji, zakłamania i cynizmu. Potraficie wszędzie kłamać, również na temat danych statystycznych, o których pan poseł mówił, do których się za chwilę odniosę. Ile czasu minęło od wszczęcia śledztwa w tej sprawie? 3 lata, prawie 1000 dni.

Jest sprawa pana senatora Gawłowskiego.

Tymczasem to przecież niezawisłe sądy stosowały tymczasowe aresztowanie i to utrzymywały, uznając, ze zebrany materiał dowodowy przez prokuraturę, którą kieruję, jest merytoryczny, zasadny i w najwyższym stopniu wskazuje na fakt czy uprawdopodabnia fakt popełnienia przestępstw korupcyjnych, prania pieniędzy i innych czynów przestępczych, jakie zostały zarzucone jemu i osobom z nim współdziałającym. Ale rozumiem, to wasz przyjaciel polityczny i kolega, którego, idąc w zaparte, broniliście nawet wtedy, kiedy niezawisłe sądy, tak bardzo przez was bronione i pokazywane jako przykład, wskazywały, że są bardzo mocne przesłanki, by sądzić, że doszło tutaj do poważnych przestępstw kryminalnych. A więc jeśli porównujecie szybkość prowadzenia postępowań za naszych czasów i za waszych czasów, to byście się wstydzili, jeśli chcecie nas (Dzwonek) krytykować bez odwoływania się do własnych doświadczeń. Nie, nie, bardzo proszę. Myślę, że dobrą puentą tego wystąpienia jest to, co przed chwilą powiedziałem, że skala zarzutów, które państwo tutaj podnosicie, jest niczym innym jak oceanem zakłamania. Otóż zapomniał pan dodać, że w okresie, kiedy państwo odpowiadaliście za wymiar sprawiedliwości, za bezpieczeństwo Polaków, Polacy w 66% wskazywali, że czują się bezpiecznie, a dzisiaj w 89%. Otóż ta różnica jest. Ona z czegoś wynika. Zakłamuje pan dane CBOS-u, mówiąc, że rzekomo za waszych czasów było duże zaufanie do sądownictwa, ono jakoby spadło. Teraz jest, można powiedzieć, odwrotnie. Pierwszy raz w historii, nawiasem mówiąc, nastąpił wzrost zaufania, był większy poziom zaufania do działań prokuratury niż poziom nieufności wtedy, kiedy pierwszy raz zostałem prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. To są twarde dane, badania CBOS-u. Niech pan sprawdzi, niech się pan przygotuje do wystąpienia, a potem niech pan się do nich odwołuje. Otóż mógłbym przywoływać mnóstwo danych, które całkowicie zaprzeczają temu fałszywemu obrazowi, który państwo tutaj malujecie, zakłamanemu, jeżeli chodzi o działania prokuratury, bo w każdym, można powiedzieć, przypadku, jeśli popatrzymy na zwalczanie mafijnej zorganizowanej przestępczości, jeżeli popatrzymy na zwalczanie przestępczości gospodarczej, jeżeli popatrzymy na klasyczną kryminalną przestępczość, to widzimy ogromną różnicę w stosunku do czasów poprzednich. Każdy może do nich sięgnąć, skoro czasu już nie mam. Odwołam się tylko do jednej sprawy, która wymaga jednak reakcji.

Bo wy żeście nic albo niewiele robili, by ścigać realnie pedofilów, by zaostrzać w stosunku do nich Kodeks karny. Możecie zobaczyć statystyki różnych inicjatyw ustawodawczych, które żeście blokowali, kiedy proponowaliśmy skuteczną walkę z pedofilią. Ale to, co jest najbardziej uderzające. Nie wprowadziliście też ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, którą myśmy wprowadzili, bo wy lubicie dużo mówić, ale nie wynika z tego realne działanie. Ale to, co zrobiliście tym kobietom pokrzywdzonym w tej sprawie, to, jak instrumentalnie, cynicznie żeście je wykorzystali, to jest naprawdę szczyt, który przekracza nawet moje wyobrażenia o tym, do czego jesteście zdolni. To właśnie te dzielne kobiety, kiedy doszło do popełnienia przestępstwa przez ich partnera, ojca, człowieka bardzo mocno pogrążonego w chorobie alkoholowej, zainicjowały postępowanie karne, to one doprowadziły do tego. że prokuratura prowadziła w tej sprawie śledztwo, to one doprowadziły do skutecznego oskarżenia tego sprawcy za okrutne czyny, których się dopuścił.

Ale potem to również one, kiedy ten sprawca wyszedł z zakładu karnego, kiedy dowiedziały się, że wyleczył się, że poddał się terapii, kiedy nawiązały z nim relację i trwało to przez dobrych kilka lat, zwróciły się do pana prezydenta, żeby skorzystał z prawa łaski - nie w stosunku do morderców, bandytów, których ułaskawiał wielokrotnie częściej, trzy razy częściej pan prezydent Komorowski, a jeszcze wielokrotnie częściej pan prezydent Kwaśniewski, np. zabójców, wbrew zresztą opiniom sądów i prokuratorów - żeby, powtarzam, pan prezydent skorzystał z prawa łaski wobec sprawcy, który odbył całą karę, od dnia pierwszego do dnia ostatniego, który odbył tak samo większość środka karnego zakazującego mu kontaktu z tymi kobietami, bo przecież ten środek został orzeczony w ich interesie, wyłącznie w ich interesie, na okres 6 lat, a minęło 5 lat.

Mianowicie powiedziały: Jesteśmy bardzo wdzięczne panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że dał nam szansę na normalne i spokojne życie. Wszystko wskazywało, że tak się stanie, aż do ostatniego tygodnia. Nie spodziewałyśmy się, że nasze prawo do godnego życia i oderwania się od dramatycznej i smutnej przeszłości zostanie tak bezwzględnie złamane i wykorzystane do brudnej kampanii politycznej. Publikacja dziennika „Fakt” spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Nikt nas przed nią o nic nie pytał - rzetelność, prawda? - nie uprzedzał, nikt nie próbował poznać naszego zdania. Nikt nie zastanawiał się, ile już w życiu wycierpiałyśmy.

Co oznacza bycie ofiarą tego rodzaju przestępstwa? i rozpocząć nowe życie.

Bardzo proszę panią o zachowanie spokoju.

Dziennikarze - dodają te panie - i politycy, politycy, również panie posłanki, nie mają prawa tak działać, nie mają prawa w taki sposób niszczyć psychiki zwykłych ludzi. Fundusz Sprawiedliwości. Mógłbym podać tu wiele danych Funduszu Sprawiedliwości, ale to jest strzał w kolano, pani poseł. Fundusz Sprawiedliwości działał za waszych rządów i wtedy jego rolą było pomóc tym kobietom.

Czy rządziła wtedy Zjednoczona Prawica, czy przypadkiem Platforma i PSL? Dlaczego nie pomogliście tym kobietom? Gdzie byliście? Gdzie wasza empatia? Ja wam powiem. Bo pieniądze szły.

Tak bardzo przejmujecie się ofiarami przestępstw.

Widzicie różnicę?

chociaż jeden przykład upolitycznienia sędziego, sądu lub jakiegoś wyroku. Nie proszę nawet o pięć. Podajcie jeden przykład. Nie potraficie. Tyle w temacie upolityczniania wyroków.

Tam dokonano weryfikacji i lustracji sędziów i prokuratorów po czasach komunistycznych. Wiecie, ilu pozostawiono? I to, myślę, jest właściwa liczba. Zostawiono wtedy w NRD ok. 30% prokuratorów i ok. 30% sędziów.

Chcemy naprawić wymiar sprawiedliwości. Aby obnażyć jego słabości, najlepiej przytoczyć kilka spraw.

Otóż, śmiejecie się z tego, ale nic mu się nie stało. Inny przykład.

Gdy inna osoba zapłaciła tę grzywnę, sąd ukarał też tę inną osobę za ten niedopuszczalny czyn. To jest prawo, które jest silne dla słabych.

Dlatego pan minister Ziobro podejmuje próby, które w pełni popieram, zaostrzenia Kodeksu karnego, zaostrzenia kar dla najgorszych przestępców, za najgorsze przestępstwa, z premedytacją. W tym kierunku trzeba iść, drodzy państwo.

Praworządność jest wtedy - bo lubicie się na to słowo powoływać - praworządność, Wysoka Izbo, jest wtedy, kiedy prawo chroni obywateli i słabszych obywateli chroni bardziej niż silniejszych obywateli, bardziej niż oszustów. Bo rzeczywiście wystarczy, dla potwierdzenia skuteczności działania prokuratury, przytoczyć kilka przykładów. Ten, o którym mówił pan minister Ziobro, Amber Gold, ponad 2 lata czekał. Inne przykłady - ponad 3 lata, w czasach Platformy Obywatelskiej. Teraz GetBack - inna afera, tak, wielka, bardzo niedobra afera. Tu macie 2 lata, a tutaj macie 2 miesiące. Ciężko wam się tego słucha, prawda? Szanowni Państwo!

Ale niektóre z nich rzeczywiście (Dzwonek) ośmieszają wymiar sprawiedliwości do tego stopnia, że pewnie należałoby opuścić na nie kurtynę milczenia. Ja w związku z tym przytoczę tylko kilka.

Kopiował je tak, że nawet skopiował dane osobowe, dane adresowe, w niewłaściwy sposób. Jak nazwalibyście takie zachowanie?

Ślad na duszy tej biednej kobiety, a tutaj mniej niż dwukrotne wynagrodzenie tego sędziego. A sędzia Milewski w waszych czasach? Sędzia na posyłki? To jest wymiar sprawiedliwości, który chcecie budować? Odwołajcie się do spraw, które dobrze znamy z niedawnej przeszłości, z czasów, kiedy prokuratura była oddzielona od ministra sprawiedliwości, prokurator generalny.

Takich sytuacji są dziesiątki, jeśli nie setki, i dotyczą one bardzo dużych spraw. Czy to jest wymiar sprawiedliwości, którego wy chcecie? Wysoka Izbo!

Tej reformy, którą. pan minister sprawiedliwości, pan minister Ziobro z determinacją cały czas stara się urzeczywistnić. Przerywała pani panu ministrowi, przerywa pani panu premierowi. Bardzo proszę, miała pani czas na wystąpienie, obrażała pani Wysoką Izbę, nikt pani nie przerywał, więc bardzo proszę zachować się spokojnie i godnie, [[Oklaski]] jak przystało parlamentarzyście tej Izby. Chcę wspomnieć o jeszcze jednej sferze, gdzie współpracuję blisko z panem ministrem Ziobrą i jestem przekonany, że bez tej determinacji, jaką wykazuje prokuratura, nie byłoby pewnych fundamentalnych sukcesów, sukcesów związanych z walką z przestępczością gospodarczą, z mafiami VAT-owskimi.

Kilkukrotnie większa kwota świadcząca o determinacji, skuteczności, efektywności i profesjonalizmie działania prokuratury i organów ścigania. To są środki, drodzy rodacy, Wysoka Izbo, które przeznaczamy właśnie na cele społeczne, na cele rozwojowe, na infrastrukturę, a te środki wcześniej lądowały w kieszeniach przestępców.

Wysoka Izbo! Proszę o odrzucenie wniosku o wotum nieufności wobec pana ministra Ziobry, ponieważ pan minister stara się naprawiać jedne z najtrudniejszych obszarów życia publicznego, gospodarczego i społecznego jednocześnie, które stanowią niechlubną spuściznę III Rzeczypospolitej.

Od naprawy tych instytucji zależy również przyszłość polskiej gospodarki i przyszłość naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo, panie premierze. Pan poseł Arkadiusz Myrcha prosił o wystąpienie w trybie sprostowania. Ale, panie pośle, 1 minuta, dobrze?

Mówiłem wprost, badanie z 2019 r., na str. 2 jest wyraźna grafika, odpowiedź na pytanie, czy Polacy czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Odsyłam. Jeśli pan nie wie, to proszę zwolnić swoich zastępców. Jeżeli chodzi zaś o ocenę prokuratury, cieszę się, że pan o tym wspomniał, bo mogę się pochwalić. 2008 r. - 44 pozytywnie, 28 negatywnie, 2010 r. - też przeważały oceny pozytywne, 2011 r. - również przeważały oceny pozytywne. A jeżeli chodzi o zajęte kwoty, zabezpieczone kwoty przez prokuraturę, odsyłam do raportu NIK.

Na 1 miesiąc. Dziękuję, panie pośle. No dobrze. Minuta, panie ministrze. Wysoka Izbo! Skoro rozmawiamy o badaniach, pan poseł podał wynik jednego badania, tylko tak jakoś umknęło panu posłowi podanie wyników badań w zakresie.

Pan poseł Myrcha podaje wyniki badań, [[Gwar na sali, oklaski]] tylko zapomina o tym, że badanie dotyczy wielu spraw.

W tym badaniu właśnie jest 86%. z tego powodu, że opinia publiczna i Wysoka Izba nie ma pewnej informacji, którą z przyjemnością przytoczę: zagrożenie bycia pokrzywdzonym przestępstwem.

Wznawiam obrady. A więc bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Bardzo proszę.

Zieloni złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: pierwsze, drugie i trzecie czytania: - poselskiego projektu ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druki nr 278 i 278-A, - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druk nr 304. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym rozpatrzenia projektu ustawy zawartego w drukach nr 278 i 278-A. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym rozpatrzenia projektu ustawy zawartego w druku nr 304. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść ręką i nacisnąć przycisk.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Przypominam, ze zgodnie z art. 159 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, zechce nacisnąć przycisk.

Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przypominam, że zgodnie z art. 159 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zechce nacisnąć przycisk.

Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 15 lipca br.